Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że pan poseł Waldemar Olejniczak złożył ślubowanie poselskie. Rada Ministrów przedłożyła pilny projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, druk nr 56. W związku z tym, na podstawie art. 73 ust. 1 regulaminu Sejmu, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Grupa posłów przedłożyła projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz Prawo celne, druk nr 51. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący pierwsze czytanie tego projektu. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych przedłożyła sprawozdanie o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, druk nr 55. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o projektach ustaw: - o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, - o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Sprawozdania to odpowiednio druki nr 54 i 52. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań. Proponuję, aby w tych przypadkach Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, przedłożyło wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych, druk nr 53. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego wniosku. Prezydium Sejmu proponuje, aby Sejm wysłuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła w dyskusji nad sprawozdaniem w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydium Sejmu proponuje, aby w dyskusjach nad pozostałymi punktami porządku dziennego Sejm wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycje przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Informuję, że Konwent Seniorów jednomyślnie zaopiniował propozycję rozpatrzenia na bieżącym posiedzeniu informacji w sprawie „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”, o której przedstawienie wnosił Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Punkty porządku dziennego bieżącego posiedzenia będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów. Z wnioskami formalnymi zgłosili się posłowie. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam wielką prośbę do pani marszałek, ponieważ klub Koalicji Obywatelskiej 3 grudnia zgłosił projekt uchwały w sprawie wyrażenia uznania dla laureatki Nagrody Nobla Olgi Tokarczuk. Rozumiem, pani marszałek, że na posiedzeniu Prezydium zapadły ustalenia, że ta uchwała będzie podjęta podczas tego posiedzenia, ale w przyszłym tygodniu. Sejm Rzeczypospolitej będzie ostatnią instytucją, ale ważne, żeby to się stało. Dlatego bardzo proszę panią marszałek, żeby zobligować przewodniczącego komisji kultury do tego, by ta uchwała była przeprocedowana na tym posiedzeniu Sejmu. To jest sprawa zbyt ważna, tu nie może być żadnej polityki. Dziękuję, panie pośle. W pełni się zgadzam, że Komisja Kultury i Środków Przekazu powinna jak najszybciej przygotować projekt tej uchwały, tak żeby on był ponad podziałami, żeby mógł być przyjęty przez całą Izbę. Bardzo proszę. Minuta, panie pośle.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Na podstawie art. 184 ust. 3 pkt 1 regulaminu Sejmu chciałbym zgłosić wniosek formalny o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów - Konwentu, który jest niezbędny, aby można było skutecznie uzupełnić porządek obrad o punkt, który zgodnie z regulaminem Sejmu zgłosił już klub Koalicja Polska, dotyczący informacji o działaniach zmierzających do przeciwdziałania rozprzestrzeniającemu się wirusowi ASF, który niszczy polskich producentów trzody chlewnej.

Panie pośle, chciałam tylko poinformować, że nie zwołam Konwentu Seniorów, ponieważ przed chwileczką odbyło się posiedzenie Konwentu Seniorów i ta sprawa była omawiana i w Prezydium Sejmu, i w Konwencie. Ten wniosek, który jest bardzo ważnym wnioskiem, kierujemy do komisji rolnictwa. Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Michał Szczerba, Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Składam wniosek formalny o przerwanie posiedzenia i zwołanie Konwentu Seniorów w celu rozszerzenia porządku obrad o punkt dotyczący informacji ministra sprawiedliwości na temat nieprawidłowości w realizacji programu „Praca dla więźniów” i nadzorze nad nim. Szanowni Państwo! Mamy do czynienia z wynikami, które są bezprecedensowe. NIK skierował 16 zawiadomień do prokuratury w sprawie realizacji tego programu.

Szanowni Państwo!

Dziękuję panu bardzo. 1 minuta, pani poseł. Wysoka Izbo!

Wielkopolska to 40% hodowli trzody chlewnej w Polsce.

Owszem, ale w tym czasie zabito 50 tys. świń, a 100 tys. stad zniknęło z Polski.

Pani poseł, to jest wniosek, który już wcześniej padł, i wyjaśniałam, jaka będzie procedura. Sprawa jest ważna i trafi do komisji rolnictwa, pani poseł. 1 minuta, panie pośle. Wysoka Izbo! Zgodnie z pismem, które złożyliśmy do pani marszałek, klub parlamentarny Lewicy zwraca się na podstawie regulaminu Sejmu o rozszerzenie porządku obrad o informację pana premiera dotyczącą afery związanej z prezesem Najwyższej Izby Kontroli panem Marianem Banasiem. W dniu dzisiejszym pan minister, wicepremier Jacek Sasin powiedział, że to opozycja bierze odpowiedzialność za to, że prezes NIK dalej pełni swoją funkcję. To skandal i hańba, że jako parlamentarzyści pozwalamy na to, żeby pan minister, pan prezes Najwyższej Izby Kontroli dalej pełnił tę funkcję. Pan premier powinien wytłumaczyć się z tego, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość dopuściło do tej nominacji i dlaczego służby specjalne zawiodły przy sprawdzaniu pana Mariana Banasia, a przede wszystkim z tego, dlaczego dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość - ręka w rękę z panem prezesem NIK - chce go utrzymać, hańbiąc Najwyższą Izbę Kontroli.

Ostatni wniosek formalny, pan poseł Romuald Ajchler, Lewica. Wysoka Izbo!

Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji: - Finansów Publicznych wspólnie z Komisją Gospodarki i Rozwoju - godz. 11, - Edukacji, Nauki i Młodzieży - godz. 13, - Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych - godz. 15.30, - Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - godz. 16, - Finansów Publicznych - 15 minut po zakończeniu ewentualnych głosowań, o godz. 11.30.

Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 1. porządku dziennego: Pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (druk nr 56) Proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów pana Tomasza Robaczyńskiego o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019. W przypadku tego projektu Rada Ministrów podjęła decyzję o szybkiej ścieżce legislacyjnej wynikającej z art. 123 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W projekcie ustawy zawarto przepisy, zgodnie z którymi w roku 2019 proponuje się przekazanie dodatkowych środków Narodowemu Funduszowi Zdrowia z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu zapasowego do wysokości 2 mld zł na pokrycie zwiększonych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej. W roku bieżącym dokonano już zaangażowania znacznej części środków funduszu zapasowego NFZ na pokrycie zwiększonych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej o wysokości 2,2 mld zł.

Aby ta operacja mogła zostać przeprowadzona, przekazanie tych środków musi nastąpić do końca roku 2019, co oznacza, że ustawa musi wejść w życie jeszcze w tym roku.

Przepis ten pozwoli na realizację w większym zakresie ustawowych zadań funduszu polegających na pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakup na ich potrzeby niezbędnych towarów i usług. Kolejne regulacje dotyczą możliwości wydatkowania środków na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, zakupu nowych karetek dla ratownictwa medycznego oraz wydatków majątkowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przepisy te wprowadzają wyjątek od zasady wyrażonej w art. 181 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który przewiduje, że niezrealizowane kwoty wydatków budżetu państwa wygasają z upływem roku budżetowego. Zgodnie z art. 109 ust. 4 ustawy o finansach publicznych rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy. W związku z tym celem projektowanych rozwiązań jest umożliwienie wydatkowania środków ujętych w budżecie państwa na realizację ww. zadań do końca kwietnia 2020 r. Środki te będą traktowane w podobny sposób jak wydatki niewygasające przewidziane w ustawie o finansach publicznych. Mając na uwadze powyższe oraz konieczność wypełnienia dyspozycji art. 181 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, czyli konieczność przekazania środków do końca roku na wyodrębniony rachunek wydatków centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, istnieje uzasadnienie procedowania przedmiotowego projektu w trybie pilnym. Mówiłem o tym, że uzasadnieniem tego jest także fakt konieczności przekazania środków - czy też umożliwienia przekazania środków - na fundusz zapasowy NFZ oraz Fundusz Wsparcia Policji do końca bieżącego roku. Mając na względzie powyższe, zwracam się do Wysokiej Izby z prośbą o przyjęcie tego projektu ustawy. Dziękuję bardzo. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jako pierwsza głos zabierze pani poseł Gabriela Masłowska, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 z druku nr 56 ma na celu stworzenie podstawy prawnej do przekazania jeszcze w tym roku dodatkowych środków z budżetu - w kwocie do 2 mld zł - na powiększenie funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na świadczenia opieki zdrowotnej oraz dodatkowych środków - w kwocie do 1 mld zł - na Fundusz Wsparcia Policji, fundusz centralny. Jednocześnie drugim ważnym przesłaniem, zadaniem tego projektu, pilnego projektu rządowego, jest uczynienie pewnych wydatków niewygasającymi, co umożliwi ich wykorzystanie po zakończeniu roku budżetowego, w terminie do 30 kwietnia 2020 r. Środki te będą przekazane z budżetu państwa, a konkretnie z wydatków zablokowanych na podstawie ustawy o finansach publicznych, bez uszczerbku dla zadań zaplanowanych dla tych wydatków, ponieważ będą one pochodzić z poczynionych oszczędności budżetowych, co jest rzeczą naturalną przy realizacji budżetu. Wykorzystanie środków zarówno przez NFZ, jak i centralny fundusz wsparcia nastąpi po uzyskaniu zgody ministra ds. finansów publicznych, właściwych ministrów zdrowia oraz spraw wewnętrznych i administracji.

Przedłożony projekt zasługuje na poparcie z tego względu, że dzięki oszczędnościom poczynionym przy realizacji budżetu umożliwia on zwiększenie środków na wykonanie takich zadań, w zakresie których są ogromne potrzeby, m.in. jeśli chodzi o dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej, poprawę ich jakości, a także kwestię bezpieczeństwa państwa. Projekt, nad którym debatujemy, jednocześnie świadczy o skutecznej, efektywnej polityce finansowej, fiskalnej państwa, budżetowej państwa, która pozwala na dostosowywanie możliwości budżetowych bez uszczerbku dla finansów publicznych do lepszego, bardziej racjonalnego wykonywania zadań przez niektóre resorty. M.in. dzięki tym zmianom będą zwiększone środki na inwestycje, modernizacje, remonty, jeśli chodzi o jednostki Policji, a także na zwiększone koszty utrzymania niektórych jednostek Policji, na zakup różnych towarów i usług, czyli na wydatki majątkowe. Jesteśmy przekonani, że projekt jest uzasadniony, umożliwi znaczną poprawę stopnia realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia, a także w zakresie bezpieczeństwa. Uważamy, że trzeba pilnie debatować nad tym projektem, tak żeby móc efektywnie, zgodnie z przedłożeniem, te środki wykorzystać. Dlatego Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość jest za szybkim procedowaniem nad tym projektem, który popieramy. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł Izabela Leszczyna, klub Koalicja Obywatelska. Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! To kolejny odcinek w piątym roku serialu pt. „Psucie państwa, psucie prawa i psucie finansów publicznych przez PiS” Psucie finansów publicznych - ponieważ tą ustawą wypychacie kolejne środki poza limit wydatków ze stabilizującej reguły wydatkowej, panie ministrze, [[Oklaski]] i wie pan doskonale, że tak naprawdę chodzi o to i tylko o to.

Przekroczyliście limit ze stabilizującej reguły wydatkowej i w gruncie rzeczy za to samo moglibyście postawić Mariana Banasia przed Trybunałem Stanu. Ale złapaliście się tą lewą ręką za prawe ucho i dociskacie Fundusz Solidarnościowy, bo boicie się, że Banaś przed Trybunałem Stanu pociągnie całą Radę Ministrów, bo cała Rada Ministrów przecież zgodziła się na wydanie 15 mld zł więcej, niż prawo polskie rządowi pozwala. Gdybyśmy chcieli poszukać paraleli ze światem ludzi zwyczajnych, którzy nie muszą się znać na zasadach budżetowych, funkcjach finansów publicznych, ale rozumieją doskonale, że stabilność finansów publicznych to jest gwarant tego, że każdy polski emeryt każdego miesiąca dostanie swoją emeryturę. I teraz wy tę stabilność psujecie i zachowujecie się tak jak człowiek, taki hulaka, lekkoduch, utracjusz - który wyda wszystko, co ma, zaciągnie bezpieczne kredyty, ale wciąż mu mało. No to bierze chwilówki i wchodzi w ten sposób w spiralę zadłużenia. To robicie Polakom.

Nie przyjmujemy Misiewiczów. Wie pan doskonale, że nie robiliśmy żadnej czystki w Ministerstwie Finansów i nie sprowadziliśmy ludzi, którzy założyli tam mafię VAT-owską. Nie wiem, czy to na pana piętrze oni siedzą, czy na innym. Więc współczuję panu, panie ministrze, bo pan tę żabę będzie w kolejnych latach prawdopodobnie z nami i z wszystkimi Polakami zjadał. Otóż na trzy sposoby PiS psuje ustawę o finansach publicznych i obchodzi ustawę o finansach publicznych tą ustawą. Po pierwsze, tak jak powiedziałam, łamie stabilizującą regułę wydatkową.

Dokładnie to robicie tą ustawą i tymi poprzednimi, które przyjmowaliśmy i które dzisiaj są w Senacie. Ta ustawa to kolejne 3 mld zł, a może nawet 4, którymi przekroczylibyście ten limit, więc wyjmujecie je z tego limitu, za który odpowiada minister finansów, wkładacie do NFZ-u.

Te 2 mld nic wam nie dadzą. Ubieracie to w Narodowy Fundusz Zdrowia, dlatego nie możemy zagłosować przeciwko, bo przecież wasza propaganda wyjdzie na ulicę i powie: „no chcieliśmy dać do NFZ-u, ale zła opozycja nie chce”, co jest oczywistą nieprawdą. Drugi sposób, w jaki łamiecie prawo w tej ustawie, to tworzycie rezerwę, która zgodnie z ustawą o finansach publicznych ze środków zablokowanych art. 177 może służyć tylko do wypłacania zobowiązań wymagalnych państwa. A wy będziecie je wydawać inaczej. Na co? Uwaga, na Policję.

Ten fundusz, szanowni państwo, będzie zupełnie poza Sejmem, bo Policja, czyli pan minister Kamiński, wyda go, jak zechce i na co zechce. Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo proszę, pani poseł Hanna Gill-Piątek, klub Lewica. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Ustawa budżetowa jest jedną z najważniejszych ustaw dla działania państwa. Dziś przedstawiany jest nam projekt dotyczący realizacji tegorocznego budżetu, który ma umożliwiać przekazanie środków na realizację zadań publicznych w bieżącym roku oraz wykorzystanie ich po upływie roku budżetowego. Szanowni państwo, rozumiemy, że rząd chce w ten sposób, w sposób jak najbardziej prawidłowy zrealizować budżet. W końcu zapewniał ostatnio, że jego wykonanie będzie poddane wnikliwej analizie. Jej jakość, zgodnie ze swoimi obowiązkami, zapewni prezes Najwyższej Izby Kontroli, który bez wątpienia bardzo dokładnie sprawdzi, jak rząd gospodarował finansami publicznymi. Cieszy nas, że poprawiają się standardy kontroli państwowej, choć nie cieszą nas przyczyny tego faktu. Uważamy jednak za nie do przyjęcia tryb, w jakim wnoszony jest projekt. Otrzymujemy go jako posłanki i posłowie o godz. 20 dzień przed posiedzeniem Sejmu. W takim terminie nie jesteśmy w stanie dogłębnie zanalizować propozycji rządu, a nasi eksperci nie są w stanie ocenić realnych jego skutków. Decydowanie z dnia na dzień o przeznaczeniu niemałej kwoty 3 mld zł jest niepoważnym traktowaniem przez rząd PiS i nas wszystkich w tej Izbie, i naszych wyborców. Świadczy to dobitnie o stopniu bałaganu i degrengolady, z jakimi mamy do czynienia obecnie w państwie. W państwie, które powinniśmy chronić i mądrze gospodarować, bo tego oczekują od nas ludzie.

Tak nie działa odpowiedzialna władza. Tak nie wygląda nowoczesne państwo. Efektem jest wiele ustaw pisanych na kolanie i bubli prawnych, których konsekwencje ponoszą potem obywatele. Nie za to jako posłowie bierzemy niemałe pieniądze, żeby firmować tak niskie standardy zarządzania państwem. Oczekujemy od rządu szybkiego naprawienia tego stanu. Jako Lewica jesteśmy zawsze za poprawą sytuacji w służbie zdrowia i za podwyższaniem standardów usług publicznych. Wiemy, jaka jest jakość pracy na komisariatach - jesteśmy za podniesieniem jakości pracy Policji. Dlatego zdecydowaliśmy się poprzeć przedstawiony projekt, choć nie popieramy trybu, w jakim jest procedowany.

Nie ma pana posła. Czy ktoś z pań i panów posłów chce zgłosić się jeszcze do zadania pytania? Jeżeli nie, zamykam listę. Jako pierwszy pan poseł Wiesław Szczepański, klub Lewica. 1 minuta na zadanie pytania. Nie ma pana posła. Bardzo proszę.

Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Pojawiają się zapisy dotyczące wydatkowania środków na Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną - i bardzo dobrze, że tak się dzieje; rzeczywiście wiemy, że to są jednostki, które są niedofinansowane. Natomiast moje pytanie jest takie: Jak w przeciągu najbliższych 3 miesięcy, biorąc pod uwagę ustawę o zamówieniach publicznych, wydacie ponad 100 mln zł? Albo już są jakieś projekty, które są realizowane, na które nie ma pieniędzy i trzeba je uzupełnić, albo rzeczywiście będzie poważny problem z wydatkowaniem tych środków. Podobnie jest, jeżeli chodzi o zapis mówiący o tym, że sfinansowanie tych zadań nastąpi ze środków uzyskanych z wydatków zablokowanych. No, 3 mld zł wydatków zablokowanych. Pytanie jest więc takie: Czego nie wykonamy w tym roku i w tym budżecie po to (Dzwonek), ażeby można było tę ustawę zrealizować? Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Pani poseł Zofia Czernow, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Chciałam zapytać w sprawie kwoty 2 mld zł, która zostanie przekazana do Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia opieki zdrowotnej. Może pytanie dotyczy tego, ile z tej kwoty zostanie przekazane na oddłużenie szpitali, bo sytuacja w szpitalach jest dramatyczna. Kiedy te pieniądze zostaną przekazane na oddłużenie tych szpitali i jakie kryteria będą stosowane przy podziale tych środków na poszczególne placówki?

Wysoka Izbo! Prawo i Sprawiedliwość od kilku lat ma na sztandarach, jeżeli chodzi o system ochrony zdrowia, dwa postulaty: skrócenie kolejek do lekarzy specjalistów oraz oddłużenie szpitali, w szczególności tych powiatowych.

Dziś ich zobowiązania sięgają kwot pomiędzy 14 a 17 mld zł, w zależności od tego, jak będziemy je liczyć. Panie ministrze, w związku z tym moje bardzo konkretne, precyzyjne pytania. Na co dokładnie zostaną przeznaczone te środki, które będą skierowane do Narodowego Funduszu Zdrowia? I czy możemy liczyć realnie na poprawę sytuacji w systemie ochrony zdrowia? Bo dziś wiemy, że ten system jest na skraju zapaści, on ledwo zipie. Dzisiaj szpitale są niewydolne. A jak dobrze pan pewnie zgaduje, każdy z nas interesuje się systemem ochrony zdrowia, bo albo mamy kogoś bliskiego (Dzwonek), kto niestety został dotknięty chorobą, albo sami chorujemy. A więc to jest pilne zobowiązanie względem Polaków.

Także nie ma. Bardzo proszę, pani poseł Marcelina Zawisza, Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Trwa protest mieszkańców Grodkowa i gminy Grodków przeciwko likwidacji od 1 stycznia 2020 r. nocnej i świątecznej opieki medycznej w Grodkowie w ramach planu naprawczego dla Brzeskiego Centrum Medycznego. Mam pytanie: Czy te pieniądze, które zostaną przeznaczone na NFZ, będą przeznaczone na zatrzymanie likwidacji szpitali, oddziałów szpitalnych nocnej i świątecznej opieki medycznej, tak żeby obywatele i obywatelki mogli poczuć się bezpiecznie? Likwidacja nocnej i świątecznej opieki medycznej w Grodkowie pozbawi dostępu do sprawnej i bezpiecznej opieki medycznej 20 tys. osób.

Chciałabym wiedzieć, na co dokładnie zostaną przeznaczone te pieniądze, i w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość planuje zatrzymać tę plagę zamykania oddziałów szpitalnych nocnej i świątecznej opieki (Dzwonek) medycznej oraz szpitali. Bardzo proszę, pani poseł Krystyna Skowrońska, Koalicja Obywatelska. Powiem, z czego się cieszę - że w tej ustawie okołobudżetowej nie idą pieniądze na telewizję publiczną, bo to są zmarnowane pieniądze. Ale nie cieszę się z trybu przekazania pieniędzy na Narodowy Fundusz Zdrowia. Dlaczego? Panie ministrze, no, jest pan cesarzem: 2 mld zł i nikt nie wie, na co one zostaną przeznaczone. W ubiegłym roku kwota lekko powyżej 1 mld zł dawała panu dowolność: na nadwykonania, na niektóre procedury, które państwo chcieli wprowadzić, żeby były wyższe świadczenia za to. Tu nic, nic nie wiemy. 17 mld długów szpitali, wyrok Trybunału Konstytucyjnego mówiący, że to rządzący odpowiadają za ochronę zdrowia i za te wszystkie długi, a państwo śpicie. 18 miesięcy - trzeba zmienić przepisy prawa. I w tym zakresie, panie ministrze, czekamy, że rzetelnie minister i premier podejdą (Dzwonek) do sprawy ochrony zdrowia, tak aby nie zamykać szpitali.

Dziękuję bardzo.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Koleżanki i Koledzy! Panie Ministrze! Usłyszeliśmy tutaj o kierunkach przesunięć, ale tak naprawdę nie usłyszeliśmy, na co dokładnie te środki mogą pójść. Chciałbym, panie ministrze, powiedzieć, że sytuacja w szpitalach powiatowych na Pomorzu Zachodnim jest katastrofalna. To są niedoszacowane procedury. Szanowni państwo, oczekuję jasnej odpowiedzi, czy te środki mogą pójść i pójdą również na szpitale powiatowe. Jeżeli jest, szanowni państwo, tak dobrze, to pomóżmy tym samorządom, bo one dzisiaj biorą kredyty na funkcjonowanie. Naprawdę taka sytuacja jest. Bardzo o to proszę i apeluję o to. Pani poseł Małgorzata Pępek, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Wsparcie jednostek Policji i ochrony zdrowia jest zasadne, niemniej jednak nie przestrzegacie państwo reguły wydatkowej, nie dbacie o stabilność finansów publicznych. Jak można łamać regułę wydatkową? Rezerwa, która ma służyć do wypłaty zobowiązań wymagalnych, powinna być skierowana, tak jak mój poprzednik powiedział, do jednostek samorządu terytorialnego na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, ponieważ samorządy rezygnują z inwestycji służących mieszkańcom z tego powodu, brakuje im już na bieżące wydatki. Pytam: Kiedy zwrócicie jednostkom samorządu terytorialnego wydatkowane pieniądze na utrzymanie oświaty - to jest ogromny problem, nie wiem, czy pan minister zdaje sobie z tego sprawę - oraz kiedy zrekompensujecie utracone dochody z PIT-ów? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Mirosław Suchoń, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

I od razu, panie ministrze, rodzi się pytanie, czy to są takie same ambulanse jak te, które stoją we Wrocławiu, wobec których prokuratura prowadzi postępowanie. Nie wiadomo dlaczego karetki, które miały ratować Polaków, stoją nieużytkowane, ponieważ ktoś nie dopilnował podstawowych elementów w zakresie zamówienia publicznego. A więc, panie ministrze, bardzo proszę o wyjaśnienie: Jakie to będą ambulanse? Czy to jest tak, że te ambulanse znowu będą stały i zamiast ratować życie Polaków, będą elementem wystroju parkingów, czy też państwo wdrożyli jakiekolwiek procedury, które zapobiegają tego typu (Dzwonek) skandalicznym przypadkom, które państwa rząd przez ostatnie lata Polakom fundował? Bardzo proszę, pani poseł Izabela Leszczyna, Koalicja Obywatelska. Trzy pytania, bo sprawa jest naprawdę poważna. Proszę, żeby pan minister potwierdził, czy środki wydane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Fundusz Wsparcia Policji są poza limitem wydatków reguły, poza tą częścią, za którą odpowiada minister finansów. Drugie pytanie dotyczy tego trzeciego sposobu psucia ustawy o finansach publicznych. Chodzi o niewygasy. Można te środki wydawać do 30 marca następnego roku. Po co wydłużacie ten termin o kolejny miesiąc? Naprawdę nie da się ambulansów kupić w ciągu 3 miesięcy? Wtedy się nie robi niewygasów. Dlaczego środki wydawane w ramach Funduszu Wsparcia Policji pozwala pan wyjąć nie tylko spod kontroli Sejmu, o czym już mówiłam, ale nawet spod kontroli ministra finansów? Otóż środki w tym funduszu mogą być (Dzwonek) zmieniane dowolnie, bez zgody ministra finansów i Komisji Finansów Publicznych. Biorąc pod uwagę to, co służby specjalne robią w Polsce, to jest rozbój na prostej drodze. Bardzo proszę, pan poseł Artur Łącki, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Dajemy już te pieniądze i najprawdopodobniej Koalicja Obywatelska nie będzie przeciwna tej ustawie. Ale od razu cisną się na usta pytania, i to w związku z wystąpieniem pana premiera Morawieckiego, który mówił chociażby o pomocy dla szpitali powiatowych. Szczególnie chodzi mi o szpital w Kamieniu Pomorskim, któremu grozi już nie zamknięcie jakichś tam oddziałów, tylko w ogóle zamknięcie. A jest to szpital położony na terenie nadmorskim, turystycznym, który co roku odwiedza przynajmniej 200 tys. ludzi, i dla tych ludzi również ten szpital jest, czyli dla bezpieczeństwa naszych Polaków, naszych turystów. Panie ministrze Kamiński, nie wiem, czy pan wie, ale samorządy, szczególnie samorządy w miejscowościach turystycznych, co roku partycypują (Dzwonek) w kosztach bezpieczeństwa naszych turystów. Bardzo proszę, pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! 2 mld jest to kwota niewystarczająca, żeby zlikwidować największe w historii kolejki do specjalistów, jak również żeby nie zadłużać szpitali. Panie ministrze, w mojej opinii rząd nie realizuje ustawy dotyczącej 6% PKB na ochronę zdrowia. Obiecywaliście to rezydentom, w zamian rezydenci otrzymywali pouczenia marszałka Senatu, który na bezpłatnym urlopie odbywał płatne dyżury. Szanowni państwo, procenta PKB nie odnosicie do PKB sprzed roku czy też do prognoz. Jaka jest sytuacja? Polacy wydają rocznie średnio 1551 zł na prywatne usługi medyczne i to jest realny problem. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że serial pt. „Zrównoważony budżet państwa” trwa w najlepsze.

Chciałem, po pierwsze, zapytać pana ministra zdrowia, jak to jest, że na poprzednim posiedzeniu Sejmu nie chciał 2 mld, mimo że proponowaliśmy mu ten wzrost akcyzy na papierosy i alkohol, żeby to przejął, a już teraz chce 2 mld, bo tyle jest zapisane na szeroko rozumianą służbę zdrowia. Drugie pytanie. Prosiłbym rozwinąć, co w ramach tego funduszu zapasowego NFZ mają te pieniądze zabezpieczyć, bo jest to dosyć niejasne.

Dziękuję bardzo, panie pośle. Wysoka Izbo! Chciałem zapytać pana ministra, jak to się stało, że rząd wreszcie odkrył, że polska Policja jest niedoinwestowana. Chciałbym zadać konkretne pytania. Czy to będą prezenty świąteczne dla wybranych komisariatów? Czy pójdą te pieniądze na nasze bezpieczeństwo, czyli zwiększenie liczby policjantów? Przypominam, że liczba wakatów w Policji za rządów Prawa i Sprawiedliwości ciągle się zwiększa i pod koniec 2018 r. liczba tych wakatów doszła do 4294. Chciałbym zapytać pana ministra zdrowia, na jakim etapie jest ministerstwo z pracami w sprawie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że samorządy nie mogą pokrywać strat szpitali. Dziękuję bardzo, panie pośle. Na tym zakończyliśmy zadawanie pytań. Jako pierwszy na pytania odpowiada podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia pan minister Janusz Cieszyński. Bardzo proszę.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Dziękuję bardzo za te pytania. Przede wszystkim chciałem też podziękować za to, że - wygląda na to - mamy już taką zupełnie ponadpolityczną zgodę co do tego, że te środki do Narodowego Funduszu Zdrowia warto przekazać. Bardzo mnie cieszy, że te deklaracje, które państwo składaliście też przed wyborami, teraz znajdują swoje potwierdzenie w państwa stanowiskach. Jeżeli chodzi o konkretne pytania, to pani poseł Czernow pytała, kiedy będzie oddłużenie szpitali. Z pewnością pani wie, że Narodowy Fundusz Zdrowia zgodnie z ustawą nie może być organem założycielskim żadnego podmiotu leczniczego. Co więcej, Narodowy Fundusz Zdrowia nie ma wśród swoich zadań oddłużania placówek ochrony zdrowia, tylko zakup świadczeń, czyli zakup kolejnych usług dla polskich pacjentów. Staram się odpowiedzieć na pytania najlepiej, jak potrafię. Dziękuję. Szanowni Państwo! Warto powiedzieć, że dzięki dobrej sytuacji gospodarczej, dzięki dobrym wynikom budżetu państwa udaje się systematycznie od 3 lat każdego roku właściwie w bardzo podobnej formule - to zawsze dzieje się mniej więcej w okolicach grudnia - przeznaczać dodatkowe środki właśnie poprzez ten fundusz zapasowy na Narodowy Fundusz Zdrowia. W 2017 r. Narodowy Fundusz Zdrowia dostał 1 mld zł, który przeznaczył na spłaty nadwykonań z czasów, kiedy rządziła Platforma Obywatelska i tych nadwykonań nie płacono.

My jako Ministerstwo Zdrowia, jako Narodowy Fundusz Zdrowia z projektem ustawy zapoznaliśmy się wczoraj. Te środki trafią do ogólnego budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia i w momencie, w którym już. W momencie, w którym te środki wpłyną do Narodowego Funduszu Zdrowia, dokonamy odpowiedniej zmiany planu finansowego i taka zmiana planu finansowego za każdym razem jest opiniowana przez komisje sejmowe, zarówno przez Komisję Zdrowia, jak i przez Komisję Finansów Publicznych, której członkowie tutaj wiele razy już dzisiaj zabierali głos w tej sprawie, więc na wszystkie te pytania chętnie państwu odpowiemy, kiedy zaprezentujemy państwu właśnie zmianę planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia. To jest też odpowiedź na pytanie pani poseł Zawiszy, która pytała, na co te pieniądze zostaną przeznaczone. Szanowni Państwo!

Tam jest jednoznacznie wskazane, na co chcemy przeznaczyć te środki. To jest m.in. rozszerzenie programu nielimitowanego finansowania porad specjalistycznych.

W podstawowej opiece zdrowotnej program płacenia za wynik.

Tylko w tym roku są trzy wzrosty wycen w ciągu roku, ze skutkiem od stycznia, i ponad 900 mln zł dodatkowych środków dla szpitali powiatowych, tych szpitali, które są najbliżej pacjentów. Pan poseł Suchoń pytał, czy są to takie same ambulanse jak te, które stoją we Wrocławiu, i czy ktoś nie dopilnował przetargów. Szanowny panie pośle, ambulanse, które stoją we Wrocławiu, zostały kupione przez podległą województwu, w którym rządzi Platforma Obywatelska, dyrekcję pogotowia ratunkowego. Te ambulanse, szanowni państwo, trafią do placówek w całym kraju, natomiast nie wszyscy dysponenci byli w stanie te środki wykorzystać, m.in. zachodniopomorskie pogotowie ratunkowe siedmiu karetek nie było w stanie wykupić w terminie. Przypomnę, że przeznaczyliśmy środki na 200 karetek: 150 udało się kupić, a na kupno 50 potrzebujemy trochę więcej czasu, do końca kwietnia przyszłego roku. Pan poseł Szczerba pytał o ustawę 6% i dlaczego to jest w ten sposób liczone. Szanowny panie pośle, miałem okazję sprawdzić, że pan głosował za przepisem tej treści. głosował pan za przepisem tej treści i prawdopodobnie głosował pan za nim dlatego, że to jest przepis w kształcie, który jeden do jednego jest przeniesiony z porozumienia, które pan prof. Łukasz Szumowski zawarł z przedstawicielami porozumienia rezydentów. Szanowni państwo, treść. Szanowni państwo, na szczęście jest to porozumienie, którego treść jest dostępna w Internecie i każdy może się z nim zapoznać. Każdy może też zapoznać się z treścią ustawy o świadczeniach i tego konkretnego przepisu, i kiedy państwo sobie te kwestie porównacie, zobaczycie, że sytuacja jest dokładnie taka, jak ją teraz państwu opisuję. Jeżeli chodzi o pytanie pana posła Paszyka - dlaczego nie chcieliśmy 2 mld zł z podatku akcyzowego - to, szanowni państwo, są to środki, które właśnie w budżecie. Te środki, które przeznaczamy dzisiaj, to są właśnie środki budżetowe. Szanowni państwo, dlatego popieraliśmy projekt, który prowadził do wzrostu wpływów z podatku akcyzowego, żeby w budżecie państwa było więcej środków i żeby takie zasilenia, o których dzisiaj mówimy, mogły być realizowane. Kiedyś wpływy z podatków były na o wiele niższym poziomie i nie było dodatkowych środków dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeżeli chodzi o wyrok Trybunału Konstytucyjnego, szanowni państwo, my szanujemy wyroki sądów. Jak państwo z pewnością wiecie, po tym, jak taki wyrok zapadnie, sąd przygotowuje szczegółowe uzasadnienie i trudno wyobrażać sobie, żeby na kolanie pisać przepisy, zanim takie uzasadnienie zostanie nam zaprezentowane. Kiedy ministerstwo je otrzyma, ono będzie też dostępne, podane do publicznej wiadomości, niezwłocznie przystąpimy do prac, żeby wyrok Trybunału Konstytucyjnego w terminie, który został wskazany, czyli 18 miesięcy, niezwłocznie wykonać. Dziękuję, panie ministrze. Proszę teraz o zabranie głosu sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pana ministra Macieja Wąsika. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Odpowiadając na pytania, które padły w tej debacie, powiem tak. Wydatki niewygasające programu modernizacji w wysokości 103 mln to nie są wydatki, które są uzależnione od bieżących zamówień publicznych. Te zamówienia już zostały przeprowadzone, zresztą dosyć sprawnie. Z różnych przyczyn pewna część wydatków inwestycyjnych z programu modernizacji uległa opóźnieniu, z różnych przyczyn opóźnione zostały pewne inwestycje, tj. 41 pozycji, które będą ukończone bądź oddane na początku przyszłego roku. W związku z tym te płatności muszą być przesunięte jako wydatki niewygasające, tj. 61 mln wydatków Policji, to 19 pozycji inwestycyjnych, Straży Granicznej - 13 pozycji, 37 mln niespełna, Państwowej Straży Pożarnej - 5 pozycji, 4,5 mln, i Służby Ochrony Państwa - 1,3 mln zł. Tu są podpisane umowy, to są klasyczne wydatki niewygasające, które będą zrealizowane na początku przyszłego roku.

Musi realizować utrzymanie swoich obiektów, środków transportu.

To istotne zwiększenie finansowania ustawowych zadań Policji dotyczących bezpieczeństwa publicznego, wewnętrznego i bezpieczeństwa obywateli. Szanowni państwo, pamiętam czasy nie tak odległe, 5 lat temu, 6, 7, 8 lat, kiedy słyszeliśmy ciągle, że brakuje na papier w Policji, że brakuje na paliwo w Policji, że brakuje wszystkiego w Policji. My staramy się, żeby polska Policja była dobrze zaopatrzona i żeby mogła sprawnie realizować zadania z dziedziny bezpieczeństwa. Jestem przekonany, że realizuje je coraz sprawniej, ale do tego potrzebne są środki finansowe, gdyż - jak doskonale wiecie, szanowni państwo posłowie - bezpieczeństwo jest dziedziną niezwykle kosztowną. Dlatego chcemy realizować te zadania i przeznaczamy środki na Fundusz Wsparcia Policji. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Ogólnie od strony finansowej. Było pytanie, czy Narodowy Fundusz Zdrowia jest ujmowany w regule wydatkowej. Konstrukcja reguły wydatkowej jest wielostopniowa. Pani poseł sprecyzowała pytanie: Czy jest w części, za którą odpowiada minister finansów? Generalnie minister finansów odpowiada za czy sprawuje ogólny nadzór nad finansami publicznymi, w związku z czym wszystko, co mieści się w szeroko rozumianym pojęciu środków publicznych, znajduje się pod ogólnym nadzorem ministra finansów. Oczywiście pod nadzorem bezpośrednim ministra finansów tak naprawdę jest budżet państwa jako taki. Wszystkie inne fundusze czy wszystkie inne formy, w jakich wydatkowane są środki publiczne, są podporządkowane poszczególnym dysponentom, przy czym oczywiście budżet również jest podzielony na części podporządkowane poszczególnym dysponentom. Minister finansów o tyle ma kontrolę nad całością, że dokonuje de facto fizycznych płatności na rzecz tych dysponentów czy przekazuje środki, zwiększa plany finansowe i kontroluje wykonanie. No i jest, i nie jest, natomiast środki, które są wydawane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, również są ujmowane w konstrukcji reguły wydatkowej, przy czym, tak jak mówiłem, to jest dosyć skomplikowany proces wyliczania środków, które mogą być wydatkowane w danym roku budżetowym. Ta konstrukcja jest wielostopniowa, ale w skrócie rzecz ujmując, środki Narodowego Funduszu Zdrowia również wpływają na wielkość stabilizującej reguły wydatkowej. Po drugie, padały tutaj takie głosy, one gdzieś się już pojawiały też wcześniej, że została złamana stabilizująca reguła wydatkowa. Otóż nie została złamana stabilizująca reguła wydatkowa.

W trakcie roku jak do tej pory.

Jeżeli będzie przekroczona, to oczywiście stosowne kroki podejmą stosowne organy, w tym zapewne Wysoka Izba, ale - jak mówię - rolą ministra finansów jest do tego nie dopuścić i do tego nie doszło. Jeśli chodzi o całkowite wyjęcie spod kontroli ministra finansów tych środków na Fundusz Wsparcia Policji, to ten przepis, który jest w ustawie, dotyczy tylko i wyłącznie zmiany planu finansowego, jeśli chodzi o tę wpłatę, która jest dokonywana tą ustawą, natomiast to, jak przeznaczenie środków. Skoro jest już ustawa, to ta wpłata nie musi przechodzić całej procedury sejmowej, tak jak wszystkie inne zmiany w funduszach celowych, ponieważ to już jest uregulowane właśnie w tej ustawie. Natomiast jeżeli te środki już będą wydatkowane z Funduszu Wsparcia Policji, ukierunkowywane na konkretne rzeczy, to każda zmiana takiego przeznaczenia oczywiście będzie opiniowana, będzie pod nadzorem ministra finansów i będzie opiniowana przez Wysoką Izbę. Padały też tutaj pytania o subwencję oświatową, o zwiększenie tej subwencji, wsparcie dla samorządów.

Ta dyskusja ma doprowadzić do zasadniczego przebudowania finansów samorządów jako takich, chodzi tu nie tylko o subwencję oświatową, tylko w ogóle o kwestie finansowania samorządu i zasilania samorządu, jednostek samorządu terytorialnego, ale to wymaga przebudowy całego systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Mam nadzieję, że uda się do tego doprowadzić, bo rzeczywiście ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ma swoje lata i wymaga zmian. Jeszcze jedna rzecz istotna w tej ustawie.

Czekamy teraz na wynik budżetu państwa i ostateczne rozliczenia.

Będziemy blokować to, co nie będzie wykorzystane w normalnym procesie wykonywania budżetu państwa.

Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował pilny rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, zawarty w druku nr 56, do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Jednocześnie marszałek Sejmu na podstawie art. 73 ust. 2 regulaminu Sejmu wyznacza termin przedstawienia sprawozdania przez komisję umożliwiający jego rozpatrzenie w dniu dzisiejszym. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 2. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 43) Proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury pana Andrzeja Bittela o przedstawienie uzasadnienia projektu. Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, zawarty i opisany w druku nr 43. Projekt ten stanowi jeden z priorytetów rządu, jeden z priorytetów Ministerstwa Infrastruktury, ponieważ łączy się z działaniami związanymi z przeciwdziałaniem wykluczeniu komunikacyjnemu wielu polskich miast, miasteczek i wsi. W roku 1990 w Polsce funkcjonowało blisko 26 tys. km linii kolejowych.

Stąd też celem rządu jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, eliminowanie tego niedobrego zjawiska. Takie działania podejmujemy konsekwentnie w ramach realizacji krajowego programu kolejowego, programu utrzymaniowego.

Po pierwsze, uściślamy warunki likwidacji linii kolejowych, po to aby wyeliminować ich niekontrolowaną likwidację bez wiedzy i zgody odpowiednich organów. W tym celu jest przywracana zgoda ministra właściwego ds. transportu na likwidację linii kolejowej bocznicy czy odcinka linii kolejowej. Doprecyzowujemy procedurę likwidacyjną poprzez obowiązek przeprowadzenia analiz i poinformowania zainteresowanych podmiotów i organów o zamiarze likwidacji. Wprowadzamy również możliwość karania pieniężnego za likwidację linii kolejowej lub bocznicy kolejowej z naruszeniem przepisów ustawy. Ta możliwość zostaje stworzona, jeśli chodzi o prezesa Urzędu Transportu Kolejowego jako niezależnego regulatora w tej sferze. Drugi ważny aspekt to umożliwienie użyczania jednostkom samorządu terytorialnego nieruchomości pozostałych po zlikwidowanych liniach kolejowych lub ich odcinkach. I to jest uelastycznienie, bo w tej chwili możemy w ramach procedur, które już występują w polskim prawie, przekazywać na rzecz samorządu terytorialnego nieruchomości do wykorzystania na dzieło transportowe, ale chcemy też mieć możliwość niekoniecznie rozporządzenia ostatecznego, przekazania nieruchomości. Chodzi też o elementy związane z użyczeniem, po to aby samorząd mógł ewentualnie zagospodarować je na swoje cele, ale żebyśmy mieli utrzymany korytarz transportowy w rozumieniu niekoniecznie drewnianych podkładów i starej, wyeksploatowanej linii kolejowej, ale w rozumieniu nieruchomości, które taki korytarz transportowy.

Trzecia ważna kwestia to realizacja wojewódzkich połączeń kolejowych poza granicą województwa. W tej chwili ta sytuacja jest opisana inaczej: najbliższą stacją. To nie jest rozwiązanie, które powoduje, że system kolejowy jest spójny.

Jednocześnie stwarzamy zachęty związane z możliwością dofinansowania ze środków Funduszu Kolejowego modernizacji napraw pojazdów taborowych, taboru lub też jego zakupu, jeśli takie dobre, korzystne dla sieci kolejowej rozwiązania dotyczące systemu kolejowego będą wprowadzane.

Będziemy inwestować w polską kolej ogromne pieniądze w najbliższych latach i w kolejnej perspektywie unijnej.

Można powiedzieć, że jest to przepis, który jest zbliżony do przepisu specustawy drogowej.

Ważne są przepisy dotyczące umożliwienia przekazywania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na wniosek ministra właściwego do spraw transportu na rzecz PKP PLK skarbowych papierów wartościowych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego oraz możliwości przeznaczenia środków uzyskanych z tych papierów na realizację inwestycji. Doregulowujemy również kwestię związaną z utrzymaniem infrastruktury drogowej lub sieciowej realizowanej w ramach inwestycji modernizacyjnych, mam na myśli wiadukty i drogi równoległe, aby ciężar utrzymania tych dróg w określonym zakresie brały na siebie właściwe samorządy.

To też w sposób oczywisty ułatwi inwestowanie w ten środek transportu. Jest jeszcze kilka drobniejszych spraw, takich jak doprecyzowanie zasad kalkulacji opłat za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej lub świadczonych usług, wprowadzenie w życie do naszego porządku prawnego wyroku TSUE, który nakazał peron pasażerski zakwalifikować do elementów infrastruktury kolejowej, czyli do pakietu minimalnego dostępu. Jest także kwestia związana z uregulowaniem ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych tajemnic prawnie chronionych w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Urząd Transportu Kolejowego. Chodzi o zmianę w Kodeksie postępowania cywilnego, która ma zabezpieczyć ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa w tym postępowaniu. Szanowni Państwo! Wysoka Izbo! Jest to bardzo istotne przedłożenie, które będzie stwarzało nam warunki do tego, aby realizować krajowy program kolejowy i programy utrzymaniowe oraz budować jeszcze lepszy system transportowy naszego państwa. Dziękuję bardzo. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jako pierwszy pan poseł Jerzy Polaczek, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawić stanowisko naszego klubu w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, druk nr 43. Bardzo szczegółowo zreferował ten projekt pan minister Andrzej Bittel. Chciałbym tylko raz jeszcze wyróżnić te najważniejsze elementy, które oddają istotę tej bardzo ważnej rządowej nowelizacji przyspieszającej inwestycje kolejowe, dającej nowe możliwości współpracy z samorządami terytorialnymi i realizującej również w sposób bardzo aktywny rozwiązania europejskie. Chciałbym przypomnieć, iż założenia tego projektu obejmują stworzenie właśnie takich instrumentów prawnych, dzięki którym będzie można lepiej niż dotychczas zapobiegać przede wszystkim niepożądanej degradacji infrastruktury kolejowej w Polsce, a to było jedno z najbardziej dostrzeganych w opinii społecznej zjawisk, w szczególności po 1989 r. Bardziej szczegółowymi celami tej nowelizacji są, tak jak powiedziałem, utrudnienie likwidacji linii kolejowych i zatrzymanie degradacji infrastruktury kolejowej na terenach po liniach kolejowych, co do których została już wydana decyzja o ich likwidacji. To jest, dalej, uregulowanie kwestii połączeń kolejowych na granicach województw, usunięcie barier i problemów dotyczących efektywnej realizacji inwestycji kolejowych, w szczególności w ramach krajowego programu kolejowego, z udziałem środków europejskich, to stworzenie możliwości realizacji i realizacja infrastruktury drogowej w ramach prowadzonych inwestycji dotyczących modernizacji infrastruktury kolejowej, a następnie zarządzanie i utrzymywanie wybudowanej infrastruktury drogowej czy powstrzymanie nieuprawnionej komunalizacji gruntów Skarbu Państwa zajętych pod infrastrukturę kolejową. W punktach można przedstawić ten projekt w sposób następujący. Tak lapidarnie, najważniejszym celem ustawy jest wstrzymanie procesu likwidacji linii kolejowych. Po drugie, to użyczenie nieruchomości pozostałych po zlikwidowanych liniach kolejowych lub odcinkach tych linii. Mówił już o tym szczegółowo pan minister Andrzej Bittel i to przyjmujemy jako klub parlamentarny z wielką satysfakcją. Myślę, że w szczególności ten pozytywny odbiór będzie na poziomie samorządów wojewódzkich. Po czwarte, celem ustawy jest usprawnienie realizacji inwestycji kolejowych.

Myślę, że to zostanie również odnotowane bardzo pozytywnie przez jednostki samorządu terytorialnego realizujące tego rodzaju zadania. Po szóste, to zmniejszenie obciążeń wojewodów i ograniczenie nieuzasadnionej komunalizacji gruntów Skarbu Państwa zajętych pod infrastrukturę kolejową czy ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa prawnie chronionej w postępowaniu administracyjnym. Reasumując, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość bardzo pozytywnie ocenia rządowy projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Ta ustawa w swoim założeniu i, myślę, w zakresie efektów, jakie będzie przynosiła, ułatwi procesy inwestowania w infrastrukturę kolejową, zmaksymalizuje wykorzystanie tej infrastruktury po to, aby przewozy kolejowe były wykonywane w sposób należyty, i zapobiegnie niezasadnemu i pospiesznemu likwidowaniu linii kolejowych. A zatem przeciwdziałamy tym procesom, które obserwowaliśmy w różnych odsłonach w niektórych kadencjach po 1989 r. Projekt zawiera również bardzo konkretne instrumenty prawne, które przyczynią się do rozwoju i efektywnego wykorzystania infrastruktury kolejowej. Biorąc powyższe pod uwagę, zaproponowane zmiany oczywiście zasługują na nasze poparcie. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość będzie aktywnie pracował w Komisji Infrastruktury po to, aby to przedłożenie rządowe weszło w życie w jak najszybszym racjonalnym terminie. Bardzo serdecznie wyrażamy również tutaj uznanie przedstawicielom rządu, Ministerstwu Infrastruktury za podjęcie tego bardzo ważnego aspektu inwestycji w infrastrukturę, która oddziałuje w sposób bardzo konkretny na komunikację wieluset tysięcy ludzi w Polsce codziennie. Bardzo proszę, pan poseł Mirosław Suchoń, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam przyjemność i zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, druk nr 43. Szanowni Państwo! Projekt ustawy, który był przedstawiony bardzo obszernie przez pana ministra, jest prezentowany jako ten, który wnosi pewną nową jakość w obszar związany z transportem kolejowym. Rzeczywiście jest tam kilka elementów, o których można powiedzieć, że są interesujące: możliwość nieodpłatnego przejęcia przez samorząd bądź zarządcę linii kolejowej odcinka w zarządzanie, wprowadzenie zmiany w definicji przewozów międzywojewódzkich, które będą mogły być wykonywane na obszarze do 30 km w głąb województwa, a nie, tak jak jest teraz, do najbliższej stacji, czy też wprowadzenie przez pana ministra, przez ministerstwo i rząd, procedury postępowania w przypadku likwidacji linii kolejowych - poszerzonej, bym powiedział. Ale oczywiście zazwyczaj rząd głośno mówi o tym, co jest pozytywnego w projektach, a już ciszej jest o tym, co budzi kontrowersje, co w tych projektach wymaga bardzo głębokiej debaty, a może nawet zmian. Po pierwsze od tego, że z likwidacją linii kolejowych, panie ministrze, jest tak, że przecież pański rząd, rząd, w którym pan jest ministrem od 2016 r., zlikwidował co najmniej 272 km linii kolejowych. Co więcej - bo można powiedzieć, że to było zaraz po przyjęciu, więc być może siłą jakiegoś rozpędu - w styczniu 2017 r. ogłoszono przetarg na likwidację linii Brodnica-Kowalewo Pomorskie, odcinając Golub-Dobrzyń, czyli miasto stolicę powiatu, od połączeń kolejowych. A więc to pokazuje, że tak naprawdę wprowadzenie przepisów dotyczących tych zmian nie bardzo ma się do rzeczywistego postępowania i rzeczywistych chęci. Bo gdyby ta chęć zachowania linii kolejowych w obecnym stanie, deklarowana chęć, była chęcią rzeczywistą, to do tych likwidacji z pewnością by nie doszło. Co więcej, likwidacja czy zachowanie linii kolejowych wcale nie oznacza tego, że one nie podlegają dalszej degradacji. Możemy w całej Polsce znaleźć takie przykłady, jak choćby linia nr 190 na odcinku Bielsko-Biała - Skoczów.

Warto zatem, wprowadzając te przepisy do porządku prawnego, rozpocząć również rzeczywiste działania, bo te przepisy nie uratują linii kolejowych, nie spowodują, że będzie jeździło więcej składów i że będzie to bardziej przyjazne dla pasażerów.

Musimy jasno sobie powiedzieć, że drastyczne podwyżki cen prądu, które czekają nas od nowego roku, spowodują wzrost kosztów działalności przewoźników kolejowych, w związku z czym bardzo silna będzie presja dotycząca podwyżki cen biletów. To jest oczywiście kolejny koszt dla przewoźników, który wygeneruje impuls skutkujący chęcią podwyższenia cen biletów na przewozy kolejowe.

Ten obowiązek - bo w zasadzie wprowadzają państwo obowiązek przejęcia przez samorządy tej infrastruktury, tych dróg czy wiaduktów - nie wiąże się z żadnym dodatkowym dochodem dla samorządów, czyli pomimo że państwo już tak drastycznie obniżyli dochody samorządów, to jeszcze dodatkowo wprowadzacie kolejne elementy, które powodują, że samorządy będą miały coraz mniej środków na nowe inwestycje, które są przydatne mieszkańcom. Tego nie ma. Tych uwag jest bardzo wiele, w związku z czym projekt wymaga głębokiej dyskusji. Wnoszę o przekazanie go do Komisji Infrastruktury celem odbycia bardzo głębokiej debaty i wypracowania jak najlepszego kształtu tego projektu. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Wiesław Szczepański, klub Lewica. Pani Marszałek! W imieniu klubu Lewica mam zaszczyt przedstawić stanowisko dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, druk nr 43. Składa się on z trzech komponentów: inwestycyjnego, organizacji przewozów pasażerskich i ochrony infrastruktury przed likwidacją. Podstawowym komponentem jest projekt inwestycyjny. Pozostałe mają charakter uzupełniający. Rozpatrywany dziś projekt ustawy ma według uzasadnienia wspierać realizację programu „Kolej+” To część prawna tego programu. Z uwagi na upływ czasu nie został on przyjęty w poprzedniej kadencji i po niewielkiej poprawce trafił z powrotem do Izby. Jest to jeden z trzech projektów zmiany ustawy o transporcie kolejowym i nie wiem, panie ministrze, dlaczego są one procedowane w ministerstwie równolegle, a nie jako jeden projekt. Pierwszy projekt dotyczący uniezależnienia Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych od zarządcy infrastruktury wszedł w życie już w poprzedniej kadencji. Jeden jest na etapie prac w komisji prawniczej, nad drugim dziś debatujemy. Zgodnie z omawianym projektem tereny kolejowe, które obecnie są niewykorzystane, zostaną przywrócone do ponownego użytkowania w celach transportowych. Możliwe będzie przekazywanie linii kolejowych do nieodpłatnego korzystania przez samorządy. Likwidacja linii kolejowych będzie możliwa pod warunkiem uzyskania zgody przez ministra infrastruktury. Działania te według wnioskodawcy mają przywrócić eksploatację infrastruktury kolejowej na terenach nieczynnych lub po zlikwidowanej infrastrukturze kolejowej. Samorządy wojewódzkie będą mogły realizować przewozy kolejowe dalej niż do najbliższej stacji za granicą swojego województwa. Według wnioskodawców winno się to przyczynić do poprawy komunikacji na terenach pozbawionych obecnie dogodnych połączeń. Możliwe będzie przeznaczenie środków z funduszu kolejowego na sfinansowanie lub współfinansowanie przez województwo zadań dotyczących zakupu, modernizacji oraz naprawy pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług, ale pod warunkiem zapewnienia połączeń komunikacyjnych pomiędzy sąsiednimi województwami.

Uproszczony zostanie system udzielania gwarancji finansowych umożliwiających rozpoczęcie procedur przetargowych. Wprowadzono nowe źródła finansowania przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych, w tym środki uzyskane z emisji skarbowych papierów wartościowych. To tylko niektóre zmiany. Tempo prac nad tą ustawą zarówno w maju, jak i teraz, było ekspresowe, a projekt nie został przekazany do konsultacji stronie związkowej, z wyjątkiem związku zawodowego „Solidarności” kolejarzy, który i tak nie skorzystał z możliwości przedłożenia państwu swojej opinii. Rodzi się pytanie, czy obowiązek uzyskania decyzji ministra infrastruktury w celu likwidacji linii kolejowej nie będzie elementem zwiększonego nacisku na ich likwidację, a nie - na jej pozostawienie. Jak zostaną zagospodarowane dzisiaj nieczynne bocznice kolejowe? Należy zwrócić uwagę, że umożliwienie emitowania skarbowych papierów wartościowych w celu podniesienia kapitału zakładowego PKP PLK, co jest novum, nie zostało w sposób należyty wyjaśnione. Co więcej, Rządowe Centrum Legislacji w obszernej analizie w żaden sposób nie odniosło się do tej sprawy. Zapis ten budzi niepokój strony związkowej, bo przywołuje najgorsze wspomnienia związane z prywatyzacją, pan pamięta, PKP Energetyka.

Chciałbym zapytać, ile będzie kosztowała emisja i obsługa 11,3 mld papierów wartościowych. Kiedy zostaną one wykupione przez Skarb Państwa?

Co prawda w ustawie mówimy o nieodpłatnym przekazaniu majątku na rzecz samorządów, jednak są to wartości finansowe. W roku 2019 nie wyemitujemy już bowiem papierów wartościowych. Już kończę, pani marszałek.

Widząc potrzebę uchwalenia tej ustawy, klub Lewicy wnosi o skierowanie niniejszego projektu do dalszych prac w Komisji Infrastruktury. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Jacek Tomczak, Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15.

Mam przyjemność przedstawić w imieniu klubu PSL - Kukiz - Koalicja Polska stanowisko wobec niniejszego projektu ustawy. Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw obejmuje zmianę Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe oraz ustawy o transporcie kolejowym. Wśród ciekawych zmian, na które warto zwrócić uwagę, są na pewno zmiany dotyczące wykonania orzeczenia TSUE dotyczącego peronów pasażerskich jako elementu infrastruktury kolejowej oraz zmiany umożliwiające zastosowanie przepisów rozdziału 2b ustawy o transporcie zbiorowym do realizacji inwestycji w zakresie linii tramwajowych poza pasami dróg publicznych.

Nakłada także obowiązek porozumienia w tym zakresie pomiędzy PLK i jednostkami samorządu terytorialnego. Wedle projektodawców celem projektu jest m.in powstrzymanie degradacji infrastruktury kolejowej, w tym korytarzy transportowych, również na terenach linii kolejowych, co do których zostały wydane decyzje o ich likwidacji, oraz uregulowanie kwestii połączeń kolejowych w granicach województw, a także wprowadzenie zmian, które postulowali uczestnicy rynku kolejowego, które mają na celu usunięcie barier i problemów dotyczących efektywnej realizacji inwestycji kolejowych funkcjonujących w praktyce, m.in. dotyczących zapewnienia finansowania projektów realizowanych przez PKP PLK chociażby w postaci ułatwienia udzielania gwarancji. W ramach krajowego programu kolejowego, przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, ustawa wprowadza możliwość organizacji infrastruktury drogowej w ramach prowadzonych inwestycji dotyczących modernizacji infrastruktury kolejowej i późniejszego zarządzania, utrzymywania i budowania tejże infrastruktury drogowej.

Pytanie, czy rozwiązaniem będzie zgoda ministra.

Tego do końca nie wiemy. Wydaje nam się, że wymaga to doprecyzowania. Do tej pory było z tym słabo. Było widać, że projekty unijne realizowane są zaledwie w niewielkim stopniu. A więc zwiększając obciążenia, emitując obligacje bez poprawy działania PKP PLK, nie da się tak naprawdę poprawić jakości inwestycji w infrastrukturę kolejową.

Dziękuję bardzo, pani marszałek. Generalnie oceniamy ten projekt jako bardzo ciekawy.

Bardzo proszę, pan poseł Michał Urbaniak, Koło Poselskie Konfederacja.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mówimy teraz o druku nr 43 dotyczącym ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym i innych ustaw. Koło Konfederacji z uwagą przyjrzało się temu projektowi.

To jest słuszna linia, żeby jednak to upraszczać i regulować.

Problemy te także wymagają pilnego rozwiązania i w tym zakresie zasługują na uwzględnienie.

Otóż dostrzegamy naturalnie plusy tego projektu, m.in. właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, deregulację. Dostrzegamy też potrzebę upraszczania procedur dotyczących tworzenia linii pomiędzy województwami, jednak zapis, który mówi o tym, że połączenia wojewódzkie będą mogły być wyprowadzane tylko 30 km od granicy danego województwa, uważamy za niewystarczający. Przykładem niech będą linie dotyczące Kutna i Torunia czy np. Głogowa i Leszna. Dziękuję bardzo, panie pośle. Czy ktoś z pań i panów posłów chce jeszcze zgłosić się do zadania pytania? Jako pierwszy pytanie zadaje pan poseł Tadeusz Tomaszewski, klub Lewica. Minuta na zadanie pytania. Wysoki Sejmie! Szanowny Panie Ministrze! W ramach remontu linii kolejowej Poznań - Warszawa oddano do użytku nowe perony, a obecnie trwa przebudowa przejść podziemnych w Koninie. Mieszkańcy Konina i władze samorządowe od blisko 2 lat czekają na rozpoczęcie budowy dworca PKP jako elementu zintegrowanego centrum komunikacyjno-handlowego. W związku z tym pytanie: Dlaczego tak długo trwa proces rozpoczęcia budowy dworca PKP w Koninie? Kiedy przewiduje się rozpoczęcie tej inwestycji? Drugie pytanie dotyczy tego, czy w programie „Kolej+” do 2028 r. przewiduje się środki na uruchomienie linii kolejowej Śrem - Czempiń. To jest linia nr 369, która została otwarta tak a propos w 1885 r.

Dziękuję. Bardzo proszę, pan poseł Wiesław Szczepański, klub Lewica. Panie Ministrze! Modernizacja linii kolejowej nr 271, która miała być zakończona na Euro 2012, jest dzisiaj opóźniona. Mam pytanie: Kiedy zostanie rzeczywiście ukończony odcinek od Czempinia do granicy województwa wielkopolskiego? Czy zamierzacie państwo po ukończeniu tej linii uruchomić ponownie pociąg bezpośredni przez Leszno do Warszawy? To ułatwiłoby połączenia komunikacyjne dla mieszkańców województwa dolnośląskiego, powiem np. o Głogowie, czy też województwa lubuskiego. Czy w świetle ustawy przewidywane jest przywrócenie linii kolejowej Leszno - Gostyń i elektryfikacja linii kolejowej z Krotoszyna do Głogowa? Ile gruntów zbędnych PKP, myślę o bocznicach, liniach kolejowych, przekazano do Krajowego Zasobu Nieruchomości lub zbyto na rzecz PFR-u? Mówię tu o oficjalnym zbyciu, a nie o toczących się negocjacjach, dlatego że według mojej wiedzy dzisiaj udział PKP w programie „Mieszkanie+” jest jednak fikcją, a ta ustawa, panie ministrze, jeszcze bardziej ograniczy po prostu tej spółce przekazywanie gruntów na rzecz KZN. Bardzo proszę, pan poseł Romuald Ajchler, klub Lewica. Wysoka Izbo! W VII kadencji zabiegałem o to, aby reaktywować linię kolejową nr 368 z Międzychodu do Szamotuł.

Bardzo o to bym prosił pana ministra.

Ile mamy do dzisiaj wykorzystanych środków?

Panie Premierze! Wysoka Izbo!

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Jan Szopiński, klub Lewica. Wysoka Izbo!

To powoduje frustrację mieszkańców Kcyni i całego powiatu, którzy nie są w stanie zrozumieć, że muszą dojeżdżać samochodem do Gołańcza, aby pociągiem dotrzeć do Poznania, gdzie studiuje bardzo wiele młodzieży. Czy nastąpi skomunikowanie miejscowości Kcynia i Nakło, co dałoby szansę na rozwój tej części województwa? Jakie są perspektywy dla linii kolejowej nr 241, łączącej Koronowo z Tucholą? Czy przewiduje się budowę połączenia Maksymilianowo - Koronowo? Kiedy zacznie się realizacja tego zadania? Panie Ministrze! Ostatnie pytanie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Zdzisław Wolski, klub Lewica. Kiedyś bardzo ważną linią była linia warszawsko-wiedeńska. Ważną stacją była Częstochowa. Pewnie trzeba je chronić.

Od lat nie wiadomo, co z tym dworcem. Będzie wyburzony? Nie będzie? Trwają prace SARP nad koncepcją architektoniczną. Mam pytanie do pana ministra. Kiedy będzie nowy dworzec? Wszystko wskazuje, że należałoby łącznie z PKS (Dzwonek), również państwowym, coś bardzo fajnego wymyślić. Dziękuję bardzo. Pan poseł Maciej Konieczny, klub Lewica. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Lewica stawia na kolej.

Sytuacja, w której rząd ma pieniądze na ekspresowe połączenie z Baranowa do Ostrawy, a takie miasta jak chociażby Jastrzębie-Zdrój do dzisiaj pozbawione są kolei, jest absurdalna. Stąd moje pytanie: Czy rząd przewiduje, i w jakim zakresie, finansowanie z budżetu centralnego projektu rozwoju kolei metropolitalnej w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii? Przypominam, że na takie centralne finansowanie mogło liczyć warszawskie metro. Zakładam, że największa aglomeracja w tym kraju może liczyć na przynajmniej równie dobre traktowanie. Proszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani poseł Daria Gosek-Popiołek, klub Lewica. Nie ma pani poseł. Pan poseł Tomasz Piotr Nowak, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Czy w świetle tej ustawy, kiedy samorządy inwestują w infrastrukturę kolejową, Fundusz Dróg Samorządowych będzie mógł być tym instrumentem, który pomoże w realizacji bardzo dużych inwestycji? Proszę sobie wyobrazić, że w Koninie powstaje wiadukt, który jest częścią modernizowanej trasy Berlin - Moskwa.

Miasto musi się zadłużyć, wziąć stosowne obligacje, ażeby zrealizować projekt, który tak naprawdę jest projektem infrastrukturalnym w ramach bardzo ważnej trasy międzynarodowej.

Bardzo liczę (Dzwonek), że te 30 mln stanie się rzeczywistością. Bardzo proszę, pan poseł Krzysztof Gadowski, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! które do dzisiaj nie ma przewozów kolei pasażerskiej. Oczywiście odjeżdżają pociągi z węglem. Nie ma z tym problemów. Te tory są utrzymywane przez spółkę węglową. Natomiast od kilkunastu lat brakuje przewozów pasażerskich. Wielokrotnie tu, z tej trybuny sejmowej, pytałem ministra, na jakim etapie są przygotowania i czy w ogóle są. Mamy nową panią prezydent, która przygotowała już wstępne studium techniczno-ekonomiczne. Panie Ministrze! Chciałbym dzisiaj wiedzieć, czy pan będzie realizował tę kolej pasażerską do Jastrzębia, skoro niedawno z tej trybuny pan premier Morawiecki wyraźnie mówił, że te miasta, które dzisiaj nie mają kolei, będą ją miały. Proszę o odpowiedź na piśmie. Bardzo proszę, pani poseł Paulina Matysiak, Lewica. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chciałabym zwrócić uwagę na dwie kwestie, które pojawiają się w tym projekcie.

I druga sprawa to tak naprawdę nieszczęsny zapis o limicie odległości 30 km od granicy województwa.

Pani poseł Wanda Nowicka, klub Lewica. Szanowna Pani Marszałkini! Panie Ministrze! Kolej i tramwaje to najbardziej zielona, najbardziej ekologiczna forma transportu, a więc rozwój transportu publicznego, zwłaszcza kolei, to także inwestycja w czyste powietrze i w nasze zdrowie. Nie stać nas na odkładanie tego na później. Jednak żeby ludzie realnie przesiedli się z samochodów na kolej, to musi ona dojeżdżać także do mniejszych miejscowości, i to dojeżdżać często. Jest to szczególnie ważne w okręgu gliwickim z uwagi na wysokie stężenie smogu. Dlatego pytam: Kiedy plany inwestycji przedłużenia linii S1 do Pyskowic oraz kolei miejskiej w Knurowie i Gierałtowicach zostaną zrealizowane? Dzięki temu mieszkańcy tych miejscowości będą mogli szybko i wygodnie dojechać do pracy bez konieczności wsiadania do samochodu, a my wszyscy skorzystamy z czystego powietrza i mniejszych korków. Gdyby pan minister nie odpowiedział na to pytanie podczas debaty, bardzo proszę o odpowiedź na piśmie. Bardzo proszę, pan poseł Mirosław Suchoń, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Panie ministrze, oczywiście papier, tak jak mówiłem, cierpliwy jest i wszystko przyjmie, natomiast te szczytne założenia, które zapewne panem kierowały, kiedy ministerstwo przygotowywało projekt ustawy, nijak się mają do rzeczywistości. Bo weźmy choćby linię nr 190 na odcinku Bielsko-Biała - Skoczów. Ta linia jest nieczynna od wielu lat, nie jeżdżą tam pociągi, a teraz państwo podejmują decyzję o rewitalizacji drugiej części tej linii, czyli gdzieś tam Skoczów - Cieszyn, Bronowice - Wisła, i pozostawiają państwo bez rewitalizacji kluczowy odcinek właśnie dla tego połączenia Bielsko-Biała - Skoczów.

Te pieniądze są po prostu wyrzucone w błoto i te działania nie będą miały pozytywnych skutków dla wszystkich mieszkańców całego regionu. Bardzo proszę, pan poseł Robert Kwiatkowski, klub Lewica. Bardzo dziękuję. Panie Ministrze! Zwracam się z prośbą o informację na temat sytuacji dworca w Grudziądzu. Szef PKP nawet zwołał konferencję prasową na ten temat.

Zresztą nie chcę opowiadać już o tym, jak ważne są dworce w życiu naszego społeczeństwa. Lista pytań, które klub Lewicy przedstawia, jest tego wystarczającym dowodem. Tak że prosiłbym o informację na temat tego, kiedy dworzec w Grudziądzu zostanie oddany. Drugie pytanie dotyczy przyszłości czy elektryfikacji linii nr 207 na odcinku między Grudziądzem a Toruniem. Trzecie pytanie, które już się tutaj pojawiało (Dzwonek), dotyczy odcinka Kowalewo Pomorskie - Brodnica.

Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Nie jestem w stanie powiedzieć panu o tym, że pendolino musi dojeżdżać do Szczecina, a nie dojeżdża, i musi dojeżdżać do Świnoujścia, a nie dojeżdża. Nie jestem w stanie panu powiedzieć o tym, że linia Goleniów - Kołobrzeg musi być zelektryfikowana, a nie jest.

Mam w takim razie jedno pytanie, panie ministrze, jedno pytanie od posła opozycji: Czy byłby pan tak uprzejmy zaprosić posła opozycji do siebie na pół godziny? Ja to wszystko panu wytłumaczę i zadam pytania. Dziękuję bardzo. Proszę, pan poseł Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15. Panie Ministrze! Ważnym punktem tej noweli jest sprawa dotycząca użyczenia terenów i dróg kolejowych również samorządom.

I teraz jest pytanie: Które samorządy będą mogły się o to ubiegać? Druga kwestia, która jest z tym związana, to jest kwestia podatków, jeżeli chodzi o te nieczynne linie kolejowe, a w szczególności obiektów towarzyszących, jak również kwestia remontów, np. obiektów inżynierskich, np. wiaduktów. To jest bardzo trudny problem dla tych samorządów, które chciałyby, aby to materialne dziedzictwo pozostało na tym terenie i było jakoś wykorzystywane. Druga sprawa to jest kwestia remontu, modernizacji dworca w Lesznie przy modernizowanej trasie Wrocław - Poznań. W tej sprawie otrzymuję sporo pytań ze strony mieszkańców Leszna (Dzwonek) i Wielkopolski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Dariusz Wieczorek, klub Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przecież prawda jest taka, że jeżeli chodzi o wydatki PLK, w roku 2018 miano wydać 11 mld, wydano zaledwie 10, w związku z czym widać wyraźnie, że ta ustawa jest absolutnie potrzebna. Rzecz druga. Co jest z kwestią związaną z infrastrukturą, a więc PKP Energetyka, zasilaniem nowych czy odtworzonych linii kolejowych? Bo możemy budować linię kolejową, ale do niej trzeba jednak mieć infrastrukturę energetyczną. Trzecia sprawa to jest pytanie, na które prosiłbym o odpowiedź na piśmie. To jest kwestia linii nadodrzańskiej, linii 273, o którą, mówię jako poseł i samorządowiec Zachodniopomorskiego, zabiegamy od wielu, wielu lat. Pytanie: Na jakim etapie jest realizacja tej inwestycji i czy ta ustawa wpłynie na to, że ta inwestycja będzie (Dzwonek) realizowana szybciej? Bardzo proszę, pani poseł Urszula Nowogórska, Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15. Wysoka Izbo! Reprezentuję Małopolskę, obszar piękny, aczkolwiek trudny w dostępie. Jest wiele białych plam, które stanowią tzw. utrudnienia komunikacyjne na terenie naszego regionu. Intencja sama w sobie jest bardzo słuszna, natomiast powstaje pytanie. Chodzi o przekazanie, dobrowolne użyczenie samorządom tych obszarów, które są mocno zdegradowane i zniszczone. To się wiąże z bardzo poważnymi wydatkami finansowymi, choć samorządy są do tego przyzwyczajone i mają wprawę w wydatkowaniu tych pieniędzy. Moje pytanie: Czy za przekazaniem pójdzie finansowanie i czy w momencie kiedy to finansowanie się pojawi albo nie pojawi i kiedy samorządy dokonają modernizacji tych obszarów kolejowych, rzeczywiście potem te obszary nie powrócą do właścicieli, od których pierwotnie pochodzą? To znacznie utrudniłoby działania i, myślę, znacznie ograniczyłoby również wszystkie te inwestycje, które samorządy, również wojewódzkie, realizują ze swoich budżetów, a w tym momencie byłyby bardzo mocno ograniczone. Jak te inwestycje mogłyby się wpisywać w plany rozwoju np. powstałej zaprojektowanej linii Piekiełko - Podłęże na terenie województwa małopolskiego? Czy to nie pokrywałoby się, jeżeli chodzi o samo inwestowanie, działanie, obszar i oddziaływanie? Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam pytanie, bo mówimy tutaj tyle o przekazywaniu gruntów. Jednym wielkim problemem dla miasta Inowrocław, leżącego w województwie kujawsko-pomorskim, z którego pochodzę, jest teren pod ul. Magazynową. Ten teren miał być modernizowany, przebudowywany ze środków także urzędu marszałkowskiego, w którym do niedawna też pracowałem. Niestety od 4 lat jest opór ze strony PKP, jeżeli chodzi o przekazanie tego gruntu. Jest duży problem, aby ten grunt uzyskało miasto Inowrocław. Zapewnione środki, które były przekazane przez urząd marszałkowski, już w tej chwili zapewne nie wystarczą na tę inwestycję, bo jej koszt z 8 mln zwiększył się, poprzez zwyżkę cen na rynku, do 28 mln. Oczekuję odpowiedzi na piśmie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o przekazanie tego gruntu i o przyspieszenie przekazania gruntu pod ul. Magazynową w mieście Inowrocław. Bardzo proszę, pani poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, klub Lewica. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Moje pytanie jest proste: Czy zdarza się panu podróżować koleją? Jeśli tak, czy jeździ pan nocą? Proszę państwa, mamy taką sytuację, że państwo polskie rezygnuje z wagonów, które mają kuszetki, i wagonów sypialnych. Bardzo nad tym boleję.

I wiecie państwo, co się dzieje?

Dziękuję za te oklaski, panie pośle. To jest może na marginesie tego, [[Oklaski]] co jest dzisiaj szalenie ważne, ale bardzo proszę, żeby państwo się tym zajęło. To jest dla nas wszystkich szalenie ważne. Dziękuję bardzo. Proszę, pan poseł Andrzej Gawron, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Dziękuję za tę ustawę, bo to bardzo dobry ruch, jeżeli chodzi o nowelizację ustawy o transporcie kolejowym. Na pewno przez takie działanie zmniejszymy wykluczenie komunikacyjne. Mnie szczególnie interesuje możliwość wsparcia przewozów osobowych na granicach województw. To jest dosyć istotna sprawa. Są np. miejscowości w różnych województwach i rzeczywiście jest problem, żeby te miejscowości skomunikować.

Tak że proszę, panie ministrze, uszczegółowić to i powiedzieć dokładnie, jakie wsparcie będzie tutaj przewidziane w nowelizacji ustawy, jakie będą formy tego wsparcia, jeżeli chodzi właśnie o przewozy między województwami.

Bardzo proszę, pan poseł Przemysław Koperski, klub Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze!

Mieszkańcy wspierani przez liczne samorządy czekają od kilkunastu lat na przywrócenie tego połączenia kolejowego, umożliwiającego dotarcie do szkoły czy pracy dziesiątkom tysięcy osób.

Dzisiaj jest dla kolejnych rządów powodem do wstydu. Panie ministrze, czy ta zmiana ustawy pozwoli w tej kadencji Sejmu w końcu zrewitalizować skutecznie linię kolejową 190 Bielsko-Biała - Skoczów - Cieszyn? Dziękuję uprzejmie. Pani poseł Joanna Fabisiak, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Świadczą o tym liczby: 4 mln odwiedzających rocznie albo i więcej, w czasie weekendu 250 tys. O tym, że trzeba mieć dużo hartu ducha i dobre zdrowie, żeby dojechać do Zakopanego, świadczą znów liczby. O tym, że zakopianka stoi - czasami z Zakopanego do Krakowa jedzie się 6 godzin - też pewnie państwo słyszeliście z mediów. Dlaczego ludzie nie jeżdżą pociągami? Ano dlatego, że od 2016 r. trwa - jak mówią strony PKP - modernizacja tej trasy. Ale ludzie chcą jeździć, ludzie chcą uprawiać sporty, ludzie chcą być w Zakopanem. Dlaczego wobec tego muszą jeździć busikami, które są nie najgorsze, ale wyobraźcie sobie, jak straszliwie te tysiące busików zatruwają środowisko? Wobec tego zwracam się z ogromnym apelem i z pytaniem do państwa: Jak ten problem będzie rozwiązany i kiedy? Bo minęły 3 lata, a modernizacja trwa nadal. To jest jeden pociąg.

Dziękuję bardzo, pani poseł. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Chciałam zapytać o linię kolejową Jelenia Góra - Lwówek Śląski. Linia kolejowa została zlikwidowana, ruch na tej linii został zlikwidowany w 2017 r., a więc za tego rządu. Ta linia przebiega przez obszar wykluczony komunikacyjnie. Młodzież szkolna ma bardzo duże problemy z dojazdem do szkół w Jeleniej Górze. Takie miasteczka jak Lwówek Śląski, Wleń są po prostu odcięte od Jeleniej Góry.

Mieszkańcy wielokrotnie o to pytali. Co dalej z tą linią? Kiedy zdecydujecie się, czy otrzyma ją marszałek, czy rząd będzie ją remontował? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Jerzy Paul, klub Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Pan minister przedstawił nam cały pakiet propozycji zmian ustaw dotyczących ruchu szynowego. Zdajemy sobie sprawę, że inwestycje na torach są bardzo drogie i bez wsparcia Unii Europejskiej po prostu niemożliwe do wykonania. Ale obserwując poczynania rządu Donalda Tuska, wszyscy zgadzają się z tym, że te inwestycje były ciągle opóźniane i Polska musiała liczyć się ze zwrotem niewykorzystanych funduszy unijnych. Dlatego moje pytanie brzmi: Czy proponowana zmiana przepisów wpłynie pozytywnie na wydatkowanie środków unijnych związanych ściśle z inwestycjami przeprowadzanymi na torach kolejowych i tramwajowych i czy te nowe przepisy nie będą opóźniały procesu inwestycyjnego związanego z ruchem szynowym? Pan poseł Ryszard Bartosik, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Ministrze! Przede wszystkim chciałbym podziękować za to, że taki projekt ustawy powstał. Za to, że wreszcie została zahamowana likwidacja połączeń kolejowych, jak to miało miejsce przez całe lata 90. i za rządów Platformy Obywatelskiej oraz PSL-u. Chciałbym także podziękować za to, że dzięki temu projektowi taka miejscowość jak Turek w Wielkopolsce, region, który reprezentuję, będzie miała szansę na połączenie z Koninem, i za to, że w projekcie „Kolej+” miasto Turek znalazło się i ma szansę na nowe połączenie, którego dotychczas nie miało.

Będzie to duże obciążenie, mimo że jest to 15% dla samorządów. Proszę, pani poseł Karolina Pawliczak, klub Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Tak istotne, ważne i planowane przecież od lat. Przypomnę krótką historię. W 1993 r. pierwsze studialne przymiarki Dyrekcji Generalnej PKP. W 2005 r. za rządów Sojuszu Lewicy Demokratycznej pojawiły się pierwsze przygotowania dotyczące wstępnego studium w Instytucie Kolejnictwa, a w 2011 r. przeprowadzono konsultacje społeczne. Pytam, panie ministrze, jak dziś wygląda program kolei dużych prędkości, czy został on zarzucony i jak wygląda sprawa stacji przesiadkowych na terenie byłego już województwa kaliskiego. Proszę, pan poseł Janusz Korwin-Mikke, Konfederacja. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam cztery pytania. 35 lat temu byliśmy 30 lat przed Chinami, dzięki Niemcom oczywiście, a w tej chwili jesteśmy 10 lat za Chinami. Chiny już budują, ponieważ nie weszły do Unii Europejskiej i dlatego mają szybkie koleje. Mam jeszcze pytania: Ile kilometrów miesięcznie budował w XIX w. Jake Gold w Ameryce? Proszę nie mówić, że im było łatwiej, bo wtedy mierzono we wiorstach, w milach i w li. Dziękuję za uwagę. Bardzo proszę, pan poseł Jacek Tomczak, Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15.

Wysoka Izbo! Chciałbym zadać trzy pytania. Pierwsze będzie dotyczyło realizacji inwestycji przez PKP PLK. Chciałem zadać pytanie: Jaki jest obecny poziom realizacji inwestycji przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej? Jakie są zagrożenia dla wykorzystania tych środków Unii Europejskiej, ponieważ mamy niepokojące informacje, że ponad połowa tych inwestycji jest opóźniona lub

Chciałbym zapytać: Kiedy wreszcie ruszy budowa nowego dworca w Koninie? Bardzo proszę, pani poseł Klaudia Jachira, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zawsze z wielką przyjemnością przyjmuję takie wiadomości, że rząd chce zadbać wreszcie o kolej, o transport publiczny. Natomiast mam pytanie do rządu: Kiedy zamierza przesiąść się z tych swoich drogich, czarnych, ciemnych, z przyciemnianymi szybami limuzyn właśnie na transport publiczny, właśnie na kolej? Z tych limuzyn, które są opłacane z pieniędzy podatników, z tych limuzyn, które już wielokrotnie rozbijaliście. Może wtedy, gdy przesiądziecie się właśnie z tych limuzyn na kolej, na transport publiczny, zrozumiecie, że nie jest on idealny, że jest dużo do naprawienia.

Bardzo zachęcam i pytam: Kiedy rząd zamierza zacząć jeździć koleją (Dzwonek) i transportem publicznym? Zachęcam. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Czesław Mroczek, Koalicja Obywatelska. Niezwykle ważne są wszystkie działania podejmowane w celu usprawnienia transportu kolejowego.

Mianowicie budowa bezkolizyjnych przejazdów przez tory kolejowe i dworce kolejowe. Jeżeli chodzi o pierwszą sprawę, bezkolizyjne przejazdy przez tory kolejowe, to dla mnie takim symbolem nieporadności w tym zakresie jest miejscowość Mrozy. Miasto, gdzie w pozwoleniu na budowę w zakresie przebudowy linii kolejowej Moskwa - Berlin wpisano budowę dworca bezkolizyjnego przejazdu (Dzwonek) przez tory i do dzisiaj to nie zostało zrealizowane. To jest skala porażki państwa, że linie zmodernizowano, inspektorat kolejowy wpisał potrzebę wybudowania wiaduktu bezkolizyjnego, a do dzisiaj go nie zbudowano. W tym zakresie rząd powinien ustanowić specjalny program. Tak jak był program Orlików, tak musi być program związany z budową bezkolizyjnych. Bardzo proszę, pan poseł Paweł Krutul, klub Lewica. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Ciągle trwa debata mieszkańców Białegostoku i okolic na temat wyprowadzenia z centrum miast tranzytu kolejowego. Mieliśmy takie zdarzenie kilkanaście lat temu, że jedna z cystern z chlorem właśnie wybuchła w centrum Białegostoku. Było to bardzo, bardzo, ale to bardzo niebezpieczne zdarzenie. Proszę o jak najszybsze przedstawienie przez PKP PLK wariantów przebiegu tej inwestycji w konsultacji z mieszkańcami Białegostoku i okolic. Jest to bardzo istotna sprawa dla mieszkańców województwa podlaskiego. Proszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję bardzo. Ostatnie pytanie zadaje pani poseł Daria Gosek-Popiołek, klub Lewica. Szanowna Izbo! Dwie sprawy. Skoro przedstawiona ustawa ma na celu powstrzymanie likwidacji linii kolejowych, to dlaczego w jednym z artykułów dopuszcza ona całkowitą tych likwidację linii? Cytuję: Grunty pozostałe po zlikwidowanych liniach kolejowych lub bocznicach kolejowych wraz z zabudowaną infrastrukturą mogą być przekazane w użyczenie jednostkom samorządu terytorialnego na cele transportowe. Co to oznacza? To oznacza, że tych zamkniętych już linii kolejowych nie będzie można przywrócić do użytkowania. Dlaczego? Bo na ich miejscu będzie można wybudować obwodnice, drogi i ścieżki rowerowe. I to nie są przykłady z głowy, dlatego że mamy w Polsce kilka miast, w których istniejące tory, linie kolejowe zostały zamienione na obwodnice, np. Barlinek czy Mrzygłód. To jest zły kierunek. Bardzo proszę o to, abyście państwo po prostu to zmienili i dopisali jedno słowo: na cele transportowe kolejowe albo szynowe. Jedno słowo, a rzeczywiście uniemożliwi niszczenie linii. I druga sprawa, chciałabym zaapelować o szybsze rozwiązanie kwestii transportu kolejowego pomiędzy Krakowem a Olsztynem... przepraszam, Olkuszem. To było ostatnie pytanie. Proszę sekretarza w Ministerstwie Infrastruktury pana ministra Andrzeja Bittela o udzielenie odpowiedzi na pytania.

Wysoka Izbo! Jestem niezwykle rad, że ten projekt ustawy spotkał się z tak żywym odzewem, choć mam też nieodparte wrażenie, że wiele pytań nadaje się bardziej na interpelację niż dotyczy tego przedłożenia.

Cieszy mnie niezwykle zainteresowanie czy niezwykle duży udział w tej debacie przedstawicieli klubu Lewica. Jestem niezwykle z tego rad, szczególnie cieszę się z udziału w debacie pana posła Szczepańskiego, który był ministrem, wiceministrem infrastruktury w dwóch rządach, podczas których zostały. Wydaje mi się, że w dwóch.

Z tego się tym bardziej cieszę, bo to oznacza, że mamy wspólny cel. Tym celem wspólnym jest odbudowanie polskiej kolei, jest jej finansowanie, jest realizowanie programów inwestycyjnych takich jak „Krajowy program kolejowy”, który stanowi niezwykle istotny instrument interwencji w zakresie głównych korytarzy transportowych, który jest finansowany z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”, który jest finansowany z Programu „Łącząc Europę” Jesteśmy liderem w pozyskiwaniu środków europejskich na linie kolejowe, na modernizację linii kolejowych, jesteśmy liderem w wykorzystywaniu tych środków. Myślę, że to państwo powinni dostrzec z całą pewnością, bo poziomy wykorzystania środków związanych z koleją, modernizacją kolei, jeśli porównać rok obecnej perspektywy do roku poprzedniej perspektywy, to są w ogóle zupełnie dwa światy.

Jesteśmy niezwykle zaawansowani w tych działaniach. O tym należy pamiętać i należy też pamiętać o programie utrzymaniowym, który został uchwalony.

Trzeba też powiedzieć, że na każdym poziomie administracji publicznej są pewne obowiązki, tak jak obowiązkiem rządu jest organizowanie połączeń międzywojewódzkich i transgranicznych, tak obowiązkiem samorządu wojewódzkiego jest organizowanie połączeń regionalnych.

Samorząd województwa wskazuje swoje priorytety, oczywiście w uzgodnieniu z beneficjentem, jakim jest PKP Polskie Linie Kolejowe.

Dlaczego wprowadzamy element użyczenia do porządku prawnego dla samorządu terytorialnego? Wprowadzamy to nie po to, żeby przerzucać jakieś obowiązki, tylko po to, żeby dać samorządowi możliwość czasowego, w krótszej perspektywie, w dłuższej, bo przecież proces przywracania połączeń kolejowych to nie jest proces o, taki. Likwiduje się łatwo: wydaje się decyzję, najpierw wygasza się popyt, potem wygasza się linię kolejową od strony przewoźnika, a następnie wydaje się decyzję o likwidacji, bo jak nic nie jeździ, to nie ma się interesu ekonomicznego w tym, żeby taką linię utrzymywać. I wygasza się łatwo: tutaj decyzja, tam decyzja. Żadna tego typu decyzja nie zapadła w poprzedniej kadencji. Jeśli pan poseł mówi o likwidacji linii kolejowej, to mówi o rozbiórce dawno zlikwidowanej linii kolejowej. Pytanie jest - i tu się pewnie różnimy - czy warto jest pozostawić na gruncie wyeksploatowane tory kolejowe, które powoli, powoli lokalny biznes, oczywiście mówiąc w cudzysłowie, rozbierze i zaniesie do skupu złomu, czy należy to samemu zebrać, uzyskać z tego jakiś przychód, niewielki, bo niewielki, ale jednak to jest nasz wspólny majątek, a utrzymać korytarz z punktu widzenia nieruchomości, bo to jest podstawowa bariera, jeśli chodzi o odtwarzanie linii kolejowej, to jest najważniejsza kwestia, żeby był korytarz. Jeżeli ktoś podjął decyzję, żeby korytarz kolejowy przeciąć autostradą, to jak go utrzymać? Potem w konsekwencji są decyzje o jakimś innym sposobie zagospodarowania tego korytarza.

Ta ustawa ma również na celu porządkowanie relacji z samorządem w kontekstach wiaduktowych czy przejazdów przez tory kolejowe, które były realizowane w ramach inwestycji, po to aby sobie powiedzieć jasno, kto za co odpowiada.

Oczywiście tak.

i konsekwentnie będziemy współpracowali, choć ten problem nie jest opisany w tej ustawie, jest w innej ustawie, już przyjętej.

A więc to jest skala tego przedsięwzięcia, które będziemy realizowali. Część tych pieniędzy, tych 11 mld, mniej więcej połowa, jest już uwzględniona w „Krajowym programie kolejowym”, który realizujemy, który też przyczynia się do likwidowania wykluczenia komunikacyjnego, który przyczynia się do tego, aby szlaki kolejowe w ramach TEN-T były takie, jak oczekuje od nas Komisja Europejska, w określonym czasie, a tym określonym czasem jest rok 2030, o odpowiednich parametrach.

Czy ta ustawa jest za późno? W mojej ocenie oczywiście można było wiele rzeczy zrobić wcześniej. Można było nie likwidować wcześniej linii kolejowej.

Ja się z tego bardzo, bardzo cieszę. Ustawa była w konsultacjach, ustawa była opiniowana przez KWRiST. Oczywiście ktoś w którymś momencie musi zdecydować, czy 30 km, czy 50 km, czy 70 km. Jeżeli będzie potrzeba zmiany tego parametru, to jesteśmy otwarci na dyskusję czy teraz, czy potem, jak już te przepisy zafunkcjonują i sprawdzimy, jak one działają, bo to przewoźnicy powinni w określonym czasie przedstawić taką swoją ofertę, że chcieliby zrobić swoją ofertę w innym kształcie, i wtedy będziemy się nad tym z całą pewnością pochylali.

Mogę powiedzieć, że przepisy prawa, które w tej chwili obowiązują, a zostały one zmienione w ostatnich 2 latach, pozwalają na budowę linii kolejowych do prędkości 250 km/h. Geometria pewnie przy nowych liniach kolejowych i przy liniach kolejowych modernizowanych będzie na to pozwalała, ale patrząc przez pryzmat potrzeb, trzeba się zastanowić, czy dla naszego państwa 300 km to jest wystarczająco czy za dużo.

To jest ten cel, który jest opisany na dzisiaj. Tempo budowy jest oczywiście uzależnione od tego, jakie mamy przepisy prawa, czy poprawimy mechanizację na placach budów. Czy będziemy mogli namówić naszych wykonawców na to, pokazując im długą perspektywę inwestowania w polską kolej, przekonać, że warto się modernizować, jeśli chodzi o sprzęt, jeśli chodzi o te wszystkie środki techniczne, które by pozwalały procesy budowlane automatyzować i dzięki temu je przyspieszać i jednocześnie nadawać im jeszcze wyższy poziom jakości. Jeśli nie odpowiedziałem na jakieś pytanie szczegółowe, to oczywiście przygotujemy odpowiedź na piśmie. Chciałbym uniknąć dyskusji, w której na podstawie tych przepisów będziemy dyskutowali, w którym roku który dworzec zostanie zbudowany. My ten plan mamy. To jest pierwszy tak duży program dworcowy, który realizujemy. Jeśli chodzi o zaproszenie, to oczywiście jestem gotów się spotykać z każdym posłem, a nawet powiem, że mam taki obowiązek, który wynika z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Panie Ministrze! Jeśli pan studiował mój życiorys, to zapomniał pan powiedzieć, że byłem wiceministrem infrastruktury, ale od spraw budownictwa, a nie od spraw kolei.

Zamykam dyskusję. Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, zawarty w druku nr 43, do Komisji Infrastruktury w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę.

Proszę pana posła Marka Suskiego o przedstawienie uzasadnienia projektu. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy Prawo celne, druk nr 51. Szanowni Państwo. Ta ustawa jest, można powiedzieć, bardzo krótka, aczkolwiek istotna, ponieważ wprowadza zmiany do Prawa celnego oraz ustawy o podatku akcyzowym od wyrobów, które są zwolnione z tego podatku. Głównie chodzi tutaj o paliwa, o dostarczenie paliw lotniczych czy paliw żeglugowych albo do przemysłu chemicznego na rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, zmywacze do farb. Ta ustawa wydłuża okres, w którym przedsiębiorcy będą musieli dostosować swoje wykazania przemieszczania się tych wyrobów, chodzi o rezygnację, przejście z papierowej dokumentacji na dokumentację elektroniczną. Co to oznacza? To oznacza, że podmioty będą dysponowały dodatkowym czasem na wdrożenie systemu pozwalającego na przejście z papierowego dokumentu dostawy na system elektroniczny.

To umożliwi zainstalowanie nowego oprogramowania, czyli jest to ułatwienie dla przedsiębiorców. Chodzi o takie płynne przejście z systemu papierowego na system elektroniczny, który pasuje też do paliw płynnych. Szanowni Państwo!

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. Unia Europejska zresztą tego zagadnienia nie reguluje.

Nie ma tutaj również norm technicznych, które by powodowały, że ustawę należałoby notyfikować, a zatem ustawa nie podlega notyfikacji.

Dziękuję bardzo. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Jerzy Materna, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawić stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz Celem nowelizacji ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz Prawo celne jest wprowadzenie dodatkowego, 13-miesięcznego vacatio legis umożliwiającego stosowanie papierowego dokumentu dostawy w systemie EMCS PL 2 i elektronicznego dokumentu dostawy.

Przedłużenie stosowania papierowego dokumentu dostawy nie ma wpływu na zwiększenie wydatków po stronie przedsiębiorców. Projekt ustawy nie ma wpływu na sektor finansów publicznych. Projekt ustawy nie wpłynie na zwiększenie wydatków i zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość chciałbym wnieść poprawkę do projektu ustawy.

Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość popiera projekt ustawy i będzie głosować za jego przyjęciem. Dziękuję. Nie może pan zgłosić teraz poprawki. Poprawkę można zgłosić w drugim czytaniu, więc musi pan zabrać tę poprawkę i jak będzie drugie czytanie, ją zgłosić. To nie jest drugie czytanie. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko naszego klubu wobec projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy Prawo celne. W pierwszej kolejności chcę się odnieść do słów posła wnioskodawcy Marka Suskiego, który powiedział na zakończenie swojego wystąpienia, że ta ustawa jest dobra dla polskiej gospodarki. Chcę, panie pośle, panu uświadomić, że ta ustawa z dobrem polskiej gospodarki nie ma absolutnie nic wspólnego. Ta ustawa ma za to wiele wspólnego z niechlujstwem legislacyjnym, które obowiązuje w tym parlamencie za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Właściwie może nie posłowie PiS-u, tylko nie pamiętało o tym w ogóle Ministerstwo Finansów, które tak naprawdę skupiło się wyłącznie na tym, aby podnieść akcyzę o 10% na alkohol, na wyroby tytoniowe, aby zabezpieczyć wpływ do budżetu, potencjalny wpływ do budżetu państwa w wysokości 1700 mln zł.

Senatorowie ten problem wychwycili i nawet podjęli inicjatywę legislacyjną na poziomie Senatu, niemal tożsamą z przedłożeniem, które później wpłynęło do Sejmu. Oczywiście jako klub Koalicji Obywatelskiej będziemy za tym projektem ustawy, bo to jest naturalne. Oczywiście poprzemy te przepisy, żeby ten obrót papierowy dokumentacji był możliwy jeszcze przez kolejny rok, ale tak jak powiedziałem, państwo musicie się zastanowić, bo funkcjonowanie państwa pod waszymi rządami to jeden wielki chaos, a tak naprawdę prestiż bycia parlamentarzystą nie powinien nam pozwalać, aby tak funkcjonować. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Wiesław Szczepański, Lewica. Pani Marszałek! W imieniu klubu parlamentarnego Lewica mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy z dnia 5 grudnia br. zmieniającego ustawę o podatku akcyzowym oraz ustawę Prawo celne, zawartego w druku nr 51.

Jak już mówił mój przedmówca, znów o rok wydłużamy termin wejścia w życie kolejnej ustawy. Ustawą z lipca 2018 r. zmieniającą ustawę o podatku akcyzowym oraz Prawo celne wprowadzono stosowanie systemu EMCS PL2 i elektronicznego dokumentu dostawy eDD do pomieszczeń na terytorium kraju poza procedurą zawieszania poboru akcyzy od wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy z uwagi na ich przeznaczenie.

Jednocześnie w 2019 r. zmieniono ustawę i postanowiono, że do dokumentów dostawy wystawionych przed dniem 1 stycznia 2020 r. stosuje się przepisy art. 138 zmienionej ustawy w brzmieniu dotychczasowym, a więc dokumentację papierową.

To komputerowy system wykorzystywany do przemieszczania wyrobów akcyzowych, wyrobów energetycznych, alkoholowych, tytoniowych w procedurze zawieszania poboru akcyzy bez zapłaconego podatku akcyzowego w obrocie krajowym, jak również wewnątrzwspólnotowym pomiędzy państwami członkami Unii Europejskiej w ramach eksportu i importu. Uczestnikami tego systemu są podmioty, organizacje międzynarodowe, przedstawicielstwa dyplomatyczne dokonujące przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszania poboru akcyzy wewnątrz Unii Europejskiej oraz przedstawiciele organów podatkowych nadzorujących ww. przemieszczenia w obrocie zarówno krajowym, jak i wewnątrzwspólnotowym.

Według wnioskodawców czas od poprzedniej nowelizacji omawianej dzisiaj ustawy nie pozwolił wszystkim przedsiębiorcom, podmiotom na dostosowanie swoich wewnętrznych systemów informatycznych do zmian funkcjonalności, jakie przewiduje ustawa o podatku akcyzowym. Zaproponowana zmiana pozwala więc na utrzymanie papierowego dokumentu dostawy do okresu wskazanego w ustawie, co pozwoli przedsiębiorcom na dostosowanie się do uchwalonych wcześniej rozwiązań.

Dodatkowy rok vacatio legis dla tego rozwiązania według wnioskodawców umożliwi przedsiębiorcom zainstalowanie nowego oprogramowania, jego przetestowanie, współdziałanie z wewnętrznymi systemami informatycznymi przedsiębiorców z różnych dziedzin branży paliwowej, którzy posiadają różne systemy rozliczeń księgowych i magazynowych, a następnie płynne przejście z papierowego systemu na elektroniczny sposób monitorowania towarów objętych akcyzą. Ale tak jak zawsze, jak powiedziałem, nie dopilnowaliśmy sprawy i musimy przedłużać o kolejny rok wejście tej ustawy w życie. Wysoka Izbo! Mój klub popiera zaproponowane rozwiązania. Wnoszę o przekazanie tego projektu do dalszych prac w komisji. Bardzo dziękuję panu posłowi. Proszę o zabranie głosu pana posła Mieczysława Kasprzaka, klub parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Zabierając głos w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15, chcę powiedzieć, że jeżeli słuchamy tych wszystkich wypowiedzi, to wydawać by się mogło, że dzisiaj uchwalamy wielką rzecz, że tworzymy jakieś ciekawe rozwiązania, że to naprawdę ma uzdrowić naszą gospodarkę, jak zostało powiedziane wcześniej, a tak naprawdę my tylko zmieniamy datę wejścia w życie rozwiązań, które już dawno były uchwalone.

Tyle i aż tyle. Dlatego że - trudno - nie zdążono przez dłuższy czas wprowadzić rozwiązań zawartych w ustawie i w tej chwili na szybko trzeba tworzyć takie rozwiązanie. To jest strata czasu Wysokiej Izby, rządu i tych wszystkich, którzy muszą pracować w całym procesie legislacyjnym, bo te dwa drobne zapisy muszą przejść cały proces legislacyjny. Można było albo pospieszyć się i wprowadzić te rozwiązania wcześniej, przygotować oprzyrządowanie, albo zrobić to przy innej okazji. Przecież już od dłuższego czasu, jeszcze w tamtej kadencji można było dojść do wniosku, że nie zdążymy, więc o rok wydłużamy i nikt by nie miał pretensji. Lepiej szukać dobrych rozwiązań, żeby to zafunkcjonowało, niż tworzyć jakąś prowizorkę. Klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego - Kukiz15 poprze to rozwiązanie, bo ono jest logiczne. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Bardzo dziękuję panu posłowi za zabranie głosu. Proszę teraz o zabranie głosu w imieniu Koła Poselskiego Konfederacja pana posła Michała Urbaniaka. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Cóż, trzeba zacząć od tego, że ten projekt poprzemy. Zrobimy to głównie dlatego, że zależy nam na dobru przedsiębiorców, zależy nam na dobrostanie naszej gospodarki czy też na zmniejszeniu chaosu administracyjnego i jednocześnie na zmniejszeniu chaosu dotyczącego też samych procedur wdrażania większych systemów informatycznych w spółkach. Wiemy, że jest to proces długi, że jest to proces kosztowny dla większości przedsiębiorstw, stąd też rozumiemy propozycję przedłużenia okresu wdrożenia jeszcze o rok. Jednocześnie wyrażamy dość głębokie zaniepokojenie związane z faktem, że rząd nie potrafił przewidzieć skutków tego, co wdraża, że nie potrafili państwo przygotować projektu z założeniem większego horyzontu czasowego na wdrożenie konkretnych zmian. Zakładam, że wiedzą państwo, że jest to długi proces, ale jednak gdzieś coś nie zagrało. A więc, tak jak powiedziałem, tylko dlatego poprzemy ten projekt, że chcemy uniknąć chaosu. I nalegamy, zachęcamy do tego, żeby w przyszłości bardziej zwracać na to uwagę. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu posłowi. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja chciałem tylko wyjaśnić, że my popieramy tego typu vacatio legis, bo im więcej czasu mają ludzie do przygotowania się do zmian, tym lepiej.

Dzięki temu był ogromny rozwój gospodarczy, bo nikt tego nie kontrolował. Rozumiem niestety, że wraca PRL, wraca ta komuna z czasów przedwilczkowych. I niestety obawiam się, że ta jeszcze lepsza zmiana jest trudna do powstrzymania. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo panu posłowi za zabranie głosu. Przystępujemy do pytań. Informuję, że zapisało się do pytań siedmiu posłów. Zatem proszę o zabranie głosu pana posła Michała Szczerbę, Koalicja Obywatelska.

Panie Ministrze! Na podstawie art. 51 pkt 2 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, działając w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, wnoszę o przystąpienie do drugiego czytania niezwłocznie po zakończeniu pierwszego, bez odsyłania projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz Prawo celne, druk nr 51, do komisji. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość składam wniosek o nieodsyłanie poprawek do projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz Dziękuję bardzo panu posłowi za zabranie głosu. To jest pierwsze czytanie, panie pośle. W drugim czytaniu proszę to złożyć. Zresztą to będzie akurat zgodnie z intencją marszałka Sejmu, tak że proszę się nie denerwować. Teraz proszę o zabranie głosu panią poseł Martę Wcisło, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Wprowadzacie państwo zmiany w ustawie o podatku akcyzowym, które m.in. obligują do zmiany formy rejestrowania zakupów z formy papierowej na formę elektroniczną i dostosowania do systemu EMCS PL 2000. Moje pytanie brzmi. Co z mikroprzedsiębiorcami? Czy ich ta zmiana również będzie obligować? Nie ma możliwości, szanowni państwo, bezkosztowego wprowadzenia systemu komputerowego, dostosowania go do wymaganego systemu, bo niekiedy ten system nie funkcjonuje w małych, w mikroprzedsiębiorstwach. Myślę tutaj o małych punktach handlowych typu kioski, sklepy spożywcze, które przy okazji sprzedają wyroby akcyzowe i podlegają takim samym przepisom prawnym w myśl projektu ustawy, który państwo przygotowaliście, jak wielkie koncerny paliwowe.

Dziękuję bardzo, pani poseł. Proszę o zabranie głosu pana posła Tadeusza Tomaszewskiego, klub parlamentarny Lewica. Panie Marszałku! Szanowni przedstawiciele resortu! Można powiedzieć, że to ustawa typowo techniczna, niemniej jednak przekładamy jej wejście w życie już po raz kolejny. Czy państwo dzisiaj nie dostrzegacie pewnego zagrożenia w funkcjonowaniu obiegu papierowego, jeśli chodzi o dochody do budżetu państwa? Czy występuje jakieś niebezpieczeństwo, że brak elektronicznego rejestru może być powodem zmniejszenia dochodów do budżetu państwa?

Czy istnieje system publicznego wsparcia dla tych podmiotów, które są zobowiązane do wprowadzenia rejestru elektronicznego, pomocy publicznej przy wprowadzeniu tego systemu? Jako kolejny głos zabierze pan poseł Paweł Krutul, klub parlamentarny Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Proszę państwa, ta ustawa według mojej oceny w żadnym wypadku nie wpłynie na zmniejszenie spożywania alkoholu. A, okej, to przepraszam. Dziękuję bardzo panu posłowi. Ostatnim mówcą będzie pan poseł Romuald Ajchler, klub parlamentarny Lewica. Wysoka Izbo! Przed chwilą rozmawiałem z panem ministrem Suskim na temat tejże ustawy, a jak państwo wiecie, życie jest bogatsze niż nasza wyobraźnia. Ta ustawa nie dotyczy tylko mikroprzedsiębiorców itd., dotyczy także wszystkich tych, którzy kupują olej opałowy. Mianowicie jeśli emeryt, rencista ma domek jednorodzinny i potrzebuje do opalania tego domu czy ogrzewania tego budynku kupić 500 czy 1000 l oleju opałowego, musi mieć możliwość wprowadzenia systemu elektronicznego.

Lista osób zgłaszających się do pytania została wyczerpana. Proszę zatem o zabranie głosu pana Leszka Skibę, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.

Panie Marszałku! To bardzo ciekawa debata, bo rzeczywiście sprawa nie jest prosta, jeśli chodzi o wprowadzenie tylko i wyłącznie elektronicznego systemu wprowadzania danych do systemu EMCS. System e-DD właśnie zakłada ten mechanizm, że rezygnujemy z papieru i mamy tu wyłącznie system elektroniczny. Ale wbrew temu, o czym mówili tutaj posłowie, podstawowy problem, który jest, to jest właśnie problem implementacji - to też padało ze strony części posłów - czyli problem po stronie przedsiębiorców. Mamy do czynienia z systemem, który jest skomplikowany, który wymaga od firm ogromnych nakładów w zakresie zmian systemów informatycznych.

Uproszczeniem polegającym na tym, jeżeli ktoś nie chce wprowadzać. Nie wprowadzamy za pomocą dokumentacji papierowej, tylko elektronicznej. Ale w sytuacji, w której mamy do czynienia z ogromnymi firmami, takimi, które obracają ogromną ilością towarów objętych akcyzą, i jednocześnie tych zjawisk, zdarzeń codziennie jest bardzo dużo, to po prostu nie wystarczy zmuszenie człowieka, pracownika do klikania, wprowadzania danych. Potrzebujemy systemu automatycznego wprowadzania danych. To jest podstawowy problem, który pojawił się wiele, wiele miesięcy temu.

Tych zdarzeń, o których jest mowa, które dotyczą stosowania tej ustawy, jest tak wiele, że nawet na etapie jeszcze rok temu, gdy było wiadomo, że przesuwamy ten projekt o rok, nie było to zidentyfikowane, w związku z tym, że wdrażanie systemów informatycznych w wielkich organizacjach ma to do siebie, że po prostu w trakcie tego pojawiały się tam kłopoty. To jest właśnie podstawowy problem. Tu było pytanie, czy nie będzie jakichś nieprawidłowości, czy nie generujemy tutaj problemów.

Wiemy, że chcemy uprościć przedsiębiorcom życie, wprowadzając system elektroniczny, ale musi to być wprowadzane wtedy, kiedy oni będą na to gotowi, kiedy te projekty informatyczne się zakończą, kiedy te systemy będą przetestowane i nie będzie żadnych problemów z funkcjonowaniem, żadnych ryzyk prawnych związanych ze stosowaniem tej ustawy. Było też pytanie o mikroprzedsiębiorców.

Jeśli ktoś od czasu do czasu ma obowiązek wprowadzenia danych do systemu EMCS, to właśnie w ten sposób, za pomocą aplikacji Generator może to zrobić. Oczywiście to rozwiązuje problem mikrofirm w takim znaczeniu, że tych zdarzeń po prostu nie jest dużo i one mogą z tej aplikacji skorzystać.

Warto pamiętać, że mamy do czynienia. Tu też jest, mam wrażenie, jedno nieporozumienie. System EMCS dotyczy systemu, w którym.

W tym sensie jest to dobry przykład, bo pokazuje mechanizm zawieszonej akcyzy, czyli od tego alkoholu, który jest sprzedawany do apteki, nie ma pobieranej akcyzy.

W związku z tym mówimy o bardzo nielicznych przypadkach, w których mali i średni przedsiębiorcy korzystają z systemu EMCS.

Tu jest jedna ważna rzecz.

Możemy tutaj mówić tylko o ogrzewaniu gazowym.

Jest to uproszczona metoda, tak żeby nie było żadnych innych sposobów, które sprawiają, że jest to trudne. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu ministrowi za zabranie głosu. I teraz proszę o zabranie głosu przedstawiciela wnioskodawców pana posła Marka Suskiego. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wydaje mi się, że na większość pytań, może nawet na wszystkie pytania, wyczerpująco odpowiedział pan minister, natomiast tu pojawiła się też jedna kwestia, którą chciałbym sprostować. Powiedziano, że rząd nie zdążył i że to jest niechlujstwo, że teraz naprawiamy jakiś błąd, który jest po stronie rządu. Otóż, szanowni państwo, oczywiście można powiedzieć, że rząd mógł dać dużo więcej czasu na spełnienie tych wymogów, ale jak wiemy, natura ludzka jest taka, że jak taki czas wynosi 2 lata, to ludzie pewne rzeczy odkładają na przyszłość i później, na koniec też nie są w stanie zdążyć.

Nie jest to jakieś zaniedbanie rządu, więc bardzo prosiłbym o niewprowadzanie opinii publicznej w błąd. To tyle, szanowni państwo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi. W trybie krótkiego sprostowania pan poseł Romuald Ajchler. Panie Ministrze!

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi. Zamykam dyskusję. W dyskusji zgłoszono wniosek o przystąpienie niezwłocznie do drugiego czytania projektu ustawy. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy zatem do drugiego czytania projektu ustawy. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos w drugim czytaniu tego projektu ustawy? W takim razie proszę o zabranie głosu pana posła Jerzego Maternę. Wysoka Izbo! Klub Prawa i Sprawiedliwości w drugim czytaniu chce zgłosić poprawkę do projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz

Prawo celne i przystąpienie do drugiego czytania po doręczeniu posłom poprawek. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu posłowi.

Czas na wystąpienie ustalam na 3 minuty. To jest właśnie sposób procedowania nad ustawami przez Prawo i Sprawiedliwość.

Tak naprawdę nie wiemy. Może któryś z tych posłów chciałby złożyć poprawkę, może nie.

W związku z tym, panie marszałku, proszę o uwzględnienie faktu, że siedząc tam, zgłosiłam sprzeciw. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani poseł. W tym samym trybie, w imieniu klubu parlamentarnego Lewica, pan poseł Romuald Ajchler.

Macie 11 miesięcy. Lewica powiedziała, że poprze ten projekt ustawy, ale wykorzystajcie w ramach tego.

Papierowe zamówienia, jak do tej pory to funkcjonowało, i papierowy odbiór. A elektronicznie będzie musiał potwierdzić wpływ oleju opałowego emeryt. Zastanówmy się, Wysoka Izbo, co chcemy zgotować tym ludziom? Chodzi o to, żeby przekonać resort finansów.

Dlatego apeluję do pana o to, aby właśnie z tej sytuacji skorzystać. Dziękuję bardzo panu posłowi. Stwierdzam, że lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana.

Panie Marszałku! Ważne, żeby zrozumieć nieporozumienie, czyli to, na jakiej podstawie pan poseł Ajchler twierdzi, że system EMCS - tzn. mechanizm zgłaszania elektronicznego czy nieelektronicznego - nakłada na emerytów kupujących olej opałowy jakiekolwiek obowiązki. Tzn. ja rozumiem, że rzecz dotyczy tego, żeby mieć świadomość, że są dwa oddzielne systemy, które obejmują towary akcyzowe. Jest system europejski EMCS, który dotyczy wszystkich transakcji międzynarodowych i też tych z zawieszoną akcyzą, i też w obrębie Polski, czyli wtedy, kiedy akcyza nie jest płacona.

Lepiej elektronicznie. Jest drugi system, o którym mówił pan poseł - system SENT, który został stworzony 2 lata temu.

W drugiej połowie roku 2016, kiedy ten system się pojawił, pozwalał na to, żeby zgłaszać wszystkie ruchy ciężarówek, które przewoziły paliwo.

I tam rzeczywiście jest tak, że te metody, które dotyczą potwierdzania tego, że ten towar został przyjęty, nadawania, odbierania itd., mają swoją strukturę. Oczywiście pan poseł może powiedzieć: Czemu nie dostosujecie systemu SENT do systemu EMCS? Od razu odpowiadam: tak, prace nad tym, żeby dostosować te dwa systemy, żeby to uprościć, żeby były podobne sposoby, są prowadzone w Ministerstwie Finansów.

W takim znaczeniu, że te zmiany muszą dawać gwarancję, że nie wytwarzamy dziury, bo zaraz pojawią się i skorzystają z tego przestępcy. W związku z tym mogę powiedzieć i zapewnić pana posła, że na pewno robimy wszystko, żeby te dwa systemy ze sobą zintegrować w jak największej skali.

Właściwie tu nie chodzi o to, żeby posiadać komputer.

Tego oleju jest tak dużo, że właściwie to jest - że tak powiem - mało prawdopodobne, a tak naprawdę był on przeznaczany dla firm, które prowadziły transport drogowy, wlewały do swoich ciężarówek.

Zamykam dyskusję. Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm przystąpił do trzeciego czytania projektu ustawy po doręczeniu paniom i panom posłom zestawienia poprawek. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 4. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk nr 40) Proszę pana ministra Leszka Skibę o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy.

Pragnę przedstawić rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, zawarty w druku nr 40. Ustawą z dnia 6 lipca 2016 r. wprowadzono do polskiego systemu prawnego nową daninę - podatek od sprzedaży detalicznej. Jej uchwalenie było poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi, spotkało się z akceptacją wielu handlowców. Celem wprowadzenia nowego podatku, oprócz zwiększenia dochodów podatkowych budżetu państwa, było wyrównanie uszczerbku budżetowego wynikającego ze stosowania przez dużych detalistów praktyk optymalizacyjnych w podatku dochodowym od osób prawnych. Komisja Europejska wszczęła szczegółową procedurę dochodzenia w sprawie naszego podatku. Komisja twierdziła, że progresywne stawki oparte na wielkości przychodu przyznają przedsiębiorcom o niskich przychodach selektywną korzyść, dającą im tym samym przewagę nad większymi konkurentami, co narusza unijne zasady pomocy publicznej. Jednocześnie Komisja Europejska wydała nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia badania jego legalności przez Komisję. Aby uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi stosowania ustawy w przypadku niekorzystnego dla Polski rozwiązania sporu z Komisją Europejską, Sejm uchwalił 15 listopada 2016 r. ustawę zawieszającą stosowanie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej do końca 2017 r. Przewidywaliśmy, że kwestia możliwości pobierania podatku na zasadach określonych w ustawie w terminie tym zostanie rozstrzygnięta. Byliśmy wówczas w trakcie formalnej skargi do sądu Unii Europejskiej na decyzję wstępną Komisji w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej, która ostatecznie została złożona przez Polskę 30 listopada 2016 r.

Komisja stwierdziła, że dzięki progresywnym stawkom opartym na wielkości przychodu przedsiębiorstwa o niskich obrotach mają przewagę konkurencyjną. W ocenie Komisji Polska nie wykazała, że progresywne stawki podatku są uzasadnione w przypadku podatku od sprzedaży detalicznej w zakresie opodatkowania całego sektora handlu detalicznego ani że przedsiębiorstwa objęte wyższą stawką mają większą zdolność do zapłaty podatku. Polska nie zgadza się z dokonaną przez Komisję oceną polskiego podatku od sprzedaży detalicznej w kontekście zasad państwa prawa. Dlatego w dniu 13 września 2017 r. złożona została skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej również na decyzję Komisji Europejskiej z dnia 30 czerwca 2017 r. Wobec kontynuowania sporu z Komisją w postępowaniu sądowym w dniu 12 października 2017 r. uchwalono przedłużenie zawieszenia poboru podatku do końca 2018 r. Obie skargi wniesione przez Polskę zostały połączone do wspólnego rozpatrywania na rozprawie oraz wydania wyroku. Do końca tego roku nie zapadł wyrok w sprawie, jak również nie wyznaczono daty jego ogłoszenia. Wobec powyższego zawieszenie stosowania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej zostało przedłużone do końca 2019 r. Postępowanie przed sądem Unii Europejskiej zostało zakończone wyrokiem z dnia 16 maja 2019 r. Sąd całkowicie podzielił stanowisko Polski i orzekł, że podatek od sprzedaży detalicznej nie stanowi pomocy państwa. Sąd stwierdził nieważność zarówno wstępnej, jak i ostatecznej decyzji Komisji w zakresie podatku od sprzedaży detalicznej.

Brak prawomocności wyroku powoduje, że otoczenie prawne, w jakim funkcjonowałby polski podatek, nadal nie byłoby pewne. W tej sytuacji racjonalnym rozwiązaniem jest zawieszenie stosowania ustawy i poboru podatku na kolejne pół roku, podczas którego najprawdopodobniej zapadnie wyrok TSUE co do zgodności podatku z przepisami o pomocy państwa. Bez wyroku sądu II instancji pobieranie podatku na zasadach określonych w ustawie mogłoby narazić Skarb Państwa na straty ze względu na konieczność zwrotu pobranego podatku w przypadku niekorzystnego dla Polski rozwiązania.

Oczekujemy, że do tego czasu zostanie wydany korzystny dla Polski wyrok, który umożliwi pobieranie zawieszonego podatku. Wysoka Izbo! Przekazując Wysokiej Izbie projekt ustawy do rozpatrzenia, mam nadzieję, że będzie on przyjęty ze zrozumieniem, a prace nad nim przebiegną sprawnie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu ministrowi. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Przystępujemy do tej części naszego punktu. Proszę o zabranie głosu w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość pana posła Henryka Kowalczyka. Wysoka Izbo!

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość popiera przesunięcie tego terminu o pół roku.

Szanowny Panie Marszałku!

Dziękuję bardzo panu posłowi za zabranie głosu. Proszę o zabranie głosu w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska panią posłankę

Mam przyjemność przekazać stanowisko klubu Koalicji Obywatelskiej wobec projektu zmiany ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, druk nr 40. Ustawa, jak tutaj już tłumaczył pan minister, ma zawiesić, czyli opóźnić wejście w życie podatku handlowego o kolejne 6 miesięcy, czyli do lipca 2020 r. Jest to trzecie zawieszenie poboru tego podatku w związku z postępowaniem trwającym przed sądem Unii Europejskiej pomiędzy Komisją Europejską a rządem polskim, gdyż Komisja pierwotnie uznała, że progresja zastosowana w tym podatku może stanowić niedozwoloną pomoc publiczną dla części punktów handlowych znajdujących się w Polsce. Będziemy proponować, by dalej procedować tę ustawę. Jednak wydaje mi się, że lepiej, żebyśmy jednak w komisji o tym podyskutowali. Natomiast to nie znaczy, że zmieniamy zdanie w sprawie podatku handlowego od sprzedaży detalicznej, który w naszej ocenie zostanie w 100% zapłacony przez obywateli, bo jak każdy podatek sektorowy zostanie on po prostu przerzucony na konsumentów. Wcześniej już mieliśmy podobne podatki sektorowe wprowadzone do polskiego systemu podatkowego, jak np. podatek od instytucji finansowych. Doświadczenia pokazują, że w 100% zapłacili go obywatele w postaci wzrostu cen usług, z których w tych instytucjach finansowych korzystają.

Ale tak naprawdę tę drożyznę w sposób istotny zaczynamy odczuwać od około roku. I niestety czekają nas kolejne podwyżki, wzrost cen życia. Dlatego wejście w życie w połowie roku tego podatku i przełożenie go na ceny żywności nie jest rzeczą pożądaną. Sprawi, że życie obywateli będzie droższe, dlatego w naszej ocenie ten podatek powinien zostać oddalony bardziej. Dlaczego uważamy, że będą kolejne podwyżki kosztów życia? Wiemy dobrze, że za chwilę czeka nas bardzo istotna podwyżka cen prądu. Te podwyżki przełożą się na koszty produkcji, a co za tym idzie - koszty towarów, usług, z których na co dzień korzystamy i które kupujemy. Czeka nas podwyżka cen paliwa, niby niewielka, bo szacuje się, że 138 zł od 1 tys. l, ale znowu w systemie produkcji w gospodarce przełoży się to na wzrost kosztów produkcji i wytwarzania towarów i ich transportu z miejsca produkcji do miejsca sprzedaży. Powód to wzrost płacy minimalnej i zabezpieczenie środków na wyższe płace w tychże spółdzielniach. Tak można by naprawdę bardzo dużo wymieniać. Czeka nas podwyżka cen za wywóz nieczystości, która z kolei wyląduje w naszych kieszeniach, ponieważ zaostrzone zostały warunki segregacji odpadów i ich utylizacji.

Składam sprzeciw wobec przejścia od ręki do drugiego czytania. Uważam, że ta ustawa powinna trafić do Komisji Finansów Publicznych, by tam jeszcze raz można było przedyskutować, w jaki sposób ten podatek przełoży się na codzienne życie obywateli i obywatelek. Dziękuję bardzo, pani poseł. Proszę teraz o zabranie głosu w imieniu klubu parlamentarnego Lewica panią posłankę Anitę Sowińską. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić stanowisko Lewicy w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Zdradzę państwu pewną tajemnicę. Wiecie, czym zajmują się przedsiębiorcy? Zarządzaniem, planowaniem, organizowaniem, kontrolowaniem. A wiecie państwo, czym zajmuje się rząd albo czym powinien zajmować się rząd? Dokładnie tym samym. Zarządzaniem, tyle że w większej skali, w skali całego państwa. Różnica polega na tym, że przedsiębiorca każdego dnia ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje, odpowiedzialność imienną i odpowiedzialność finansową. Jeżeli przedsiębiorca nieumiejętnie zarządza swoją firmą, to ta ponosi straty i w najgorszym wypadku firma upada, ale to jest ta jedna firma. Jeżeli natomiast rząd nieumiejętnie zarządza państwem, ma to przełożenie na firmy w całym kraju. Paradoks polega na tym, za złe, nieprzemyślane albo po prostu opieszałe decyzje rządzący nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Dlatego w przypadku rządu i całego parlamentu tak ważna jest odpowiedzialność. To wasze decyzje, albo ich brak, decydują o tym, czy firmy są czy ich nie ma. W konsekwencji ma to przełożenie na wszystkich obywateli. W przypadku ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej ewidentnie zabrakło odpowiedzialnego zarządzania, zabrakło wam wyobraźni i zabrakło działania. Być może dlatego, że nie ponosicie odpowiedzialności za swoje czyny - ani finansowej, ani nawet imiennej. 24 lipca tego roku Komisja Europejska odwołała się od wyroku Sądu Europejskiego do sądu drugiej instancji. Od tego momentu wiedzieliście, pan, panie premierze, wiedział, że Polska musi poczekać z wprowadzeniem nowego podatku na prawomocny wyrok sądu. Wiedzieliście, że zegar tyka - tik tok, tik tok - ale nie zrobiliście nic. Pytam zatem: Dlaczego tej prostej ustawy przedłużającej zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej rząd premiera Morawieckiego nie przedstawił już we wrześniu? Przecież już wtedy było wiadomo, że procedowanie tej sprawy w sądzie potrwa dłużej. Jak przedsiębiorcy mają prowadzić swoje biznesy w tym bałaganie?

Wtedy, kiedy chcecie, drukujecie wyroki, kiedy nie chcecie, nie drukujecie. Wszystko się wam należy, ale - i być może będzie to zdziwienie dla was - wszystkich innych obowiązuje prawo, zarówno to dobre, jak i to złe, uchwalane w chaosie i na ostatnią chwilę, pisane na kolanie i przegłosowywane w nocy, po ciemku. Zwykli obywatele, przedsiębiorcy nie mogą w przeciwieństwie do was liczyć na wyjątki. Mamy 12 grudnia i rząd składa w końcu ustawę. Właściwie jest to już po czasie, ponieważ jeżeli Senat wykorzysta cały dostępny czas na proces legislacyjny, ryzykujemy, że ten podatek wejdzie w życie już teraz, przed prawomocnym wyrokiem sądu, a to jest w państwie prawa niedopuszczalne. Dlatego Lewica poprze ten projekt.

A rządowi chciałabym przypomnieć, że rządzenie krajem to jest służba, służba ludziom, a nie odwrotnie. Zarządzajcie tym domem z głową. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani poseł. Proszę teraz o zabranie głosu pana posła Krzysztofa Paszyka w imieniu klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego - Kukiz15. Bardzo dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

To nie oznacza, że nie mamy swoich spostrzeżeń i krytycznych uwag co do meritum zawartego w ustawie dotyczącej obrotu detalicznego, wątpliwości przede wszystkim kierowanych w stronę tych, którym dzisiaj najtrudniej związać koniec z końcem, a co do których praktyka życia ostatnich kilkudziesięciu lat pokazuje, że niestety dotkną ich konsekwencje wejścia w życie tego podatku, niemniej dzisiaj trzeba kierować się przede wszystkim troską o pewność obrotu gospodarczego i prawnego.

Teraz proszę o zabranie głosu w imieniu Koła Poselskiego Konfederacja pana posła Dobromira Sośnierza. Miło mi wziąć udział w takiej zażartej debacie przy licznej obecności państwa posłów. Właściwie najchętniej głosowalibyśmy przeciwko tej ustawie, ponieważ głosowanie nad projektami na wczoraj na pewno nie zasługuje na uznanie. Jest to absolutnie niedopuszczalne, żeby 12 grudnia rozpoczynać proces legislacyjny dotyczący wejścia w życie podatku, który ma wejść w życie 1 stycznia, bo to oznacza, że w Polsce przedsiębiorcy do końca grudnia nie będą pewni, jakie podatki będą płacić w nowym roku. Jest to sytuacja zupełnie absurdalna, nie ma ku temu żadnych rozsądnych powodów, bo fakty w tej sprawie były znane już od dłuższego czasu.

Najchętniej głosowalibyśmy przeciwko, natomiast de facto głosowanie przeciwko tej ustawie oznaczałoby głosowanie za wprowadzeniem nowego podatku.

W tej sprawie Komisja Europejska ciąga nas od kilku lat po sądach. Nasze państwo nie może wprowadzić podatku. Paradoksalnie w tym przypadku Komisja Europejska działa w interesie polskiego podatnika, aczkolwiek z uzasadnieniem absolutnie bzdurnym. Nie wiadomo komu przyznać rację i komu kibicować, ponieważ z jednej strony Komisja oczywiście nie ma racji, że jest to pomoc publiczna, a z drugiej strony dzięki temu, że nie ma racji, opóźnia o kilka lat wejście w życie szkodliwego dla podatników podatku.

Dziękuję bardzo panu posłowi, który zabrał głos w imieniu Koła Poselskiego Konfederacja. Jeżeli nie ma więcej osób, zamykam listę mówców. Proszę o zabranie głosu panią poseł Magdalenę Łośko reprezentującą Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dlaczego rząd w sytuacji, kiedy nie jest znane rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, proponuje w projekcie ustawy, aby przepisy miały zastosowanie do przychodów ze sprzedaży po 1 lipca 2020 r. Czy jeśli wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do tego czasu nie zapadnie, mamy spodziewać się kolejnych przesunięć? Na jakiej podstawie wyznaczono taki, a nie inny termin? Każde przedsiębiorstwo pracuje według pewnego planu uwzględniającego politykę cenową i finansową. Proponowany przez ministerstwo zapis wprowadza chaos.

Tego typu regulacje powinny być wprowadzane z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, tak aby przedsiębiorstwa mogły uwzględnić w swoich planach finansowych konieczność zapłaty nowego podatku i się do tego w odpowiedni sposób przygotować. Czy rząd stworzy przedsiębiorstwom możliwość dostosowania się do zmian, które mogą nastąpić po ewentualnie korzystnym dla rządu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Proszę o zabranie głosu panią poseł Zofię Czernow, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Oczywiście biorę pod uwagę te wszystkie zastrzeżenia, o których była mowa. Nie będę ich powtarzać. Ten projekt ma szczegółowe uzasadnienie. Kiedy czytamy to uzasadnienie, powstają bardzo poważne wątpliwości.

Chodzi mi o skutki dla budżetu.

Po co wprowadzamy ten podatek? Żeby były ujemne skutki dla budżetu? Dziękuję bardzo, pani poseł.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

On jest bardzo enigmatycznie nazwany: podatek od sprzedaży detalicznej. Mało kto zdaje sobie sprawę, że będzie to miało wpływ na wysokość cen produktów w sklepach. Według danych ministerstwa ma tym zostać objętych ok. 200 przedsiębiorstw, pewnie również średnich, co oznacza, że nie tylko markety, ale także polskie firmy, które próbują na tym trudnym rynku prowadzić działalność, zostaną uderzone właśnie tym podatkiem. I oczywiście nietrudno sobie wyobrazić, że te polskie firmy, dla których będzie to silny impuls kosztowy, będą chciały przerzucić te koszty na klientów, co oczywiście spowoduje wzrost cen towarów w sklepach. Panie Ministrze!

To byłoby działanie rozsądne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Głos zabierze pan poseł Krzysztof Paszyk w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska. Wysoka Izbo! Korzystając z okazji, chciałbym się zwrócić, panie ministrze, z pytaniem do pana: Czy jest jakaś refleksja w resorcie, żeby tak zmodyfikować tę ustawę, aby w momencie wejścia w życie, po pierwsze, chroniła najuboższych konsumentów na rynku przed takim wprost przerzuceniem tego podatku na konsumenta, a po drugie, żeby w należyty sposób, a nie tylko teoretycznie, zabezpieczała interes budżetu państwa? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi. Proszę o zabranie głosu pana posła Tadeusza Tomaszewskiego, klub parlamentarny Lewica. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie!

Czy ta ustawa w znacznej mierze będzie obciążać również naszych polskich przedsiębiorców, tych rodzinnych? Oczywiście ustawa przewiduje, że kwota wolna jest oznaczona właśnie w ustawie, a czy to jest jednak tylko i wyłącznie podatek od wielkich marketów (Dzwonek) czy jednak będzie dotykał również naszych przedsiębiorców? Dziękuję. Dziękuję bardzo panu posłowi. Proszę o zabranie głosu pana posła Henryka Kowalczyka, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Chciałbym prosić o potwierdzenie tezy, że wzrost cen towarów i usług oraz kosztów utrzymania był właśnie za rządów PO-PSL.

A więc jakby to sumarycznie złożyć, to w tamtym okresie było ponad 20% wzrostu i wtedy to nie przeszkadzało. Natomiast teraz straszenie bardzo małą inflacją jest absolutnie nie na miejscu.

Dziękuję bardzo panu posłowi. Proszę teraz o zabranie głosu podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów pana ministra Leszka Skibę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rzeczywiście to jest tak, że mamy do czynienia dziś z dyskusją nad opóźnieniem wejścia w życie tego projektu.

Pytania pojawiają się o to. Warto popatrzeć na kontekst czasu.

Jest to na pewno korzystne z punktu widzenia przedsiębiorców, aby mieć jeszcze czas, ale nikt tutaj nie zaprzeczy, że ten podatek po prostu wejdzie w życie.

I rzeczywiście pełna zgoda, że tych przedsiębiorców nie jest aż tak dużo.

Rozwiązania związane z wprowadzeniem tej ustawy, gdy ustawa wejdzie w życie, gdy podatek od sprzedaży detalicznej wejdzie w życie, zabezpieczą interesy budżetu w taki sposób, że po prostu pieniądze będą tam trafiać.

A teraz mamy do czynienia właśnie z dbałością o przewidywalność, o współpracę z przedsiębiorcami. Nie stracą na tym najbiedniejsi.

Ta powiększona marża będzie zredukowana, z tej powiększonej marży właśnie przedsiębiorcy będą płacić ten podatek. Z jednej strony mamy głosy wielu małych i średnich przedsiębiorców, którzy twierdzą, że jest nierówność, jeśli chodzi o konkurencję na rynku handlu, czyli mali i średni zachęcają rząd do tego, aby walczyć o ten podatek i wprowadzić go w życie. Jest to zatem oczywiste, że podatek jest korzystny z punktu widzenia polskich przedsiębiorców, szczególnie tych małych i średnich. Oczywiście należy na bieżąco monitorować wpływ tego podatku, gdy zacznie on działać, będzie wpływ na ceny, na pewno będzie to niezmiernie ważne, żeby wiedzieć, w jaki sposób ten podatek funkcjonuje i jaki ma wpływ na relacje handlowe, wpływ właśnie na to, jak działają te firmy. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Wobec zgłoszonego wniosku o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania projektu ustawy zgłoszono sprzeciw. Do głosowania w tej sprawie przystąpimy w bloku głosowań. Wysoka Izbo! Komisja Finansów Publicznych przedłożyła sprawozdanie o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, druk nr 60. W związku z tym, na podstawie art. 74 regulaminu Sejmu, marszałek Sejmu podjęła decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Marszałek Sejmu proponuje, aby w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego Sejm wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 42 i 55) Proszę pana posła Zbigniewa Babalskiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Na posiedzeniu komisji została rozpatrzona sprawa dotycząca zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W czasie dyskusji zgłoszono 5 poprawek. 4 zostały odrzucone, 1 została przyjęta. Mam zaszczyt i obowiązek w imieniu komisji zwrócić się do Sejmu o przyjęcie powyższej uchwały Sejmu dotyczącej zmiany regulaminu Sejmu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu posłowi. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Otwieram dyskusję. Proszę pana posła Krzysztofa Sobolewskiego z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość o zabranie głosu. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawić stanowisko wobec uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Poselski projekt zmiany regulaminu Sejmu, zawarty w druku nr 42, dotyczy zmiany związanej ze zmienionym Kodeksem wyborczym, którego to zmiany dokonano 11 stycznia 2018 r. w zakresie kreowania składu Państwowej Komisji Wyborczej. Zmiana ta miała na celu zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, w tym Państwowej Komisji Wyborczej. Zmiany dokonane w Kodeksie wyborczym w styczniu 2018 r. spowodowały albo przyczyniły się do tego, że wybory parlamentarne i samorządowe oraz wybory do Parlamentu Europejskiego przebiegły sprawnie, a już szczególnie wybory parlamentarne, głosowanie przebiegło sprawnie, a wyniki zostały ogłoszone pierwszy raz w historii w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania. A więc wszystkie podnoszone wtedy przy zmianach Kodeksu wyborczego zarzuty, że zmiany te doprowadzą do tego, że wybory albo nie zostaną przeprowadzone, albo zakończą się totalną klapą, okazały się, jak widać, po raz kolejny tylko rzucanymi bezpodstawnie oskarżeniami ze strony opozycji.

Oczywiście jest przewidziane, że będzie to wybór proporcjonalny do wielkości klubów i że będzie przez Prezydium Sejmu ustanowiony po przyjęciu tych zmian, po przyjęciu tej uchwały termin na zgłaszanie kandydatów.

Kończąc, panie marszałku, mam zaszczyt poinformować, że Prawo i Sprawiedliwość będzie w pełni popierało te zmiany w uchwale. Dziękuję bardzo panu posłowi. W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska głos zabierze pan poseł Jarosław Urbaniak. Polska, ale to polska Koalicja Obywatelska. Przecież to w pracy. Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie!

Te zmiany uderzają w podstawy demokracji, w podstawy państwa prawnego. Pewnie z tego powodu tak długo, do momentu, aż nastąpiły pilne terminy, PiS czekał z implementacją tych zmian w Kodeksie wyborczym do regulaminu Sejmu. I te zmiany w regulaminie Sejmu są mniej ważne, bo grzech pierworodny, a nawet powiedziałbym: grzechy pierworodne były zrobione właśnie wtedy, w styczniu 2018 r. Dwa grzechy w tej chwili implementujemy do regulaminu Sejmu. Chodzi o zerwanie z modelem sądowym Państwowej Komisji Wyborczej oraz wprowadzenie możliwości odwoływania członków Państwowej Komisji Wyborczej. Do tej pory obowiązywał system sądowy, tzn. że członków PKW wskazywał Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny.

To, co nam w tej chwili się proponuje, to że na dziewięciu członków Państwowej Komisji Wyborczej aż siedmiu będzie powołanych z wyboru Sejmu. To naruszenie nie tylko konstytucji, a w szczególności art. 2 mówiącego o tym, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym.

Wy nie łamiecie prawa. Ale, panie pośle, nie ma się z czego śmiać. Później trafiają się Banasie. Powiedziałem, że łamanie konstytucji to jedno, ale to, że siedmiu członków PKW na dziewięciu będzie wybieranych przez Sejm, to jest złamanie jednej z podstawowych zasad naszej cywilizacji, europejskiej, cywilizacji łacińskiej, że nie wolno być sędzią we własnej sprawie. Panie Marszałku! W imieniu klubu mam do przedłożenia trzy poprawki, które ratują, mam nadzieję, ten bardzo fatalny projekt regulaminu Sejmu, dotyczące m.in. tego, kto ma prawo złożyć wniosek o odwołanie członka Państwowej Komisji Wyborczej.

Proszę teraz o zabranie głosu panią posłankę Katarzynę Kotulę reprezentującą klub parlamentarny Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić stanowisko klubu parlamentarnego Lewicy w sprawie projektu z druku nr 42, tj. poselskiego projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej. Projekt uchwały dotyczy uregulowania spraw związanych ze wskazaniem przez Sejm członków Państwowej Komisji Wyborczej.

Mamy świadomość, że odwoływanie osób powoływanych na różne stanowiska faktycznie średnio się ekipie rządzącej ostatnio udaje. Odwoływanie członków PKW może zostać zgłoszone przez Prezydium Sejmu albo grupę 35 posłów. W projekcie uchwały zawierającej wniosek projektodawca zobowiązany będzie wskazać powody wystąpienia z wnioskiem, jednak przepis w tej formie, w jakiej jest tu obecny, daje oczywiście możliwość nadużycia. W przypadku członków Państwowej Komisji Wyborczej, w celu zachowania niezależności członków PKW, procedura odwołania powinna być prawnie ograniczona. Dodatkowo należy wskazać także na nieostrość terminu: uzasadniony wniosek. Rekomendowaliśmy rozważenie zawarcia konkretnych przesłanek, które mieściłyby się w terminie: uzasadniony wniosek w celu odwołania członka PKW, ale zostały one odrzucone. Mamy także świadomość, że nowelizacja Kodeksu wyborczego z 2018 r. zwiększa polityczną kontrolę nad PKW, ponieważ po zmianach tylko jeden członek PKW wskazany przez prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego nie będzie pochodził z wyboru politycznego. Chcielibyśmy móc liczyć na niezależność wybranych członków PKW, tak aby wykonywali oni swoje obowiązki bez politycznych nacisków. W połączeniu z możliwym politycznym odwołaniem członków PKW istnieje zagrożenie politycznego wpływu PKW w większym zakresie, niż przewiduje ustawa. Rozumiemy, że stosuje się to tylko w sytuacjach wyjątkowych, niecierpiących zwłoki. Trudno uzasadniać, że mamy do czynienia z taką sytuacją w przypadku tej uchwały. W związku z tym klub parlamentarny Lewicy wnioskuje o odrzucenie uchwały w obecnym kształcie. Dziękuję bardzo pani posłance. Teraz w imieniu klubu parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 głos zabierze pani poseł Jolanta Fedak.

Wysoka Izbo! Dawno, dawno temu, 11 stycznia 2018 r., zmieniono w taki sposób Kodeks wyborczy, że kreacją składu Państwowej Komisji Wyborczej ma się zająć w dużej mierze Sejm. Ma on mianowicie wybrać siedem osób spośród sędziów, którzy mają właśnie te kwalifikacje sędziowskie, aby weszli oni w skład tej komisji wyborczej. Mówię o tym z pewnym sarkazmem, dlatego że mieliśmy dosyć czasu na to, aby zastanowić się, w jaki sposób ewentualnie tę kreację - skoro ona już jest w Kodeksie wyborczym czy już w ustawie - zmienić, żeby była dość sensowna. On jest bardzo nieodległy, bo to jest raptem jakiś miesiąc na to, żeby Sejm zebrał te kandydatury, wybrał i przedstawił panu prezydentowi, czyli niedługi czas. Pierwsza zapytałam o to, jaki jest katalog - skoro już kontynuujemy, że tak powiem, wybór czy uzupełniamy regulamin Sejmu po zmianie ustawy - odwołań takiego członka komisji wyborczej?

Tym bardziej że sytuacja już na początku jest dwuznaczna. Mianowicie Sejm, czyli posłowie, którzy są wybierani w wyborach, kreują tę władzę i mają absolutnie możliwość bez żadnego istotnego powodu odwołania tego członka, czyli takiego bardzo silnego nacisku. Wydaje mi się, że ta sytuacja jest tak dalece dwuznaczna, że jeszcze raz proszę, abyście się państwo nad tym zastanowili.

Ostatnie wybory wskazywały na to, że nic takiego strasznego się nie zdarzyło, że Państwowa Komisja Wyborcza szybko podawała wyniki, że to funkcjonowało dobrze.

Wiem, że państwo możecie mieć uraz po ostatnich rzeczach, które zdarzyły się z szefem NIK-u, ale cóż, nie leczymy tu urazów, tylko uchwalamy dobre prawo. Mam nadzieję. My nie przyłożymy do tego ręki. Jako klub wstrzymamy się od głosu, uznając, że jest to po prostu.

Bardzo dziękuję, pani poseł. W imieniu Koła Poselskiego Konfederacja głos zabierze pan poseł Krystian Kamiński.

W związku z nowelizacją Kodeksu wyborczego w 2018 r. zmiana regulaminu Sejmu jest koniecznością. Zamysł nowelizacji miał polegać na zwiększeniu udziału obywateli w procesie wyborów funkcjonowania i kontroli organów publicznych, a w rzeczywistości ma zupełnie inny skutek. Wybór przez Sejm siedmiu z dziewięciu członków PKW nie jest zwiększeniem wpływu wyborców na instytucję publiczną, ale jest ograniczeniem niezależności, niezawisłości, neutralności, apolityczności i bezstronności. Stan, w którym osoby wybrane przez polityków z PiS-u, Platformy, SLD i PSL-u będą stanowiły większość tych osób, na pewno nie zwiększy prestiżu tej instytucji. Dodatkowo jest to kolejny projekt PiS-u, który ignoruje 1250 tys. wyborców Konfederacji, który powoduje, że przedstawiciele Konfederacji pomimo demokratycznego mandatu są przez PiS sekowani. Powyższy regulamin stoi w sprzeczności z demokratycznymi wyborami i każdy, kto za nim zagłosuje, zagłosuje za odebraniem głosu dużej części społeczeństwa. W związku z powyższym koło Konfederacji zagłosuje przeciwko zmianom w regulaminie Sejmu. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby? Pan poseł Urbaniak. Pan poseł Mirosław Suchoń. Czas na zadawanie pytania ustalam na 1 minutę. Proszę o zabranie głosu pana posła Michała Szczerbę, Koalicja Obywatelska. Nie ma. Zatem proszę pana posła Dariusza Klimczaka, Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 - Koalicja Polska. Wysoka Izbo! Przedmiotowa zmiana kodeksu dowodzi tylko tego, że pomysłodawcy z Prawa i Sprawiedliwości chodzi jedynie o zmiany personalne. Zresztą jak we wszystkich reformach Prawa i Sprawiedliwości chodzi jedynie o zmiany personalne, a nie o żadne usprawnienie systemu, jakikolwiek miałby być. Natomiast w uzasadnieniu, które przedstawił pan poseł, sam sobie zaprzeczył. Jeżeli tak dobrze zostały przeprowadzone te wybory, to po co państwo chcą zmieniać sędziów w PKW, chyba że państwo deklarują, że powołają tych samych. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu posłowi Dariuszowi Klimczakowi. Głos zabierze pan poseł Krzysztof Paszyk, klub parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 - Koalicja Polska. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mianowicie, co to będą za kryteria, które będą powodowały, że Wysoka Izba będzie dokonywała zmian w składzie. Czy to, nie wiem, brak zaufania klubu? Jakieś przewinienia? Czy też, nie wiem, utrata zaufania państwa prezesa będzie np. tym czynnikiem, który będzie powodował, że właściwie swobodnie państwo jako większość sejmowa będziecie mogli dokonywać zmian w organie, który powinien cechować się ekstremalnie dużą niezależnością. Ważne, panie pośle, żeby Wysoka Izba (Dzwonek) te wątpliwości miała rozwiane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi. Proszę o zabranie głosu pana posła Jarosława Urbaniaka, Koalicja Obywatelska. Chciałem zapytać wnioskodawców o te skandaliczne przepisy dotyczące odwołania członka PKW, o dwie rzeczy. 35 posłów może wystąpić z wnioskiem o odwołanie. Pani poseł wczoraj w komisji mówiła: Ale przecież 15 może wystąpić z inicjatywą ustawodawczą. Tak, bo my jesteśmy od ustanawiania prawa. To jest ta różnica. A tu się wtrącamy w PKW. Druga rzecz. Mam pytanie: Czy historia z panem prezesem Banasiem i z jego licznymi kłopotami miała wpływ na to, że wprowadzacie przepisy, na podstawie których tak naprawdę można bez podania poważnego powodu wystąpić z wnioskiem o odwołanie członka PKW? Przecież taki przepis jest jak miecz Damoklesa wiszący nad każdym członkiem PKW.

Proszę o zabranie głosu pana posła Mirosława Suchonia, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ta zmiana jest oczywista. Chodzi o zagwarantowanie sobie przez Prawo i Sprawiedliwość możliwości wpływania na decyzje Państwowej Komisji Wyborczej.

Teraz pytanie do Prawa i Sprawiedliwości: W jaki sposób chcecie zagwarantować wzrost jakości przeprowadzanych przez PKW procesów wyborczych, skoro wszystkie wasze zmiany - co do jednej - które przeprowadziliście, zmiany personalne we wszystkich instytucjach państwowych, w sądownictwie, przyczyniły się tylko do pogorszenia jakości tych urzędów, do pogorszenia, jeśli chodzi o pracę w tych urzędach (Dzwonek), o osoby, które sprawują kluczowe funkcje w tych urzędach? Proszę, aby głos zabrała pani poseł Barbara Bartuś, przedstawiciel wnioskodawców. Dziękuję. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W punkcie, w którym są zadawane pytania, posłowie zadający te pytania mówili, że przecież wszystko jest jasne. Z drugiej strony z tych oświadczeń wygłoszonych tu przed momentem wynika, że państwo tak naprawdę macie wątpliwości co do tego, nad czym teraz procedujemy.

Kodeks wyborczy, który został przez Sejm uchwalony, i zmiany tego kodeksu, które zostały uchwalone i które obowiązują, zobowiązują Sejm m.in. do wyboru pięciu członków Państwowej Komisji Wyborczej.

Jest też mowa o proporcjonalności, o zgłaszaniu przez kluby.

Ale to postanowienie wydaje na podstawie uchwały Sejmu, uchwały przyjętej przez Sejm.

Osoby, które ten projekt uchwały składają, muszą napisać uzasadnienie, napisać, dlaczego chcą odwołania danego członka Państwowej Komisji Wyborczej. Sejm może podjąć taką uchwałę i zwrócić się do prezydenta o odwołanie tego członka Państwowej Komisji Wyborczej.

Żeby określić, że jest przestępstwo, to wcześniej musi być wyrok, który określa to przestępstwo, bo jeżeli jest podejrzenie, to nie ma jeszcze przestępstwa określonego, ktoś nie jest skazany za przestępstwo. Teraz mamy sytuację, że są uzasadnione obawy, że ktoś popełnił przestępstwo.

Bardzo dziękuję pani poseł Barbarze Bartuś, przedstawicielce wnioskodawców. Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu uchwały poprawki, proponuję, aby Sejm skierował ponownie ten projekt do Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 6. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druki nr 41 i 54) Proszę pana posła Henryka Kowalczyka o przedstawienie sprawozdania komisji. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu połączonych komisji: Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Komisje: Finansów Publicznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny po przeprowadzeniu pierwszego czytania rozpatrzyły projekt ustawy na posiedzeniu w dniu 11 grudnia. W trakcie dyskusji podnoszony był problem rezygnacji z kryterium przychodowego i pozostawienia tylko kryterium dochodowego w przypadku zastosowania małego ZUS-u.

Ostatecznie połączone Komisje: Finansów Publicznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny wnoszą o uchwalenie projektu ustawy wraz z przyjętymi poprawkami według treści zawartej w druku nr 54. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła.

Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawić stanowisko klubu wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Pan przewodniczący komisji Henryk Kowalczyk omówił zmiany zaproponowane do tej pory podczas procedowania nad tym dokumentem.

To jest dobra wiadomość dla osób, które uważały, że dzisiaj koszty związane z wejściem na rynek, prowadzeniem obrotu gospodarczego są bardzo duże.

Powstała koncepcja, żeby ją obniżyć.

Takie dane pokazuje nam ZUS w założeniach nowego projektu, który podnosi wielkość przychodów dającą uprawnienie do korzystania z tego obniżonego poziomu płacenia ZUS-u.

Polska dołączy w tym momencie do krajów Unii Europejskiej i krajów OECD, które mają w wielu przypadkach spiętą wysokość płaconych składek z osiąganymi przychodami. Tutaj w toku pracy nad tym dokumentem pojawiały się stanowiska, że trzeba mocniej spiąć to z dochodami z uwagi na fakt różnej marży w wielu branżach, w których uprawiają działalność przedsiębiorcy, na polu których osiągają swoje przychody i swój wynik gospodarczy. To jest niewątpliwie dobry kierunek. Przypomnę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości też miał odwagę obniżenia do najniższego w Europie podatku CIT od działalności gospodarczej dla podmiotów osiągających przychody mniejsze niż 1200 tys. euro. I to jest cały czas ten kierunek, którym chcemy zachęcić osoby do prowadzenia działalności gospodarczej, obniżyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Oczywiście zwracam tutaj uwagę na fakt, że niższa składka będzie powodowała również wyliczanie niższego świadczenia emerytalnego w przyszłości, o czym warto pamiętać, ale na to przyzwolenie i zgoda występują u tych osób, które dzisiaj dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą. Chcemy, żeby te mikrofirmy stawały się średnimi, średnie dużymi, żeby firmy rodzinne wzrastały bardzo szybko, żeby uzyskiwały lepszą pozycję, konkurencyjną na rynku usług. Bo właśnie ta regulacja, wydaje się, będzie mocno dopasowana do firm, które utrzymują się z tego, że świadczą usługi, że mają bardzo wysoką marżę. Mniej ona będzie korzystna dla tych podmiotów, które osiągają bardzo szybko wielkie przychody i czerpią korzyści z bardzo niskiej marży. A więc ona jest skierowana do małych zakładów usługowych, do zakładów naprawy sprzętu, do, myślę, prawników, do osób świadczących usługi doradcze. Miejmy nadzieję, że to jest początek też drogi w tym kierunku, że sytuacja finansów publicznych w Polsce będzie pozwalała na to, żeby tworzyć nowe, daleko idące programy, które będą jeszcze bardziej zachęcały osoby do aktywnego zachowania na rynku usług przy podejmowanej i prowadzonej z sukcesem działalności gospodarczej. Bardzo dziękuję panu posłowi. Proszę teraz o zabranie głosu pana posła Arkadiusza Marchewkę, który przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Na każdą propozycję, która zmniejsza obciążenia fiskalne wobec przedsiębiorców, należy spoglądać z uwagą. Należy na to patrzeć z uwagą, jednak należy wspierać przede wszystkim takie projekty, które dotyczą jak najszerszego grona polskich przedsiębiorców. To te osoby każdego dnia ciężko pracują i rzetelnie, sumiennie i uczciwie odprowadzają podatki. Rolą naszą jako parlamentarzystów i rolą państwa jest tworzenie odpowiednich warunków do ich rozwoju i działalności, a nie traktowanie ich jako maszynek do przynoszenia pieniędzy do kasy państwa.

Rok temu, kiedy o tym rozmawialiśmy, wielokrotnie pojawiały się te propozycje, jednak rząd tego nie chciał słuchać i okazało się, że zaledwie 180 tys. przedsiębiorców wyraziło wolę skorzystania. Ale ilu skorzystało, tego nie wiemy. Okazało się to niewypałem. Niestety nowa propozycja może w swoich założeniach jest w pewnych miejscach słuszna, ale z drugiej strony nie odpowiada potrzebom, które zgłaszają przedsiębiorcy w tak dużej skali, i jednocześnie można powiedzieć, że to góra urodziła mysz, dlatego że spośród 1200 tys. przedsiębiorców ten projekt obejmie zaledwie 320 tys. Oznacza to, że 3/4, czyli 75%, przedsiębiorców płacących każdego miesiąca składki na ZUS zostanie z tego wykluczonych. Czy to jest najlepsze rozwiązanie? Nie. Są rozwiązania, które są lepsze, które będą bardziej wspierać przedsiębiorców w prowadzeniu własnych biznesów i ułatwią im prowadzenie tych biznesów. Ważne jest to, aby po tych 2 latach czy 2,5 roku prowadzenia działalności przedsiębiorcy nie dostali od razu skokowej podwyżki składki ZUS, bo wielu może grozić zamknięcie ich biznesów, dlatego że nie będą po prostu w stanie na te składki zarobić.

Co proponujemy i co chcemy zrobić w tym zakresie? Proponujemy, aby podstawą naliczania składki ZUS nie było 60% przeciętnego wynagrodzenia, ale płaca minimalna. Oznacza to, że w przyszłym roku przedsiębiorcy nie zapłacą składek na ZUS i NFZ w wysokości 1444 zł, a 1261 zł. To prawie 200 zł korzyści i oszczędności.

Po drugie, proponujemy, aby ci, którzy są młodymi przedsiębiorcami, którzy dopiero rozpoczynają biznes, chcą wdrażać swoje kreatywne pomysły, byli zwolnieni z konieczności płacenia składek na ZUS i NFZ. Zaledwie 35% w grupie młodych ludzi pracuje, reszta jest nieaktywna zawodowo. Więc jeśli damy im możliwość zakładania własnych firm bez konieczności płacenia składek na ZUS i NFZ, nie będą się musieli obawiać, czy wystarczy im na prowadzenie własnej firmy. Więc jeśli się zaktywizują i będą z tych podatków zwolnieni, to lepiej dla nich, lepiej dla całej gospodarki. Trzecia kwestia dotyczy limitu przychodu. Propozycja rządowa zakłada 120 tys. przychodu dla tych, którzy mogą załapać się na tzw. mały ZUS+. Powinno się, według jego propozycji, zmienić przychód do 500 tys. zł, a później go całkowicie znieść, dlatego że niektórzy pomimo że mają duży przychód, mają równocześnie bardzo wysokie koszty, i nawet marżę bardzo niską, i mogą się na ten program po prostu nie załapać, a może się okazać, że ten program byłby też dla nich bardzo przydatny. A więc proponujemy również zwiększenie tego limitu do 500 tys. Bardzo dziękuję panu posłowi. Proszę teraz o zabranie głosu pana posła Tomasza Trelę, który zaprezentuje stanowisko klubu parlamentarnego Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Niewątpliwie program mały ZUS to był krok w dobrym kierunku, więc należy również program mały ZUS+ ocenić bardzo podobnie: to jest rozwiązanie, które pomoże przedsiębiorcom, i w tym przypadku będzie tych przedsiębiorców blisko 300 tys., a nawet ponad 300 tys.

Natomiast chciałbym zaproponować w imieniu klubu koalicyjnego Lewicy poprawkę, która zastępowałaby kwotę 120 tys. zł jako tę granicę, gdzie mały ZUS+ obowiązuje, i tę kwotę zastąpić krotnością najniższego wynagrodzenia za pracę. Chcę powiedzieć, że Lewica proponuje, aby była to 45-krotność najniższego wynagrodzenia. Natomiast będziemy mieli gwarancję i przedsiębiorcy będą mieli gwarancję, że im wyższe wynagrodzenie minimalne, tym ten próg kwotowy globalnie każdego kolejnego roku jest wyższy. A jak słyszeliśmy hurraoptymistyczne zapowiedzi pana posła Kaczyńskiego, już za 3, 4 lata ma być kwota 4 tys. zł najniższego wynagrodzenia, więc łatwo policzyć, że to by była już kwota 180 tys. zł. Więc stosowne poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, która w zasadniczym kształcie zamienia kwotę 120 tys. zł na krotność najniższego wynagrodzenia, pozwalam sobie złożyć panu marszałkowi. Oczywiście dwie kolejne poprawki są poprawkami pochodnymi, które muszą od strony formalnej również konsumować tę poprawkę i propozycję zasadniczą. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu posłowi. Proszę teraz panią poseł Agnieszkę Ścigaj o zabranie głosu w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15. Wysoka Izbo!

Jest to kontynuacja rok temu procedowanej ustawy o tzw. małym ZUS-ie, minimalnego kroku, nawet nie wiem, czy bardzo minimalnego, z szumnie zapowiadanej konstytucji dla biznesu, która niestety w dużej części nie została zrealizowana w ubiegłej kadencji, i nie zapowiada się, żeby w dużej części była realizowana. Ale niewątpliwie jest to krok właściwie konieczny, taki aby ulżyć małym firmom, małym przedsiębiorcom. Fakt, że skorzystało z tego 180 tys. działalności gospodarczych, świadczy o tym, że ta zmiana była w jakiś sposób potrzebna i konieczna. Prognozowana zmiana, czyli pójście dalej, poszerzenie tej grupy odbiorców do 320 tys., oczywiście jest zawsze krokiem do przodu, i dlatego nad tą ustawą się pochylamy i prawdopodobnie ją poprzemy, jeśli chodzi o całość klubu. Natomiast ma ona małe mankamenty i pewną rzecz obiecuje, natomiast o jednej bardzo ważnej rzeczy nie mówi. Wskazuje na kwotę, która w budżecie się pojawi, i ona będzie kosztować budżet.

Jeżeli ono pozostanie w wysokości 6 tys., to tak naprawdę będzie skierowane do tych, którzy właśnie mają tworzyć zapowiadaną klasę średnią i mają dociągać zarobki, więc uważamy, że jest on niepotrzebny. Oczywiście uważamy również, że kryterium obowiązywania czasowego jest kryterium, które też nie jest potrzebne, dlatego że jeżeli mówimy o firmach, które mają się rozwijać albo w jakiś sposób mają mieć te pieniądze na start, to mamy jedną ulgę związaną z krótkim, 2-letnim czasem startowym.

Oczywiście chcę powiedzieć, że kompleksowe rozwiązanie to jest rozwiązanie, które zaproponowaliśmy w ustawie, gdzie klub Koalicji Polskiej - Polskiego Stronnictwa Ludowego - Kukiz15 złożył projekt, który jest powszechnie akceptowany, sprawdzony w innych krajach, dobrowolnego ZUS-u. Uważamy, że 20 lat płacenia przez przedsiębiorcę to jest sprawiedliwe płacenie tak samo, jak każdy inny pracownik w Polsce. 20 lat, a w pozostałe lata możliwość inwestowania w rozwój własnej firmy, odkładania we własny sposób, ponieważ mówimy o ludziach przedsiębiorczych, o ludziach, którzy potrafią gospodarować własnymi pieniędzmi, obracać złotówką z korzyścią dla gospodarki, dla własnej rodziny i dla własnej przyszłości.

Dziękuję bardzo, pani poseł. Teraz proszę pana posła Jakuba Kuleszę, który przedstawi stanowisko Koła Poselskiego Konfederacja. Wysoka Izbo! Z przykrością muszę powiedzieć, że najmniejsi przedsiębiorcy, pomimo tej całej propagandy rządowej, nie są beneficjentami dobrej zmiany, są w zasadzie jej ofiarami. Przez kolejne utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej małe i mikroprzedsiębiorstwa stają się najbardziej gnębioną grupą społeczną. JPK, split payment, biała lista podatników, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, STIR, BDO to tylko niektóre wynalazki obecnego i poprzedniego rządu, którym podlegają tak samo duża firma i korporacja, jak i najmniejsza, nawet jednoosobowa, działalność gospodarcza. Prezes Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, pani minister Emilewicz często na konferencjach prasowych w kampanii wyborczej opowiadali, jakie to ulgi, preferencje przedstawiają, wprowadzają dla małych i mikroprzedsiębiorców. Tymczasem mamy coraz większe koszty prowadzenia działalności gospodarczej, coraz więcej obowiązków i coraz więcej kar z nich wynikających. Prowadzenie nawet najprostszej działalności gospodarczej w Polsce staje się bardziej ryzykowne niż zawodowa działalność przestępcza. Tu nie potrzeba żadnych ulg, żadnych by-passów, żadnych pasów startowych, żadnych plusów, minusów, zwolnień, które są tworzone tak, że może z nich skorzystać zaledwie kilka procent firm w Polsce. Tu potrzeba gruntownej zmiany, dlatego domagamy się zmiany całego systemu ubezpieczeń społecznych przedsiębiorców, najlepiej na system dobrowolny, jaki jest w krajach Europy Zachodniej, np. u naszego sąsiada, w Niemczech. Wracając do ustawy mały ZUS, kogo będzie dotyczyć projekt? Niestety zaledwie kilku mikro- i małych przedsiębiorców, w zasadzie tylko mikro-, bo mali się już nie łapią, natomiast 90% przedsiębiorców od przyszłego roku zapłaci wyższy ZUS.

Rozumiem, że nie zmienimy dzisiaj całego systemu na jakiś uczciwy, najlepiej dobrowolny, ale przyjmijmy dzisiaj, że zostawiamy tylko kryterium dochodowe, a likwidujemy absurdalne kryterium przychodowe 10 tys. zł, co jest absurdalnie niską kwotą. Nawet kiosk Ruchu czy warzywniak nie jest w stanie przetrwać na rynku, mając tylko 10 tys. przychodu. Przychodu, nie dochodu, bo to bardzo często niektórym politykom, także ministrom, się myli. Projekt ten całkowicie dyskryminuje jakąkolwiek działalność handlową. Aby osiągnąć dochód na poziomie 5 tys. zł, inny przychód należy wypracować w branży usługowej, inny w handlowej, a jeszcze inny w produkcyjnej. Z małego ZUS według rządowego projektu mogłaby skorzystać co najwyżej część działalności usługowej. Wreszcie należy zlikwidować zupełnie niezrozumiałe ograniczenia obowiązywania małego ZUS-u do 3 lat. Ktoś, kto przygotował ten projekt i wstawił tak bzdurny warunek, nigdy nie prowadził działalności gospodarczej. Znaczna większość działalności mikro- czy małych przedsiębiorców jest prowadzona w skali, z której dochody mają zaspokoić potrzeby rodziny przedsiębiorcy. Taki przedsiębiorca pracuje na własny rachunek i nie ma ambicji stać się Orlenem czy Amazonem. Państwo zmusza go, aby pracował coraz więcej, rósł i przekształcał się w coraz większą firmę, zmusza go do tego, stosując karę od początku czwartego roku działalności, czyli podwyżkę ZUS o prawie 300%. To godzi w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy sami powinni decydować, czy chcą się rozwijać i rosnąć, czy chcą pozostawać małą firmą, a tu państwo narzuca przedsiębiorcom, jak mają funkcjonować.

Nie może być tak, że przedsiębiorca, który nie był w stanie zapłacić wysokich składek ZUS, wyrzucany jest z mieszkania, razem z rodziną ląduje pod mostem, komornik na zlecenie ZUS-u licytuje, sprzedaje to mieszkanie i wpłaca pieniądze na konto ZUS-owskie tego przedsiębiorcy po to, żeby miał zapewnioną emeryturę. To jest chory system. To jest podobno składka na własną emeryturę w przyszłości, nie może więc być ona tak ogromnym obciążeniem, które uniemożliwia normalne funkcjonowanie.

Dziękuję bardzo panu posłowi.

Zamykam listę, ustalając jednocześnie czas na zadanie pytania na 1 minutę. Proszę o zabranie głosu pana posła Michała Szczerbę, Koalicja Obywatelska. Nie ma.

Jeżeli chcemy rozmawiać o tym projekcie, to myślę, że ze wszystkich stron jest wiele krytyki i opinii o słabych stronach tego projektu. Po pierwsze, dochód - w tym zakresie mówimy o przychodzie, a nie o dochodzie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej przez podatników. Takie rozwiązanie nie do końca satysfakcjonuje i w nierówny sposób traktuje podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą.

To rozwiązanie niestety nie spełnia oczekiwanego warunku.

Dziękuję bardzo, pani poseł. Proszę o zabranie głosu panią poseł Joannę Frydrych, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Projekt ustawy zakłada rozszerzenie katalogu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą uprawnionych do obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne. W konsekwencji spowoduje to mniejsze wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Czy rząd, składając ten projekt ustawy, pomyślał o wysokości przyszłych emerytur przedsiębiorców korzystających z tej ulgi? Czy rząd zagwarantuje im minimalną emeryturę w przyszłości? Jeżeli tak, to gdzie jest ten zapis gwarantujący tę minimalną emeryturę? Czy rząd szacował, o ile niższe będą świadczenia osób, które skorzystają z tej pułapki emerytalnej? Bo można tak to nazwać? Czy rząd zamierza przeprowadzić kampanię informującą, że skorzystanie z tej ulgi będzie wiązało się nie tylko z niższymi emeryturami w przyszłości, ale także z niższymi świadczeniami chorobowymi i macierzyńskimi już w 2020 r. Proszę o zabranie głosu panią poseł Annę Wasilewską, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Po pierwsze, czy były prowadzone jakiekolwiek badania, jak zmiana ta wpłynie na przedsiębiorców? Czy rząd ma świadomość, że zaburzy tym konkurencyjność małych firm? Czy rząd wie, że już jest grudzień i przedsiębiorcy do dzisiejszego dnia nie wiedzą, jaką składkę będą płacili od stycznia 2020 r. Dlaczego w odniesieniu do małego ZUS-u wykluczeni zostali przedsiębiorcy rozliczający się w inny sposób niż na podstawie zasad ogólnych PIT? Dziękuję bardzo, pani poseł. Proszę o zabranie głosu pana posła Mirosława Suchonia, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Muszę powiedzieć, że prawdopodobnie w ministerstwie nie ma osoby zdroworozsądkowej, która ma doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Gdyby taka osoba była i prowadziła już wspomniany tutaj choćby kiosk Ruchu czy kiosk z warzywami, to doskonale zdałaby sobie sprawę z tego - i, myślę, oświeciła pracowników ministerstwa, rząd - że to jest kwota, która nie ma nic wspólnego z realną pracą, z realnym dochodem przedsiębiorców, którzy (Dzwonek) wykonują swoją działalność. Dlatego mam pytanie do ministerstwa: W jaki sposób została ta kwota wyliczona i czy prawdą jest, że chodziło o to, żeby ograniczyć, jak najbardziej ograniczyć, grupę przedsiębiorców, która mogłaby skorzystać z tego mechanizmu? Proszę pana posła Arkadiusza Marchewkę o zadanie pytania. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Wielokrotnie w wypowiedziach premiera i przedstawicieli rządu PiS słyszeliśmy o tym, że wspierane jest duże grono przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy, że ułatwia im się prowadzenie tych działalności gospodarczych, tymczasem popatrzmy na fakty.

W jaki sposób rząd zamierza to zmienić i poprawić tę sytuację? Jak się okazuje, propozycja przygotowana przez rząd, czyli mały ZUS+, będzie trafiała tylko do wąskiego grona polskich przedsiębiorców. To trzeba rozszerzyć i realnie wesprzeć tych, którzy każdego dnia ciężko pracują i uczciwe płacą podatki. Dziękuję bardzo panu posłowi.

Wysoka Izbo! Nie było mnie tu parę lat i ze zdziwieniem zauważyłam, że w systemie emerytalnym grzebią sobie jak kura pazurem wszyscy, którzy się na tym doskonale znają, najbardziej minister gospodarki, małych, średnich przedsiębiorstw, dużych i większych, i mniejszych, itd. Podatków w tym kraju jest od groma, ulgi można sobie ustalić, jakie się chce, ale system emerytalny jest po to, żeby zabezpieczyć również tego przedsiębiorcę na starość, żeby on po prostu miał emeryturę.

Bardzo dziękujemy, pani minister.

Wysoka Izbo! Ten projekt zmian przedstawia jak w soczewce, w jaki sposób rząd Prawa i Sprawiedliwości traktuje przedsiębiorców.

Dlaczego państwo np. nie zaproponują dobrowolnej składki ZUS dla samozatrudnionych przedsiębiorców? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu posłowi. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Taki projekt został przez Polskie Stronnictwo Ludowe w ubiegłej kadencji złożony.

Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana posła Wiesława Janczyka, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Wydaje mi się, że uciekło nam w dyskusji coś, co jest może szczegółem, ale wyjątkowym.

Dziękuję bardzo. Listę posłów zadających pytania zamyka pan poseł Marek Sowa, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Największą słabością tego przedłożenia jest kwestia zabezpieczenia emerytalnego właśnie tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, bo nie jest tak, jak mówił poseł Jończyk.

Takie są zapisy tej ustawy, takie są po prostu realia.

Bardzo dziękuję panu posłowi. Na zadane pytania odpowie pan minister Marek Niedużak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Wysoka Izbo!

Absolutnie jest tak - i za każdym razem my to powtarzamy, i to jest niezwykle istotny element tego projektu - że on oznacza wyjątek od zasad ogólnych i obniżkę składek na ubezpieczenie społeczne, która pociągnie za sobą - oczywiście - niższą emeryturę. I to wszyscy wiemy, musimy mieć tego świadomość. Teraz z jednej strony słyszę głosy, które mówią: czemu ta obniżka nie ma szerszego zasięgu, nie jest większa, po co ten limit. A z drugiej strony pojawia się głos o zabezpieczeniu emerytalnym. Jeden interes to jest wysokość składki tu i teraz, a drugi interes to jest emerytura w przyszłości. I właśnie dlatego ten projekt jest - wyrażenie, którego użyję - skalibrowany. On jest skalibrowany z jednej strony w ten sposób, że bierze pod uwagę koszty dla budżetu, który będzie musiał pokryć ubytki w funduszu ze względu na to, że wpłynie tam mniej składek, a z drugiej strony w ten sposób, aby objąć kilkaset tysięcy polskich przedsiębiorców. Wiadomo, że to są jednoosobowe działalności, więc tylko o tych tutaj mówimy. Wydaje mi się, że wprowadzanie ulgi, wyjątku dla najmniejszych kilkunastu procent to nie jest projekt dla nikogo albo projekt dla kilku podmiotów. Przynajmniej w moim słowniku trzysta kilkadziesiąt tysięcy podmiotów to nie jest kilka podmiotów. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz też się tutaj pojawiała wielokrotnie. Przychód jako kryterium.

Definicja MŚP, przyjęta w prawie europejskim, a zatem recypowana do naszego prawa, opiera się właśnie na kategorii nie dochodu, tylko obrotu, sprzedaży, przychodu. i na liczbie pracowników, oczywiście. To są kryteria obiektywnie mówiące o tym, czy dana firma jest duża, czy mała. To jest rozwiązanie dla firm najmniejszych i dlatego tutaj kryterium wejściowym, tym limitem, jest limit przychodu. Nie ma w ustawie limitu dochodu - to się też tutaj miejscami pojawiało w niektórych wypowiedziach. Limit dochodu, o którym czasami mówi się w debacie, wynika tylko i wyłącznie z tego, że ta proporcjonalność przestaje się opłacać i opłaca się przejście na ryczałt. I nie ma tego twardo napisanego w przepisach: że to jest limit dochodu, dla którego masz prawo skorzystać z tej ulgi. Jest proporcjonalność, która w pewnym momencie dochodzi do takiego poziomu, że opłaca się wyjść z proporcjonalności i wejść na ryczałt na zasadach ogólnych. W ustawie jest tylko limit przychodowy, przed chwilką starałem się wytłumaczyć dlaczego. Trzy na pięć. Bo też jeszcze raz zaznaczę: to jest możliwość, prawo. Ludzie, którzy są przedsiębiorcami, z definicji są osobami, które akceptują wyższy poziom ryzyka niż osoby, które są zatrudnione na etacie, i muszą się też z tym ryzykiem liczyć, jeżeli wybierają taką opcję.

Jeżeli zniesiemy ten limit, to nie będzie miała takiej szansy. Tak się składa, że np. w Niemczech teraz toczy się dyskusja właśnie na ten temat, żeby się z tej dobrowolności dla przedsiębiorców wycofać. Proszę też pamiętać, że w Niemczech jest zupełnie inna skala samozatrudnienia, to jest po prostu inna gospodarka. Z kolei w Anglii, którą też troszeczkę znam, jest tak, że owszem, są niskie składki dla przedsiębiorców, ale ta emerytura, która przysługuje, przypomina coś, co należałoby w Polsce chyba nazwać bardziej taką emeryturą z budżetu, państwową.

Więc proszę się też nie powoływać na wybiórczo traktowane rozwiązania, które gdzieś tam funkcjonują w zupełnie innym kontekście niż nasz. Dlaczego to obejmuje taką, a nie inną liczbę przedsiębiorców?

Oczywiście, że w jego przypadku była współpraca ZUS-u, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwa Finansów.

Padło też pytanie o czas wejścia w życie. Ja jako skromny podsekretarz stanu mogę powiedzieć, że akurat termin wejścia w życie w gruncie rzeczy zależy od państwa, od posłów i senatorów, tak?

Proszę też pamiętać, że mówimy nie o zasadach ogólnych, tylko o pewnym wyjątku, i to takim pozytywnym, o pewnym uprzywilejowaniu, tak? A więc na zasadach ogólnych ten system nie jest tutaj zmieniany i przedsiębiorcy wiedzą, jak te zasady ogólne wyglądają i będą wyglądać w przyszłym roku.

Nie jest też prawdą, że jest to rozwiązanie oferowane tylko i wyłącznie podatnikom rozliczającym się na zasadach ogólnych, ponieważ są tutaj też rozwiązania dla ryczałtowców, czyli rozliczających się podatkiem zryczałtowanym, a także tzw. kartowców.

Stąd ta korzyść tutaj po ich stronie. Wydaje mi się, że to są te najważniejsze kwestie. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu przedstawienia sprawozdania. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Chciałabym prosić o przywitanie młodej pacjentki Centrum Zdrowia Dziecka, która dzisiaj gości u nas w Sejmie. Maja, niezwykle dzielna młoda dama. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 7. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druki nr 44 i 52) Proszę panią poseł Annę Milczanowską o przedstawienie sprawozdania komisji. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, druk nr 44. Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu, skierowała w dniu 4 grudnia 2019 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Infrastruktury do pierwszego czytania. Komisja Infrastruktury po przeprowadzeniu pierwszego czytania, rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2019 r. wnosi, by Wysoki Sejm raczył uchwalić projekt ustawy z druku nr 44 bez poprawek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani poseł. Otwieram dyskusję. Jako pierwsza głos zabierze pani poseł Anna Milczanowska, prezentując stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, druk nr 44. Rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął wyzwanie zwalczania pogłębiającego się zjawiska wykluczenia komunikacyjnego, dotyczącego w szczególności terenów oddalonych od dużych ośrodków miejskich. Ten przejaw patologii życia społecznego postanowiono zwalczać m.in. za pomocą przeprowadzanej reformy. Jednym z jej mechanizmów jest ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dzięki niej poprzez dofinansowanie udało się przywrócić wiele lokalnych linii autobusowych. Obecnie prowadzone są prace legislacyjne mające na celu kontynuację procesu rozwoju połączeń lokalnych. Do czasu ich zakończenia istnieje potrzeba przedłużenia terminu obowiązywania przepisów przejściowych ustawy o publicznym transporcie zbiorowym o kolejny rok. Powyższe przedłużenie obowiązywania przepisów przejściowych pozwoli na dostosowanie ich do założeń ustawy budżetowej na rok 2020. Niewprowadzenie powyższych zmian prowadziłoby do przyjęcia odmiennej od zawartej w ustawie budżetowej struktury dysponentów odpowiedzialnych za finansowanie ulg. Przepisy, które w okolicznościach nieuchwalenia niniejszego projektu ustawy zaczęłyby obowiązywać, prócz tego, iż zawierają odmienny od obecnego system finansowania ulg, budzą również wątpliwości interpretacyjne. Utrzymanie obecnego systemu dotowania umożliwi większą kontrolę środków przeznaczanych na ten cel i zapewni finansowanie tego zadania na odpowiednim poziomie. Jednocześnie brak jest obiektywnych danych umożliwiających ocenę skutków realizacji postanowień ustawowych i zapewniających realizację pokładanych w przedmiotowych przepisach oczekiwań społecznych w przypadku nieprzedłużenia okresu przejściowego stosowania ustawy.

Dziękuję, pani poseł. W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska głos zabierze pan poseł Franciszek Sterczewski. Proszę bardzo.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jestem zaszczycony, że moje pierwsze wystąpienie mogę poświęcić tematowi, który jest mi szczególnie bliski, czyli komunikacji zbiorowej, tym bardziej że wypowiadam się odnośnie do projektu rządowego, dzięki czemu mogę zwrócić się bezpośrednio do tych, którzy decydują, w jakich warunkach podróżują Polki i Polacy. Niedawno premier Morawiecki w swoim exposé powiedział wiele o zrównoważonym transporcie. Brak autobusu czy pociągu w pobliżu miejsca zamieszkania dla wielu ludzi oznacza brak dostępu do szkoły, szpitala czy pracy. To jest problemem dla ok. 14 mln osób wykluczonych komunikacyjnie. Każda nowa linia kolejowa czy autobusowa jest więc przywróceniem nadziei i godności tym, którzy zostali jej pozbawieni przez krótkowzroczne i nieodpowiedzialne decyzje podjęte w przeszłości.

Uważam, że możemy w jasny sposób określić, w czym się różnimy, a w czym się zgadzamy. Naszym wspólnym celem jest stworzenie takiej komunikacji zbiorowej, z której wszyscy korzystalibyśmy z przyjemnością. Kiedy więc usłyszałem słowa pana premiera, uznałem, że oczywiście będę popierał wszystkie słuszne działania w tej sprawie, niezależnie od tego, czy zgadzam się z tym rządem w innych obszarach. Problem w tym, że na razie wiemy niewiele. Pytanie brzmi: Skąd właśnie taka liczba? Cieszę się, że premier zwrócił uwagę na ten problem, i liczę na to, że program „Kolej+” nie będzie pisany palcem po wodzie tak jak „Mieszkanie+” O tramwajach nie wspomniał pan premier ani słowem, choć sporo miejsca poświęcił samochodom, a także kontrowersyjnym, bizantyjskim projektom, takim jak Centralny Port Komunikacyjny. W każdym razie ustawa, o której dzisiaj rozmawiamy, jest dalszym ciągiem tej samej niekonsekwencji. Pod pretekstem przygotowanej reformy komunikacji zbiorowej rząd odracza unormowanie systemu finansowania ulg na bilety kolejowe i autobusowe. Ta nowelizacja początkowo miała wejść w życie w 2017 r., a co roku jest odraczana. Szanowni państwo, ile jeszcze lat będziemy czekali na wejście w życie tych regulacji? Czy możemy usłyszeć jakąś konkretną datę? Warto podkreślić, że ustawa jest odraczana w polskim parlamencie po raz czwarty, co samo w sobie powinno być dla rządzących wystarczającym powodem do wstydu. Jest 12 grudnia, a rząd dopiero teraz rozpoczyna dyskusję o tym, co wydarzy się za niespełna 3 tygodnie.

Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie pokazywało, że nie ma pomysłu na to, w jaki sposób reformować transport. Zamiast całościowych reform otrzymujemy fragmentaryczne rozwiązania i próby doraźnego uporania się z chaosem. Z kolei odrzucenie tego wniosku oznaczałoby bałagan organizacyjny w samorządach i zablokowanie transportu publicznego poza miastami, co byłoby katastrofą dla pasażerów i pasażerek. Zatem w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni rekomenduję wstrzymanie się od głosu. Przy okazji chciałbym zwrócić uwagę na temat poznański, czyli na dworzec PKP Poznań Główny, który od lat wymaga usprawnienia i przywrócenia mu świetności. W tym momencie jest obiektem kpin i parodią dworca. Liczę, że pan premier odpowie mu w krótkim czasie. Poza tym wszystkim chciałbym, żebyśmy mieli takie małe postanowienie noworoczne. Od 1 stycznia wróćmy do tej ustawy i innych ustaw dotyczących autobusów czy kolei i zacznijmy wreszcie na poważnie rozmawiać o komunikacji zbiorowej. Szanowni Państwo! W imieniu klubu parlamentarnego Lewica głos zabierze pani poseł Paulina Matysiak. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu parlamentarnego klubu Lewicy mam zaszczyt przedstawić opinię na temat rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Funkcjonująca od niemal 10 lat ustawa o publicznym transporcie zbiorowym nie powstrzymała zapaści transportu publicznego na obszarach pozamiejskich w Polsce. W ostatnich latach liczba użytkowników autobusowej komunikacji poza miastami ulega systematycznemu spadkowi, a w ślad za nim ograniczeniu ulega oferta przewoźników. Tylko w tym roku zawieszono bądź zlikwidowano 340 połączeń autobusowych, na takich liniach jak: Skępe - Lipno, Łódź -Lutomiersk - Szydłów - Łódź, Chełmno - Świecie. To jest tylko kilka wybranych przykładów. Gminy, w których nie istnieje organizowana przez samorząd komunikacja lokalna, zamieszkuje dziś aż 14 mln osób. Jeżeli ktoś nie posiada własnego samochodu, a w jego miejscowości nie istnieje czynny przystanek kolejowy, to skazany jest na łaskę albo niełaskę prywatnych przewoźników autobusowych. Tymczasem sprawny transport zbiorowy poza miastami jest kluczowym czynnikiem dla zrównoważonego rozwoju regionalnego. Umożliwia aktywizację mieszkańców terenów o wysokim bezrobociu, daje dostęp do szkół zwiększających szansę na rynku pracy, dostęp do placówek medycznych, miejsc handlu i usług czy wreszcie instytucji publicznych i kultury. Społeczeństwo dobrze skomunikowane wolne jest od barier, granic i ograniczeń. Brak dobrego transportu publicznego prowadzi nieuchronnie do wykluczenia wszystkich mieszkańców obszarów pozamiejskich pozbawionych możliwości korzystania z samochodów, osób o ograniczonej sprawności, dzieci i młodzieży, a także osób niezamożnych. Jest to wykluczenie nie tylko transportowe, ale i ekonomiczno-społeczne. Nie można mówić o żadnej powszechności oświaty, opieki zdrowotnej, kultury i ekonomicznego dobrobytu, jeżeli miliony ludzi są pozbawione transportu, żeby z nich skorzystać. Wykluczenie transportowe ogranicza możliwość podjęcia pracy, bo trzeba do niej często dojeżdżać, tak samo jak możliwość skorzystania z oferty takiej jak kino, teatr czy muzeum. Nawet swobodne spotkania z rodziną i znajomymi stają się luksusem, na który nie każdy może sobie pozwolić. Miliony Polek i Polaków są pozbawione podstawowej opieki medycznej w sytuacji, kiedy nie mogą dojechać do przychodni lub szpitala. Odkładanie w nieskończoność zmian w ustawie nie rozwiązuje żadnego z chronicznych problemów publicznego transportu zbiorowego w Polsce, a konserwuje obecny system oparty, w dużym uproszczeniu, na prowadzeniu przewozów w sposób rynkowy. Skomplikowany i nietransparentny system finansowania przewozów poprzez dopłaty do ulg prowadzi z jednej strony do niegospodarności w postaci dotowania nawet najbardziej rentownych połączeń, a z drugiej - do szeregu patologii, jak sztuczne zawyżanie cen czy sprzedawanie biletów ze 100-procentową ulgą w celu uzyskania większej refundacji. Organizacja transportu zbiorowego na podstawie zezwolenia na przewóz w połączeniu z jego finansowaniem z poziomu urzędów marszałkowskich pozbawia powiaty i gminy jakiegokolwiek wpływu na siatkę połączeń, częstotliwość kursów czy jakość taboru. Niejasny podział i rozproszenie kompetencji pomiędzy poszczególne poziomy samorządu prowadzi do braku szerszej wizji organizacji transportu publicznego, niechęci do współpracy i wreszcie rozmycia odpowiedzialności za zwalczanie wykluczenia transportowego na terenach pozamiejskich. Niestety ani odkładane dziś po raz czwarty przepisy przejściowe ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ani przygotowane na kolanie przez Ministerstwo Infrastruktury kolejne projekty ustawy nie rozwiążą żadnego ze wspomnianych problemów. Powierzchowne i chaotyczne podejście partii rządzącej do problematyki publicznego transportu zbiorowego prowadzi do coraz większej degradacji przewozów autobusowych na terenach pozamiejskich. Koszt tego poniosą miliony mieszkańców miast i wsi, którzy pozbawieni nawet minimalnej oferty przewozowej będą nadal zmagać się z wykluczeniem transportowym. Na zdecydowaną krytykę zasługuje także to, w jakim trybie ten projekt jest procedowany.

Jeśli nie zostanie podpisany przez prezydenta do 31 grudnia, od Nowego Roku ważność stracą wszystkie zezwolenia na przewóz osób w transporcie drogowym, czyli realnie w trasy nie wyruszą żadne autobusy. W niecały miesiąc projekt więc musi zostać zaakceptowany przez Sejm, Senat i prezydenta. Tryb procedowania jest gorszący, a tak późny termin przesłania projektu ośmiesza Ministerstwo Infrastruktury i cały rząd. Lewica zagłosuje jednak za przyjęciem tego projektu (Dzwonek), ponieważ jest odpowiedzialna. Nawołujemy więc rząd do poważnego potraktowania problemu wykluczenia transportowego i przygotowania zmian poprawiających jakość i dostęp do transportu zbiorowego. Dziękuję bardzo, pani poseł.

Wysoka Izbo!

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym przedłożony przez ministra infrastruktury, który to projekt był przedmiotem obrad Komisji Infrastruktury.

Do końca 2020 r. przedłużone zostaną także zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów autobusowych, realizowanych przez przewoźników komercyjnych. Obecny termin upływa w 2019 r. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia i 1 stycznia możemy obudzić się w kraju pozbawionym transportu publicznego, ponieważ z końcem roku tracą ważność zezwolenia na przewóz osób w transporcie drogowym. Jeśli nawet uda się wygrać z czasem, problem może dotyczyć biletów ulgowych. Do końca roku mamy jedno posiedzenie Sejmu: dzisiaj i jeszcze 19 i 20 grudnia. Posłowie muszą się więc spieszyć, bo Senat będzie obradował 17 i 18 grudnia. Jeśli któryś z tych elementów zawiedzie, pasażerowie będą mieli problem. Ważność stracą wszystkie zezwolenia na przewóz osób w drogowym transporcie, nie wyjedzie zatem żaden prywatny autobus, o ile wcześniej dany przewoźnik nie złożył wniosku o wydanie potwierdzenia zgłoszenia przewozu. Problem w tym, że nikt do tej pory takich wniosków nie składał, ponieważ ich ważność również jest związana z ww. przepisami. Niezależnie od tego, kiedy wnioski zostały złożone, pierwszy dzień ich obowiązywania to pierwszy dzień obowiązywania nowych przepisów.

Rząd zapewnia, że pieniądze na finansowanie ulg są i że zostały zapisane w projekcie budżetu, ale przyznaje jednocześnie, że jeżeli ustawa nie przejdzie, to nie będzie można w ten sposób finansować ulg. Brak tych przepisów oznaczałby konieczność przyjęcia odmiennej od zawartej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 struktury dysponentów odpowiedzialnych za finansowanie ulg - czytamy w uzasadnieniu. Rząd wskazuje, że uchwalenie ustawy oznacza, że 312 mln pasażerów w transporcie drogowym i 301 mln pasażerów kolei, czyli inaczej mówiąc: wszyscy ci, którzy korzystają z autobusów lub kolei, będą nadal mogli korzystać z ulg. Rząd wskazuje także, że nastąpi przedłużenie obowiązujących przepisów o rok, do czasu dokończenia reformy publicznego transportu zbiorowego. Jednak jest to już czwarte takie odroczenie. Nasuwa się więc pytanie, czy rząd, który miał wspierać transport publiczny, wspiera ten transport, czy czyni zupełnie na odwrót. Czy pomysł wsparcia samorządów w staraniach o przywrócenie lokalnych połączeń okazał się nietrafiony, czy znowu winą obarczycie samorządy, które nie chcą korzystać z dopłat państwa, bo brakuje im pieniędzy na wkłady własne?

Samorządy niechętnie korzystają z tego funduszu - pokazują to kolejne nabory - bo po prostu nie mają pieniędzy.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Uprzejmie informuję, iż do pytań zapisało się 11 osób. Zamykam listę. Jako pierwsza. Staram się nie odbierać głosu, jeśli rzeczywiście pytanie jest merytoryczne. Jako pierwsza pytanie zada pani poseł Beata Maciejewska, Lewica. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! W zeszłym tygodniu w odpowiedzi na prośbę wyborców z mojego okręgu złożyłam interpelację poselską dotyczącą białych plam komunikacyjnych, które stały się szczególnie istotnym problem na terenie Pomorza. Przykładem są Główczyce w powiecie słupskim, gdzie niedawno tamtejszy PKS zlikwidował część kursów, co spowodowało, że mieszkańcy mają problemy z dojazdem do miejsca pracy. Jak mówią samorządowcy, dopłaty nie zachęcają przewoźników do tworzenia nowych połączeń, gdyż te wciąż pozostają dla nich zbyt kosztowne i problematyczne. Co więcej, nie każda gmina czy nie każdy powiat mogą sobie pozwolić na wymagany wkład własny.

Dziękuję bardzo, pani poseł. Pan poseł Ryszard Wilczyński, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Panie Ministrze!

To bardzo ciekawy przykład i jego analiza prowadzi do jedynego możliwego wniosku.

O to w istocie chodzi. Natomiast państwo cały czas uważacie, że najważniejsze jest, żeby odjechał autobus. Nie o to chodzi. I samorządy wam oczywiście nie uwierzyły, bo pieniądze zostały niewykorzystane. No i ta piątka, ten ostatni z punktów piątki Kaczyńskiego jest klapą. Proponuję uratować ten program (Dzwonek) - poproszę o pół minuty, pani marszałek - a mianowicie zrobić program rządowy, w którym dajecie pieniądze na innowacje w transporcie publicznym, po prostu, żeby zastosować mechanizmy znane z rozwiązań typu smart, smart village, smart city, i sprawdzić, gdzie co się uda.

Ale jednak zwracam uwagę, że jesteśmy na etapie pytań. Pytań. To nie było wystąpienie klubowe.

Wysoka Izbo! Panie Premierze! Panie Ministrze! W uzasadnieniu do omawianego projektu jest mowa o dokończeniu toczących się prac legislacyjnych w zakresie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego. I stąd to przesunięcie, o którym dzisiaj rozmawiamy. Panie Ministrze! Kiedy więc - i proszę tutaj o wskazanie konkretnego miesiąca i konkretnego roku - parlamentarzyści będą mogli zapoznać się z przygotowanymi rozwiązaniami? Jeżeli pan minister nie jest dziś przygotowany do odpowiedzi na to pytanie, to poproszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Omawiany projekt został złożony przez rząd 4 grudnia, czyli mniej niż miesiąc przed planowanym wejściem w życie zawartych w nim przepisów. Jeśli ustawa nie wejdzie w życie przed końcem roku, ulgi ustawowe na przejazdy autobusami pozamiejskimi mogą po prostu zniknąć. W związku z tym mam pytanie: Co rząd zamierza zrobić, jeżeli parlamentowi nie uda się uchwalić ustawy do końca bieżącego roku? Przypominam, że czekają nas prace legislacyjne nad niniejszym projektem w izbie wyższej, a później ustawa musi jeszcze trafić na biurko prezydenta i zostać przez niego podpisana. Czy w obliczu tak poważnego ryzyka pogłębienia wykluczenia komunikacyjnego Ministerstwo Infrastruktury przygotowało jakikolwiek plan B? Pragnę również zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z czwartym już odroczeniem wejścia w życie bardzo ważnych przepisów dotyczących organizacji i finansowania pozamiejskiego transportu publicznego, przepisów, które zostały uchwalone, przypominam, już 9 lat temu. Gorąco apeluję, aby w przyszłości ministerstwo nie zajmowało się tak ważnymi sprawami dosłownie w ostatniej chwili. Dziękuję. Pan poseł Mirosław Suchoń, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Wysoka Izbo! Oczywiście ustawa musi zostać przyjęta, ponieważ groziłby wszystkim paraliż dotyczący finansowania ulg. Panie ministrze, podziwiam, szczerze mówiąc, ten optymizm wynikający z czasu złożenia tego projektu, ponieważ ustawa musi zostać przeprocedowana przez Senat, później podpisana przez prezydenta. Pan prezydent zwykł podpisywać w zasadzie bezzwłocznie wszystko, co trafia na biurko. Mam pytanie dotyczące przewozów autobusowych. W zeszłym roku, w poprzedniej kadencji został przyjęty projekt ustawy, która reguluje dopłaty do przewozów.

Drugie pytanie: Czy rzeczywiście zaplanowana kwota na rok 2020 wynosi 800 mln zł? Jaka to jest na podstawie wniosków kwota? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Wysoka Izbo! Mam w zasadzie dwa pytania. Wszyscy wiemy, że samorządy, chociażby te, które obsługują ulgi, dopłaty do biletów ulgowych, już szykowały się na zmiany organizacyjne we własnych urzędach, na przeniesienie etatów, na zmniejszenie kwot, które przeznaczały na to zadanie.

Każdy, kto pracował w samorządzie, wie, że zadania, nie tylko te zadania, ale wiele innych, zawsze pochłaniały więcej środków niż było przeznaczane ze środków budżetowych przez państwo, przez rząd. Dziękuję. Pani poseł Anna Milczanowska, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Panie Ministrze!

Panie Ministrze!

Dziękuję bardzo, pani poseł. Pani poseł Gabriela Masłowska, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Kiedy przysłuchuje się tego typu dyskusji, tym lamentom, jak to jest bardzo źle z komunikacją publiczną w Polsce na obszarach wiejskich. i w ogóle, że Polacy są odcięci od świata itd., to nieustannie nasuwa mi się pytanie odnośnie do genezy tego stanu rzeczy: Jaka jest przyczyna tego stanu rzeczy? Pamiętacie państwo chyba, jak problem transportu publicznego był rozwiązany. Pytam: Co się z nimi stało? W jakich latach zostały one zniszczone, sprywatyzowane? Mam swoje doświadczenia, jeśli chodzi o województwo lubelskie. Sprawy trafiały ostatecznie do rozpoznania przez prokuraturę, bo państwo na łeb, na szyję prywatyzowaliście PKS-y, ponieważ wszystko, co prywatne, miało być lepsze.

Pani Poseł Masłowska!

A teraz o ultimatum. Szanowni państwo, ten czas to ultimatum ministra dla wszystkich Polaków. Po pierwsze, dla samorządów.

Co państwo za to proponujecie? Niski fundusz dopłat do transportu publicznego, niską subwencję, małe kontrakty na szpitale - wszystko zawieszacie na samorządzie. Dlaczego? Jeszcze jedna sprawa lokalna. Kolega z Poznania o tym mówił, ja również. Kiedy otrzymamy poprawiony, aneksowany program dworcowy? Mówię o dworcu w Mielcu. Pan jest z Podkarpacia. Myślę, że panu ta sprawa będzie równie bliska. Dziękuję bardzo. Pani poseł Magdalena Biejat, klub parlamentarny Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Rząd mówi dużo o godności i o jakości życia. Chciałabym powiedzieć, że godność i jakość życia jest np. wtedy, kiedy seniorka może samodzielnie pojechać do przychodni i nie czekać pół dnia pod gabinetem lekarskim, bo połączenie w tamtą stronę jest teraz o świcie. Godność jest wtedy, kiedy dziecko może wrócić do domu ze szkoły, nie czekając 3 godziny na ten jedyny autobus, który tam jedzie. Godność jest też wtedy, kiedy można po prostu pojechać do kina do dużego ośrodka niezależnie od tego, w jakim się jest wieku i jaką ma się zasobność portfela. Dziś procedujemy nad ustawą o transporcie zbiorowym, która niczego nie naprawia. Dużo słyszeliśmy wcześniej o inwestycjach w infrastrukturę kolejową. Nie wiemy niestety nic o pomysłach na to, w jaki sposób poprawić jakość i częstotliwość połączeń realizowanych w ramach transportu publicznego, czy to kolejowego, czy autobusowego. Chciałabym wzmocnić głos posłanki Matysiak i posła Sterczewskiego, stąd moje pytania. Czy ewentualne plany uwzględniają zwiększenie liczby i częstotliwości połączeń?

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Z wielkim szacunkiem odnoszę się do samorządów, przedsiębiorców-przewoźników i innych przedsiębiorców, jak również do wszystkich osób korzystających z transportu zbiorowego. Czy państwo, gwarantując środki, które znajdują się w budżecie, na dofinansowanie ulg dla osób dojeżdżających, liczą się z ryzykiem, że w momencie, kiedy nie zdążymy przeprocedować tej ustawy, tego czwartego przesunięcia.

Jakie jest realne zapotrzebowanie ze strony samorządów na dofinansowanie, jeżeli chodzi o ulgi dla osób dojeżdżających np. do pracy? Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Marszałek! Panowie Posłowie! Bardzo dziękuję za dyskusję. Podzieliłbym ją na dwie części: dyskusję, która jest związana stricte z projektem i z naszą ważną i, przyznaję, pilną i szybką propozycją, która polega na tym, aby nadal rekompensować ulgi w przewozach autobusowych, w przewozach komunikacji zbiorowej.

Projekt trafi do Senatu. W przyszłym tygodniu jest dwudniowe posiedzenie Senatu. Jeżeli tam również nie będzie do samego projektu żadnych uwag, to pan prezydent będzie miał kilkanaście dni na to, żeby go podpisać.

Tutaj też jest zgoda. Ten fakt został stwierdzony przez wszystkie kluby parlamentarne. Pytanie jest inne. Jak poprzednie rządy - wszystkich opcji politycznych - walczyły z wykluczeniem komunikacyjnym?

Nie słyszałem tutaj takich głosów, nie słyszałem o tych działaniach, które były przez państwa formacje polityczne w ciągu ostatnich 30 lat podejmowane, bo tak naprawdę żadnych realnych kroków w tej sprawie nie było.

Natomiast do 2030 r. chcemy zakończyć główną bazę, główną sieć dróg szybkiego ruchu w standardzie drogi ekspresowej. W tej chwili jesteśmy piątym krajem Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o długość sieci dróg szybkiego ruchu, ponad 4 tys. km. Kolejny 1 tys. jest w fazie realizacji - albo projektowania, albo już w fazie budowania, i kolejny blisko 1 tys. jest w fazie przygotowywania dokumentacji. 2030 r. to jest ten czas, kiedy Polska będzie objęta blisko 6 tys. dróg szybkiego ruchu. To jest przede wszystkim również dbałość o bezpieczeństwo. I chociaż nasze drogi, polskie drogi są nadal niebezpieczne, nadal na nich dochodzi do zbyt dużej liczby wypadków, to trzeba jednoznacznie stwierdzić, że liczba wypadków z roku na rok spada, że liczba wypadków z roku na rok maleje. Po drugie, Fundusz Dróg Samorządowych, czyli to historycznie wysokie narzędzie wspierania inwestycji drogowych, gminnych i powiatowych.

A w perspektywie 10 lat, między 2019 r. a 2028 r., to 36 mld zł środków rządowych na to, aby wspierać modernizację, przebudowę, ale też budowę nowych ciągów komunikacyjnych na poziomie gmin i powiatów. To jest to narzędzie, które zostało w poprzednim roku stworzone przez rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego.

Przypominam, z jakim problemem się mierzymy. Raport Najwyższej Izby Kontroli z 2015 r. wskazał, że 32% dróg gminnych i powiatowych w Polsce jest w stanie niezadowalającym, a 36% jest w stanie złym.

Chcemy to w dosyć szybkim tempie zmienić, dlatego jest bardzo konkretne i wymierne wsparcie dla samorządowców w tym zakresie. Po trzecie, fundusz rozwoju przewozów autobusowych, kolejne nowe narzędzie stworzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Narzędzie, które funkcjonuje od września br., czyli nieco ponad 3 miesiące. To blisko 1500 linii autobusowych, które zostały na podstawie tego funduszu albo odtworzone, albo powołane od nowa. Wniosków z samorządów jest już więcej, to 256 wniosków w skali całego kraju, ponad 1711 linii autobusowych, które zostaną objęte tym wsparciem finansowym. Tak że jest to jaskrawy i dobitny dowód, że dopiero rozpoczęliśmy walkę z wykluczeniem komunikacyjnym, i będzie to proces, który będzie trwał lata.

Dlaczego we współpracy z samorządowcami? Bo uważamy, że samorządowcy wiedzą lepiej, niż my tutaj w Warszawie, jakie linie należy odtwarzać, jakie połączenia należy finansować. Wiem, że wielu z nich, wielu z samorządowców wykorzystuje do tego również organizacje społeczne, grupy osób, które o to wnioskują. My przekazujemy środki finansowe, maksymalnie 1 zł do wozokilometra, i oczywiście zapewniliśmy podstawę prawną, która temu służy. Tutaj współpraca między rządem a samorządem jest konieczna i wskazana. Część z państwa uważa, że wysługujemy się samorządem, a druga część, że nie dostrzegamy samorządów. Dajemy możliwości, dajemy podstawę prawną, dajemy środki finansowe, ale z drugiej strony oczekujemy aktywności i rozeznania potrzeb społecznych, jeżeli chodzi o odtwarzanie połączeń autobusowych.

Środki finansowe są, podstawa prawna jest, wystarczy zaangażowanie samorządów. Oczywiście są też problemy, których nie rozwiążemy w sposób szybki. Brakuje kierowców autobusów, firmy przewozowe borykają się z tym problemem.

Mam nadzieję, że w tej drugiej sytuacji również stworzymy program, który pozwoli na pozyskanie środków finansowych dla tych przewoźników, którzy będą chcieli postawić na nowoczesny, bardziej ekologiczny i mniej kosztochłonny tabor autobusowy. Ale to też kolejne działanie, które, mam nadzieję, w niedalekiej przyszłości rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie realizował. Jeżeli chodzi o kolej, to program modernizacji kolei również postępuje. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to 70 mld zł na modernizację sieci kolejowej, sprawienie, aby polska kolej jeździła szybciej, aby zwiększała się prędkość przepustowa na liniach kolejowych. Za tę działkę odpowiada bezpośrednio pan minister Andrzej Bittel, on na ten temat mógłby coś więcej powiedzieć.

Szanowni Państwo! Dziękuję za te głosy, które tutaj padły i były głosami bardzo poważnymi, nie skupiały się na ataku na rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale faktycznie pokazywały problemy, z którymi Polska boryka się w ostatnich dekadach, podkreślam to słowo, jeżeli chodzi o komunikację zbiorową, transport zbiorowy. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami w tej kadencji wprowadzimy kolejne narzędzia i kolejne rozwiązania i prawne, i finansowe, aby tę kwestię usprawniać.

Została w połowie tego roku skierowana do prac komitetu stałego Rady Ministrów, ale z racji dyskontynuacji - mieliśmy przecież wybory - prace nad tą ustawą zostały wstrzymane. Jestem przekonany, że w roku 2020 tak się stanie. Bardzo państwu dziękuję za dyskusję.

Dziękuję bardzo, panie ministrze. W takim razie zamykam dyskusję. Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 8. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (druki nr 56 i 60) Proszę pana posła Zdzisława Sipierę o przedstawienie sprawozdania komisji. Bardzo proszę, panie pośle.

W dniu dzisiejszym odbyła się praca związana z pilną ustawą zgłoszoną przez premiera, przez rząd, dotyczącą zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019. Dotyka ona kilku bardzo istotnych punktów dotyczących finansowania bardzo istotnych sfer życia publicznego.

W trakcie pracy komisji i analizy punktów zgłoszonych w ramach propozycji rządu nie było specjalnych sporów co do zasadności propozycji, natomiast chodziło o pewną szczegółowość. Oczywiście tutaj zawsze jest element wyboru, jak szczegółowo trzeba dane informacje przedstawiać, i jest kwestia odpowiedzi odpowiednich przedstawicieli rządu: czy Ministerstwa Zdrowia, czy Ministerstwa Finansów, czy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jedynie była zgoda na poprawki legislacyjne, które zostały wprowadzone, i ten nowy druk jest z tymi zmianami, które już wypełniają całość zakresu zmian ustawowych. I to, pani marszałek, jest wszystko, jeżeli chodzi o sprawozdanie. Dziękuję bardzo, panie pośle. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Otwieram dyskusję. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość stanowisko zaprezentuje pani poseł Gabriela Masłowska. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Projekt ustawy o zmianie ustawy o rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 po przeprowadzeniu pierwszego czytania został skierowany do Komisji Finansów Publicznych. W dyskusji ponawiano pytania, które padały podczas pierwszego czytania, mimo wyczerpujących odpowiedzi ministra finansów, ministra zdrowia i przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w czasie pierwszego czytania na sali posiedzeń.

Takie propozycje nie padły.

Nie pomagają wyjaśnienia, że pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia nie mogą służyć oddłużaniu szpitali, bo to nie jest zadanie Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie pomagają wyjaśnienia, że w 2017 r. o 1 mld zł zwiększono środki dla NFZ-u na spłatę nadwykonań, których rząd PO-PSL nie uregulował wobec szpitali.

Teraz słyszymy, że to już jest tak naprawdę nieważne. Otóż były także zarzuty, że zmiany w planie finansowym nie będą opiniowane przez komisję finansów czy poza parlamentem, co oczywiście także jest nieprawdą, bo są one opiniowane przez Komisję Finansów Publicznych i Komisję Zdrowia oraz w tym drugim wypadku, jeśli chodzi o Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przez odpowiednią komisję.

Dziękuję bardzo, pani poseł. W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska głos zabierze pani poseł Izabela Leszczyna. Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Rozumiem, że pani poseł, która reprezentuje klub PiS-u, może mówić z tej mównicy wszystko, co chce powiedzieć. Tak to zwykle bywa. Może mówić o zadłużeniu szpitali, chociaż wszyscy wiemy, że lawinowo narasta teraz i nie ma porównania w ogóle z zadłużeniem z tych naszych 8 lat. Ale to, że pan poseł Sipiera, sprawozdawca, wychodzi i mówi rzeczy, które się nie wydarzyły, znaczy, że nie rozumie, na czym polega sprawozdanie komisji.

Powtórzę jeszcze raz: w tej ustawie nie chodzi o żadne pieniądze ani dla pana, panie ministrze zdrowia, ani dla pana, panie ministrze Wąsik, na tę Policję. Jeszcze nie wiadomo, czy w ogóle je dostaniecie. W tej ustawie chodzi o jedną rzecz: PiS nie może już wydać ani złotówki z budżetu, bo przekroczył o wiele miliardów limit, jaki narzuca na niego ustawa o finansach publicznych poprzez regułę. Już musieliście wprowadzić Fundusz Solidarnościowy, wyprowadzić 9 mld, wcześniej 4 mld. W tej ustawie musicie wyprowadzić z wydatków budżetowych 3 mld, bo inaczej rząd popełniłby przestępstwo. Nie o szczegółowości planu finansowego. Wyjmujecie bezpieczniki finansów publicznych. Demontujecie regułę, którą przecież rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u wprowadził po to właśnie, żeby rząd nie wydawał więcej pieniędzy, niż to jest bezpieczne dla obywateli. Polska, powtórzę wam to, nie trwa jedną ani dwie kadencje. Polska ma trwać przez lata. Nie możecie zostawić obywateli z wyssanymi do granic niemożliwości finansami publicznymi w czasie, kiedy na całym świecie jest lato w gospodarce. 14 państw Unii Europejskiej w zeszłym roku miało nadwyżkę budżetową, a większość państw Unii Europejskiej miała zrównoważony budżet. Tym bardziej wy. A wy chodzicie od kilku tygodni czy nawet miesięcy, opowiadacie jakieś bzdury o zrównoważonym budżecie, a budżetu na 2020 r. nie ma w ogóle. Nie ma budżetu, bo szukacie 5 mld zł i nie wiecie już, komu by dołożyć jaki podatek, żeby te 5 mld do budżetu jakoś wprowadzić, albo komu zabrać, bo już nie bardzo jest z czego. Taki macie zrównoważony budżet. Mimo że chcieliście go zrównoważyć jednorazowymi dochodami, wprowadzając wieloletnie, stałe, sztywne wydatki. Taki miał być ten wasz zrównoważony budżet, a nawet i to wam nie wyszło. Jeśli minister zdrowia wczoraj wieczorem nie wiedział, że dostanie 2 mld zł, to co to znaczy? To znaczy, że minister finansów wysłał do resortów pismo: Nie wydawajcie, bo już nie wolno, bo staniemy wszyscy przed Trybunałem Stanu. I wszyscy ministrowie w resortach teraz tną wydatki. Na początku roku przychodzi premier Morawiecki i mówi, że jest świetny budżet - inwestycyjny, mamy mnóstwo pieniędzy na inwestycje. Na koniec roku przychodzi i mówi tak: Świetny budżet. Deficyt jest mniejszy, niż miał być. Dlaczego? No bośmy nie zrobili 80% inwestycji, więc nie musieliśmy wydać środków. Takie jest wasze zarządzanie finansami publicznymi. W czasie kiedy koniunktura na świecie się kręci, kiedy dochody podatkowe są wysokie, bo ludzie pracują, bo firmy się rozwijają, bo jest wysoka konsumpcja, także poprzez 500+, wyssaliście ten budżet do granic niemożliwości. Nie zostawiliście kompletnie nic na chude lata. A przecież cykl koniunkturalny, panie ministrze, jest zjawiskiem, i nikt nie powie, że tym razem będzie inaczej. Dziękuję bardzo, pani poseł. Pan poseł Krzysztof Paszyk w imieniu klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego - Kukiz15. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Otóż trudno nie odnieść wrażenia, że mamy do czynienia z serialem pt. dobra koniunktura budżetowa czy zrównoważony budżet. Większość sejmowa niestety nam ten serial funduje od kilku ładnych tygodni. Bo jak to inaczej nazwać? Zbliżał się czas kampanii wyborczej - budżet był zrównoważony, było wszystko w porządku. Po wyborach budżet już nie był zrównoważony, bo cóż przyniosło poprzednie posiedzenie Sejmu? Ano trzy podejścia do pozyskania dodatkowych środków budżetowych. Dwa udane, a jedno za sprawą pana premiera Gowina - nieudane. Idą święta, więc paru grupom zawodowym przydałoby się coś dać pod choinkę. Paru posłów, paru ministrów wysłać, przekazać coś dobrego na koniec roku. To nie jest odpowiedzialna polityka fiskalna, odpowiedzialna polityka budżetowa państwa, panie i panowie ministrowie, Wysoka Izbo. I to jest pierwsze spostrzeżenie, co dzisiaj przy okazji debaty nad tą pilną ustawą zmieniającą budżet trzeba sobie na tej sali powiedzieć. My byśmy, jako Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe wspólnie z Kukiz15, życzyli sobie przewidywalnej polityki budżetowej.

Jak złożyliśmy poprawkę, żeby to poszło na jakiś konkretny cel, bo bardzo ogólnie można powiedzieć, że będziemy poprawiać zdrowie Polaków, ale jak powiedzieliśmy: „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, to pan minister Szumowski wyszedł i mówi: Nie chcę tych 2 mld zł, nie są mi potrzebne.

Wtedy pan minister nie chciał, ale chyba po 2 tygodniach znowu chce. Bo teraz znowu mamy 2 mld zł na stole, które mają wesprzeć fundusz zapasowy w Narodowym Funduszu Zdrowia. Mój klub. Chcielibyśmy być konsekwentni, panowie ministrowie, więc ponawiamy dzisiaj naszą poprawkę do tej ustawy, propozycję, żeby te 2 mld zł, które dzisiaj pojawiają się rzekomo na wsparcie systemu opieki zdrowotnej. Panie ministrze, nie wiem, czy pan wie. Ale wspomniany przez nas właśnie „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, który państwo stworzyliście, państwo, wydaje się, stworzyliście ten program. One cokolwiek w ramach tego funduszu znaczą i dlatego pozwolę sobie złożyć poprawkę do procedowanej ustawy, aby właśnie te 2 mld zł, o których się mówi bardzo ogólnikowo i które najpewniej zginą w morzu potrzeb w polityce zdrowotnej, przeznaczyć na konkretny cel. Mamy problem ze sprostaniem temu zjawisku. Myślę, że Narodowy Fundusz Zwalczania Chorób Nowotworowych wsparty taką kwotą będzie w stanie podejmować kolejne inicjatywy, które będą hamowały plagę chorób nowotworowych, które są coraz bardziej dotkliwe.

Uprzejmie informuję, że do pytań zapisały się cztery osoby. Jako pierwszy pytanie zada pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Pani poseł Urszula Nowogórska, klub PSL - Kukiz15. Bardzo proszę.

Wysoka Izbo! Na tej dziedzinie życia nie można oszczędzać, choć jest to dziedzina bardzo wymagająca finansowo i w zasadzie wykorzystująca każde środki finansowe, które pojawiają się w danym momencie do wykorzystania. Rozumiem również, że jest to pewna forma docenienia tych ludzi, którzy realizują swoją pracę nie tylko w godzinach pracy, ale również po niej, i niejednokrotnie realizują swoją pracę również jako misję. Zważywszy na racjonalność wydatków, mam nadzieję, że te środki, które pojawiają się teraz w budżecie, w sposób nagły i nieprzewidywalny, zostaną wydatkowane racjonalnie, mądrze i nie byle jak.

Dziękuję. Dziękuję, pani poseł. Bardzo proszę.

Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chodzi tu o bardzo ważne cele, bo trzeba doposażać wszystkie służby, trzeba tych pieniędzy szukać, ale też trzeba po prostu wolniej jeździć, tak jak wszyscy jeżdżą. Nie ma miesiąca, żebyśmy się nie dowiadywali o jakiejś kolejnej kolizji, rozbiciu kolejnych aut, zarówno tych Służby Ochrony Państwa, jak i policyjnych.

Dziękuję bardzo.

Mam pytanie, panie ministrze: Czy tego typu praktyka jest dozwolona? Czy nie jest ona sprzeczna z ustawą o podatku akcyzowym?

Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Bardzo proszę. Wysoki Sejmie! Trzy krótkie odpowiedzi. Po raz kolejny pojawia się twierdzenie, że rząd, że minister finansów przekroczył limit określony regułą wydatkową. Otóż nie przekroczył, a gdyby przekroczył, to oczywiście byłoby to złamanie ustawy budżetowej i złamanie prawa. Nie jest tak, że nie można już wydać ani złotówki z budżetu, ponieważ cały czas wydatki budżetowe są realizowane i będą realizowane aż do końca grudnia, tak jak co roku.

Aczkolwiek są to oczywiście wydatki, tak jak mówiłem, potencjalne.

Tą ustawą, w przypadku gdy będą oszczędności w budżecie, będzie można przekierować środki jeszcze tegoroczne na cele, które są wskazane w ustawie. Ostatnia kwestia to sprawa przeznaczenia środków z podatków na konkretne cele.

Czy ktoś jeszcze w imieniu rządu? Dziękuję. Czy sprawozdawca komisji pan poseł Zdzisław Sipiera będzie chciał odnieść się do zadanych pytań? Wysoki Sejmie! Pan minister też już odpowiedział. Podczas procedowania nad tak istotną zmianą - bo to są konkretne pieniądze w funduszu, ale również przesunięcia środków do wydatkowania w okresie do kwietnia - nie było chyba sporu. Zgadzamy się, żeby te fundusze były wydatkowane.

Jeżeli rząd proponuje 2 mld zł na świadczenia zdrowotne, to jest to chyba dobry kierunek działania i powinien on być absolutnie poparty przez wszystkich bez żadnej dyskusji.

To oczywiście jest dociekliwość już samych posłów, ona może istnieć, ale tylko i wyłącznie odpowiedź co do tych szczegółowych zapisów będzie, mam nadzieję, udzielana przez rząd. To już było powiedziane przez panią poseł Masłowską i pana ministra. Natomiast budżetowanie ma to do siebie, że jest strona przychodów, dochodów i strona wydatkowa. Dziękuję bardzo, panie pośle. Zgłosił się również pan minister Maciej Wąsik, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, z chęcią odpowiedzi na pytania.

Pierwsze zadanie to pokrywanie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymywania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług. Drugie zadanie to rekompensata pieniężna dla policjantów za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie. Trzecie - nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm skierował ponownie ten projekt do Komisji Finansów Publicznych w celu przedstawienia sprawozdania. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Zarządzam przerwę do godz. 18, kiedy to przystąpimy do bloku głosowań. Dziękuję.

Proszę państwa, wznawiam obrady. Do protokołu 1. posiedzenia Sejmu przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zgodnie z art. 176 ust. 5 regulaminu Sejmu o przyjęciu lub odrzuceniu poprawki Sejm rozstrzyga większością głosów bez dyskusji. W poprawce wnioskodawca proponuje uzupełnienie protokołu 1. posiedzenia w punkcie 20. porządku dziennego, dotyczącym wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, o słowa wypowiedziane przez zastępcę szefa Kancelarii Sejmu, skierowane do marszałek Sejmu i odnoszące się do procedury głosowania. Zgłoszona poprawka została przedstawiona i omówiona na posiedzeniach Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów w dniu dzisiejszym. Przystępujemy do głosowania.

Bardzo proszę.

Proszę państwa, chwila.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki do protokołu 1. posiedzenia Sejmu, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz Prawo celne. Sejm podjął decyzję o niezwłocznym przystąpieniu do drugiego czytania projektu ustawy. Przystępujemy zatem do trzeciego czytania. W pierwszej kolejności poddam pod głosowanie poprawkę, a następnie całość projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę przyjął. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz Prawo celne, zawartego w druku nr 51, wraz z przyjętą poprawką, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 430 było za, nikt nie był przeciw, 1 poseł wstrzymał się od głosu. Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy Prawo celne. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. W dyskusji zgłoszono wnioski: o przystąpienie niezwłocznie do drugiego czytania projektu ustawy oraz o skierowanie projektu ustawy do Komisji Finansów Publicznych. Pod głosowanie poddam wniosek o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania projektu ustawy. Odrzucenie tego wniosku oznaczać będzie, że Sejm skierował ten projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania projektu ustawy z druku nr 40, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos w drugim czytaniu projektu ustawy? 1 minuta, pani poseł. 3 minuty, pani poseł? Panie i Panowie Posłowie! Drożyzna życia nie tylko w sklepach stanie się symbolem waszego rządu.

Będą go płacić docelowo konsumenci. Nie żadna instytucja handlowa, nie żaden międzynarodowy koncern, tylko Polacy, kupując każdego dnia, robiąc zakupy w sklepach. To nie jest jedyny problem. Drożyzna będzie nam doskwierać przez całe kolejne 12 miesięcy.

Czeka nas podwyżka cen paliwa, bo rząd podnosi opłatę paliwową.

Czeka nas podwyżka za wywóz nieczystości w związku z zaostrzeniem warunków segregacji odpadów i utylizacji śmieci. Czeka nas też wzrost różnych podatków w samorządach, bo rząd zabrał dochody samorządom, a nie zabrał im zadań. W związku z tym będą rosły lokalne podatki, bo samorządy muszą jakoś sobie poradzić z zadaniami, które rząd na nie nakłada. To wszystko sprawi, że życie Polaków będzie po prostu w przyszłym roku droższe.

Chcieliśmy o tym wszystkim rozmawiać w Komisji Finansów Publicznych, ale wy nie macie odwagi. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana.

Dobrze, dziękuję. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 40, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 55-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę pana posła Zbigniewa Babalskiego o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych przedstawiam dodatkowe sprawozdanie o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, druki nr 42 i 55. Wysoki Sejmie!

Komisja nie rozpatrywała wniosku o odrzucenie projektu uchwały w całości ze względu na opinię Biura Legislacyjnego mówiącą, że wniosek został złożony niezgodnie z regulaminem.

Komisja wnosi o uchwalenie projektu uchwały z druku nr 55. Komisja przedstawia również w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności.

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Pani marszałek, nie usłyszałem. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zmieniamy regulamin Sejmu, żeby mieć procedurę, jak wybierać siedmiu spośród dziewięciu członków Państwowej Komisji Wyborczej. Wszystkie te przepisy mówią, jak dojść do momentu, kiedy tych siedmiu Prezydium Sejmu przedstawi do głosowania. I oto w ust. 8, kiedy już Prezydium Sejmu przedstawia siedmiu kandydatów, którzy mają być wskazani, mówimy o tym, że wskazanie członków Państwowej Komisji Wyborczej odbywa się łącznie, czyli mamy tutaj taki projekt, że będziemy w Sejmie razem, proporcjonalnie, w ramach porozumienia, konsensusu ustalać, co to będzie za siedem osób. Następnie jednak w propozycji dodaliście: chyba że Sejm postanowi inaczej. A my z praktyki poprzedniej kadencji wiemy, co to znaczy: chyba że Sejm postanowi inaczej.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

Wysoka Izbo! Właśnie nie zdaliście egzaminu na wiarygodność. Nie można wam wierzyć, że macie jakiekolwiek dobre zamiary w zakresie wybierania członków Państwowej Komisji Wyborczej w kolejnej poprawce, bo wprowadzacie zasadę, że można członka Państwowej Komisji Wyborczej odwołać. A wy wpisujecie, że z byle powodu można odwołać członka Państwowej Komisji Wyborczej, że Sejm może wnioskować o jego odwołanie. Sejm, który jest najbardziej zainteresowany tym, kto zasiada w Państwowej Komisji Wyborczej. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Rozumiem, że ta część sali boi się takich przypadków, jak Marian Banaś, którego nie możecie odwołać, mimo że kompromituje swój urząd zarzutami, które są powszechnie formułowane. My proponowaliśmy w poprawce, o której mówił pan poseł Urbaniak, żeby nie można było z byle powodu odwołać członka Państwowej Komisji Wyborczej. Chcemy, żeby takie odwołanie mogło nastąpić wtedy, kiedy zostanie on prawomocnie skazany za przestępstwo przeciw wyborom i referendom, za nadużycia przy przebiegu wyborów, za zakłócenie przebiegu wyborów, za bezprawne wywieranie wpływu, za łapownictwo wyborcze czy też naruszenie tajności głosowania. Chodzi o to, żeby nie było tak, że członkowie PKW będą w pełni podporządkowani większości parlamentarnej i kiedy będziecie mieć takie życzenie, będziecie mogli tę osobę z dnia na dzień odwołać, wnioskując o to do prezydenta. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przystępujemy do głosowania nad całością projektu uchwały.

Wysoka Izbo! Ta zmiana regulaminu to implementacja zmian Kodeksu wyborczego z 2018 r. Do tej pory członków Państwowej Komisji Wyborczej wskazywał Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny. To był tzw. model sądowy. Mieliśmy gwarancję niezawisłości i niezależności członków Państwowej Komisji Wyborczej. Wy to zmieniacie.

To nie tylko złamanie konstytucji, art. 2 mówiącego o tym, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawa. To jest złamanie jednej z podstawowych zasad funkcjonowania cywilizacji europejskiej, cywilizacji łacińskiej: nie wolno być sędzią we własnej sprawie. Naprawdę, nie idźcie na wschód. Tam nie ma żadnej cywilizacji. Dziękuję, panie pośle. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu uchwały. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu uchwały w brzmieniu z druku nr 55, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Powracamy do rozpatrzenia punktu 6. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 54-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę pana posła Henryka Kowalczyka o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! W czasie drugiego czytania zgłoszono 13 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, tzw. ustawy mały ZUS. Wszystkie poprawki komisja rozpatrzyła i zaopiniowała negatywnie. Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 54. Komisje przedstawiają w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi Sejm głosować będzie w pierwszej kolejności. Poprawki od 1. do 12. zostały zgłoszone do art. 1 projektu ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Nad nimi głosować będziemy łącznie. Komisje wnoszą o ich odrzucenie. 1 minuta, panie pośle. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Rząd PiS wielokrotnie mówił o wspieraniu ludzi młodych, o tworzeniu odpowiednich szans do rozwoju, do pracy, do tworzenia własnego biznesu. Proszę was o poparcie poprawki, naszej poprawki, dzięki której młodzi przedsiębiorcy, do 25. roku życia, zostaną zwolnieni z konieczności płacenia składek na ZUS i NFZ. Dzięki temu ktoś, kto rozpoczyna studia, przez 5 lat - według obecnych przepisów - nie będzie musiał oddać do kasy państwa prawie 50 tys. zł, a te pieniądze będzie mógł wykorzystać na rozwój własnej działalności. Uzasadnię to jeszcze tym, że w tej grupie - młodych do 25 lat - tylko 35 osób na 100 jest aktywnych zawodowo. Jeśli więc większość z nich dziś nie płaci podatków, jeśli będzie zwolniona w przyszłości z płacenia podatku, a będzie aktywna, to będzie to tylko coś pozytywnego dla naszej gospodarki i coś pozytywnego dla młodych, którzy będą mogli swoje innowacyjne, nowoczesne pomysły wdrażać w życie i nie martwić się o to, czy starczy im na opłacenie składek na ZUS. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 1. i 2., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Sejm poprawki odrzucił. Komisje wnoszą o jej odrzucenie. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mały ZUS+ miał być wielkim zbawieniem dla przedsiębiorców. 75% przedsiębiorców nie będzie miało niższego ZUS-u, ale od przyszłego roku zapłaci składkę na ZUS i NFZ - prawie 1500 zł. Proponujemy w naszej poprawce, aby podstawą do naliczenia składek na ZUS była płaca minimalna. Czyli w przyszłym roku 2600, a nie ponad 3200, czyli 60% średniego wynagrodzenia. Dzięki temu w przyszłym roku przedsiębiorcy bez względu na to, jaki mają dochód, jaki przychód, czy są dużymi przedsiębiorcami, czy nie, zapłacą prawie 200 zł mniej składek na ZUS i NFZ. I to jest prawdziwa pomoc dla przedsiębiorców. To jest wyjście naprzeciw ich oczekiwaniom. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił. Nad nimi głosować będziemy łącznie. Ich przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość poprawek od 5. do 11. Bardzo proszę, pani poseł. Wysoka Izbo!

To poprawka, która znosi limit 120 tys. przychodu.

I ta poprawka pozwala jej również skorzystać z tej ulgi. Ponieważ dochód to jest to, co ludzie otrzymują ze swojej pracy, a nie przychód. Wyklucza się tych, którzy coś produkują, i wyklucza się, co najgorsze, polski, mały handel, który już wielokrotnie dostał za swoje i nigdy nie był wspierany ani przez Polskę, ani przez Unię Europejską. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 4. i 12., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Stwierdzam, że Sejm poprawki odrzucił. Nad nimi głosować będziemy łącznie. Komisje wnoszą o ich odrzucenie. Ich przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość poprawek od 6. do 8. oraz 10.

Wysoka Izbo! Ryczałtowy ZUS to seryjny morderca polskiej przedsiębiorczości. Ojeju... Państwo, wprowadzając tę ustawę, chcą ulżyć przedsiębiorcom, ale kryterium przychodowe to jedna z największych dyskryminacji, jakie widziała ta Izba. Czym się różni krawcowa, której nie stać na zapłacenie horrendalnego ZUS-u, od właścicielki warzywniaka, której dochód jest nawet często mniejszy niż krawcowej? Niczym. Państwa kryterium przychodu nie ma nic wspólnego z tym, czy przedsiębiorcę stać na zapłacenie tego ZUS-u, ile ten przedsiębiorca zarabia. Kryterium przychodowe determinuje tylko branżę, w jakiej przedsiębiorca działa: czy to jest branża usługowa, czy to jest branża handlowa, czy to jest branża produkcyjna. W związku z tym, żeby być uczciwym wobec wszystkich małych przedsiębiorców, których dobija ten horrendalny ZUS, proponujemy, by zlikwidować (Dzwonek) kryterium przychodowe. Bardzo proszę. Panie i Panowie Posłowie! Miał być system powszechny, a wyszedł tak naprawdę system wykluczający zarówno krawcowe, jak i małe sklepy. Ale moje pytanie będzie skierowane w inną stronę. Czy rząd zamierza przeprowadzić dobrą, solidną kampanię informacyjną, która uświadomi przedsiębiorców w sprawie negatywnych kwestii związanych z tą ustawą?

Czy uświadomicie przedsiębiorców, że po korzystaniu z małego ZUS-u nie będą mieli prawa do zasiłku dla bezrobotnych?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 5., 9. i 11., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Stwierdzam, że Sejm poprawki odrzucił.

Bardzo proszę. Panie Ministrze! Szanowni Państwo! Rząd obiecał przedsiębiorcom, zwłaszcza małym i średnim, że ulży ich doli w sytuacji, kiedy zbliża się spowolnienie gospodarcze i kiedy obciążenia na rzecz ZUS należą do najbardziej dotkliwych finansowych danin. Niestety propozycja rządu, która dotarła do tej Izby, jest głęboko rozczarowująca. Mam pytanie do pana ministra i do pana premiera, który składał tak daleko idące obietnice: Dlaczego jesteście tak mało ambitni?

Oznaczałoby to, przy zachowaniu dyscypliny finansowej, że znacznie (Dzwonek) większa liczba przedsiębiorstw będzie objęta działaniem tej ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 6., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił. Komisje wnoszą o ich odrzucenie. Bardzo proszę, panie pośle. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przed chwilą politycy Prawa i Sprawiedliwości pokazali, jak traktują przedsiębiorców. Dlatego mamy dla państwa systemowe rozwiązanie. Zamiast 120 tys. zł proponujemy, aby wpisać krotność - krotność najniższego wynagrodzenia. Określamy ją na poziomie 45. To powoduje, że od przyszłego roku będzie to kwota 117 tys. zł, ale przecież poseł Kaczyński mówił, że już za 3 lata najniższe wynagrodzenie będzie wynosiło 4 tys. zł, więc według naszej propozycji za 4 lata ta kwota będzie wynosiła 180 tys. zł. Jeżeli państwo macie chęć i ambicję, aby przedsiębiorcom żyło się lepiej i aby ten mały ZUS+ rozszerzał się każdego roku, to to jest właśnie ta droga i ta propozycja. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 7., 8. i 10., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Sejm poprawki odrzucił. W 13. poprawce wnioskodawcy proponują skreślić art. 3 projektu ustawy nowelizującej. Komisje wnoszą o jej odrzucenie. Wysoka Izbo! Ta poprawka znosi czasowość obowiązywania tej ulgi. Skoro państwo w uzasadnieniu podajecie, że ta ulga jest dla drobnych krawcowych, szewców czy drobnych usługodawców, a ten projekt już działa ponad rok, wcześniejszy, to proszę mi powiedzieć: Czy macie państwo takie dane, że przez ten rok ten szewc, ta krawcowa stali się nagle potentatami obuwniczymi, przemysłu odzieżowego, czy rzeczywiście ich sytuacja się zmieniła? Jeżeli nie, to dlaczego to ma obowiązywać czasowo? Dlaczego takim właśnie przedsiębiorcom, do których adresujecie tę minimalną pomoc, chcecie nagle po 3 latach to urwać? Czy nie jest tak, że większość z nich zdecyduje się po prostu na zamknięcie tej działalności? Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 13. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Ale przed tym pytania. Bardzo proszę. Panie Premierze! Wysoka Izbo! 4 lata temu była zapowiadana szumna, wielka konstytucja dla biznesu. To jest jeden z tych dwóch akapitów. Dobry akapit, nie mówię, że nie, i pewnie ten akapit wszyscy tu na tej sali poprzemy. Ale panie premierze, czy nie lepszym rozwiązaniem, sprawiedliwym, sprawdzonym w innych krajach, opartym na tym, że przedsiębiorcy są ludźmi myślącymi, odpowiedzialnymi, umieją obracać pieniędzmi i dają pieniądze do budżetu, jest projekt, który został złożony przez Koalicję Polską - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15, a popierany przez rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, przez wszystkich przedsiębiorców, projekt dobrowolnego ZUS-u? Czy nie lepiej pozwolić, aby przedsiębiorcy zdecydowali, tak jak każdy pracujący, przez 20 lat, że płacą składki, a następne 20 lat pomnażali pieniądze, które dla was, dla nas i dla wszystkich obywateli będą pracować? Dziękuję, pani poseł. Proszę.

Szanowni Państwo! Zwracam się do posłanek i posłów Prawa i Sprawiedliwości. Po tym głosowaniu pojedziecie do swoich okręgów wyborczych i

Pytanie zadaje pan poseł Jakub Kulesza, Konfederacja. Szanowni Państwo!

No i patrzę na głosowania i jestem trochę zdumiony. Przy poprawce PSL-u klub lewicy - 48 za, przy identycznej poprawce Konfederacji klub lewicy - 43 przeciw. Czy tak wygląda merytoryczna opozycja? Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 54, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 433 było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Powracamy do rozpatrzenia punktu 7. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Przystępujemy do trzeciego czytania. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 44. Bardzo proszę, panie pośle. Wysoka Izbo! Ja tylko chciałem powiedzieć, że ta ustawa, w skrócie, dotyczy bardzo ważnej rzeczy, czyli transportu zbiorowego, a mianowicie systemu ulg do biletów komunikacji podmiejskiej i pozamiejskiej. Ta regulacja powinna wejść już 4 lata temu, miała wejść od 2017 r., niestety co roku jest odraczana, co jest wielkim problemem dla samorządów oraz pasażerów i pasażerek w całej Polsce. Dlatego uważam, że to jest skandal, że transport zbiorowy nie jest traktowany wystarczająco poważnie. Uważam, że powinniśmy od stycznia na poważnie zająć się tym tematem. Dlatego klub Koalicji Obywatelskiej wstrzyma się od głosu.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 44, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk, Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Powracamy do rozpatrzenia punktu 8. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 60-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę pana posła Zdzisława Sipierę o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

2 mld zł, które przeznaczone są na sfinansowanie „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”, według wnioskodawców powinno zostać przeznaczone na sfinansowanie innego wydatku, czyli „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”

Natomiast głosowano nad nim dlatego, że był podtrzymany przez wnioskodawców.

Komisja przedstawia w dodatkowym sprawozdaniu poprawkę, nad którą Sejm głosować będzie w pierwszej kolejności. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Bardzo proszę, panie pośle. Wysoka Izbo!

Szanowni Państwo!

Wysoka Izbo, Karczewski jest wolontariuszem dekady.

Bardzo proszę. Wysoka Izbo!

To jest po prostu kpina z tej Izby, to jest kpina z obywateli, naprawdę. Bardzo proszę, żebyście państwo decyzje o przesunięciu w budżecie - a jest to jedna z najważniejszych rzeczy - ok. 3 mld zł, naprawdę. Żebyśmy wszyscy mogli to przemyśleć i poprzeć, tak jak dzisiaj popiera was Lewica. Dziękuję, pani poseł. O głos poprosił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia pan Janusz Cieszyński. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Szanowni państwo, ta poprawka w gruncie rzeczy oznacza, że zabieramy z Narodowego Funduszu Zdrowia 2 mld zł i przeznaczamy je na coś, co jest już sfinansowane z budżetu. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę. Panie Ministrze! Dobrze wiemy, że w tej ustawie wcale nie chodzi o żadne pieniądze na zdrowie. Zresztą poprzednia poprawka dokładnie to pokazała. Dobrze wiemy, że wcale nie chodzi też o żadne pieniądze na Policję. Wyjmujecie dzisiaj bezpieczniki i rozmontowujecie stabilizującą regułę wydatkową, która miała hamować apetyt rządu na wydawanie pieniędzy, których nie posiada, albo pieniędzy odłożonych na czarną godzinę.

Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 60, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 9. porządku dziennego: Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 53) Prezydium Sejmu na podstawie art. 20 ust. 1, art. 137 ust. 4 i art. 148a ust. 12 regulaminu Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, przedłożyło wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos w sprawie przedstawionych propozycji? Nikt się nie zgłasza. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku w brzmieniu z druku nr 53, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 426 posłów. Sejm podjął uchwałę w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie punktów porządku dziennego zaplanowanych na dzień 12 grudnia. Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie jeszcze wygłosić oświadczenie? Listę posłów zgłoszonych do oświadczeń uważam zatem za zamkniętą. Bardzo proszę, pani poseł. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chcę wygłosić oświadczenie dotyczące Muzeum Śląskiego. Wspomnę o historii.

Procedura konkursowa wymagałaby bowiem kilkumiesięcznych działań, a na to nie było czasu, bo termin otwarcia Muzeum Śląskiego nieubłaganie się zbliżał - tak tłumaczył ten fakt ówczesny marszałek sejmiku śląskiego z Platformy Obywatelskiej. W zamierzeniu Muzeum Górnośląskie miało być zlikwidowane. Takie były działania ówczesnych władz sejmiku śląskiego. Moja interwencja, po czterech próbach podejścia ze strony władz ówczesnego urzędu marszałkowskiego, doprowadziła do uratowania tejże placówki. Dowiadujemy się obecnie, że decyzja o odwołaniu pani dyrektor Alicji Knast jest spowodowana motywami politycznymi. Powołanie na stanowiska dyrektorskie bez konkursu i z odpowiednią gażą nie było sprawą polityczną, natomiast obecnie kontrola w katowickiej placówce, która ujawniła liczne nieprawidłowości, a w konsekwencji wszczęcie procedury odwołania dyrektor Alicji Knast, jest sprawą polityczną? Naruszanie ustawy o rachunkowości. Fakt utylizacji całych lub części wystaw bez dokumentów potwierdzających, a były to wystawy o wartości ponad 100 tys. zł, a nawet ponad 900 tys. złotych. Brak dokumentacji wskazującej na podejmowanie działań zmierzających do właściwego zarządzania mieniem placówki. Rozbieżność w kosztach wynajmu pomieszczeń itd., itd. Głośniej! Obecnie urząd marszałkowski twierdzi, że wyniki audytu przeprowadzonego w Muzeum Śląskim są równie porażające dla dyrekcji placówki. Należy podkreślić, że dyrektorzy zarządzają bezcennymi zbiorami, przekraczającymi wyobrażenie przeciętnego Polaka o ich wartości materialnej, i dlatego jeśli są nieprawidłowości, to należy rozliczyć odpowiedzialnych za ten stan rzeczy i wymienić ich na osoby z kompetencjami i odpowiednim wykształceniem, co najmniej z tytułem kustosza muzeum.

Każdy ocalony zabytek to świętość, którą należy chronić bezwzględnie.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

A warto sobie uświadomić, że jest to wydarzenie ważne nie tylko dla polskiej literatury, dla polskiej kultury czy w ogóle dla literatury europejskiej, ale to jest też ważne wydarzenie z punktu widzenia tego właśnie, co przekazuje w swoich książkach Olga Tokarczuk.

Kiedyś Stendhal mówił o tym, że literatura jest jak zwierciadło, które przechadza się gościńcem. Ale warto przypomnieć, że mówił także o tym, że w tym zwierciadle raz po raz przegląda się lazur nieba, a czasami błoto przydrożnej kałuży. I właśnie taki jest dzisiaj świat: pomiędzy lazurem nieba a tą kałużą. Jest rozciągnięty pomiędzy tym, czym chcemy być, kim chcemy być, i tym, kim czasami jesteśmy lub kim czyni nas świat. Olga Tokarczuk w swojej narracji, w swoich powieściach, rozpoczynając od „Podróży ludzi Księgi”, opowiada o nas, opowiada o naszym życiu.

Czasami zazdrościmy tego, kim są bohaterowie, chcemy być tacy, jak oni, chcemy mieć kilka żyć. Bo świat stał się bogatszy dzięki temu, że poznajemy go przez literaturę, poznajemy go przez sztukę. Olga Tokarczuk, warto o tym powiedzieć, jest też w pewnym sensie reprezentantką pokolenia świetnych polskich pisarzy. Bo to jest i Andrzej Stasiuk, to jest Natasza Goerke, to jest Marzanna Kielar, to jest Adam Wiedemann, to jest Krzysztof Siwczyk. To jest całe grono świetnych pisarzy, którzy debiutowali w latach 90. i dzisiaj są chlubą polskiej literatury. Są tłumaczeni na całym świecie. Reprezentują naszą kulturę 100 razy lepiej niż, przepraszam bardzo, minister kultury czy obecni rządzący ze wszystkimi swoimi przyległościami.

Mianowicie, że to zwierciadło, w którym się przegląda gościniec, jest dzisiaj właśnie rozbite. Właśnie ta fragmentaryzacja to jest właśnie to, co się dzisiaj stało z naszym światem także poprzez to, że odkryliśmy wiele nowych rzeczy poprzez technologię. Odkrywamy wiele światów poprzez to, w jaki sposób działa dzisiaj chociażby Internet.

Olga Tokarczuk w swoich powieściach właśnie mówi o tym, jak odnaleźć wspólną historię, wspólną drogę, wspólną narrację. Mówi o tym, że powinniśmy to zrobić przez kategorię czułości. Ale Olga próbuje to także nam opowiedzieć. Tylko trzeba czytać te powieści. Nie zaczynać i porzucać. Trzeba je czytać do końca. Trzeba czytać je mądrze.

Nagrodę tę otrzymała Olga Tokarczuk, ale tak naprawdę myślę, że Olga by się ze mną zgodziła. Zgodziłaby się z tym, że w istocie tę nagrodę noblowską otrzymała polska literatura. Wszyscy ci, którzy w niej tam cierpliwie, rzemieślniczo dłubią, próbują do nas mówić w sposób mądry i taki, w którym poniekąd starają się pomóc nam zrozumieć świat. Dziękuję. Pan poseł Jan Mosiński, klub Prawo i

Nie ma pana posła? Jest, tylko nie słyszy. Pan poseł Jan Mosiński.

Chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę Wysokiej Izby na akcję, która odbyła się kilka dni temu w całej Polsce, a mianowicie organizowanie akcji mikołajkowych dla domów dziecka, dla rodzin, którym w życiu się nie udało, dla rodzin biednych, gdzie skromne budżety nie pozwalały na to, aby zakupić dzieciom upominki.

Tysiącom młodych ludzi, którzy organizowali akcję mikołajkową w skali całego kraju. Były też organizacje, które z działalnością charytatywną nie mają wiele wspólnego, ale również włączyły się w te szlachetne działania. I tak a propos szlachetności, chciałbym zwrócić uwagę na to dzieło, które wykonała Szlachetna Paczka. Otóż w wyniku 19. edycji Szlachetnej Paczki łączna wartość pomocy przekazanej w paczkach dla dzieci, rodzin wyniosła ponad 45 860 tys. zł.

Średnia wartość paczki wyniosła ponad 3400 zł, a średnia liczba osób przygotowujących paczkę to 38. Obok Szlachetnej Paczki mamy też coś takiego, o czym chciałbym wspomnieć, a mianowicie OFF ROAD Team Kalisz. Ludzie, którzy lubią jeździć, lubią skrajne - że tak powiem - warunki uprawiania jazdy samochodami terenowymi, skrzyknęli się w Kaliszu, aby przygotować akcję mikołajkową dla dzieci z Domu Dziecka w Liskowie. Myślę, że nagrodą dla nich były uśmiechnięte buzie tych dzieciaczków, które zobaczyły potężne samochody, o potężnych silnikach, ryczące jednostki, jak niektórzy mówią, którymi to samochodami przyjechali ludzie z OFF ROAD Team Kalisz do tego domu dziecka. Chciałem podziękować - bo to są młodzi ludzie, fascynaci takiej jazdy, to jest bardzo piękny sport - za to, że znaleźli czas, aby u dzieci właśnie w Domu Dziecka w Liskowie wywołać uśmiech na buzi, kiedy zajechali z tymi paczkami.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Wierna do końca ideałom pierwszej „Solidarności”, niezwykle wrażliwa na cierpienie i krzywdę drugiego człowieka. Wzór empatii, bez przerwy uśmiechnięta i otwarta. Swoje sprawy zostawiała na później. Odeszła rok temu, zdecydowanie przedwcześnie, pozostawiając wielu ludzi dobrej woli, przyjaciół, koleżanki i kolegów w wielkim smutku. Odchodziła z godnością, z wielką wiarą i pokorą, przyjmując wolę Pana. Cierpiała w ciszy, nie upominając się o siebie ani o swoje potrzeby. Sejm bez Jolanty Szczypińskiej, bez pani poseł nie jest tym samym Sejmem.

Liczny udział wiernych w Eucharystii świadczył o wielkiej sympatii, jaką cieszyła się pani poseł w Słupsku.

Tablica została wmurowana w ścianę budynku przy ul. Lutosławskiego, w którym przez wiele lat miała biuro poselskie i pracowała jako parlamentarzystka. Po odsłonięciu tablicy uczestnicy uroczystości mieli możliwość uczestniczenia w premierze niezwykłego reportażu o Jolancie Szczypińskiej.

Znowu widzieliśmy Jolę piękną, uśmiechnięta, wspominaną przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, przyjaciół, działaczy „Solidarności”, parlamentarzystów.

Jako prezes zarządu okręgowego okręgu 26 Słupsk, czyli organizatora niedzielnych uroczystości, z tego miejsca składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do uświetnienia uroczystości rocznicowych.

Dziękuję bardzo wicewojewodzie Mariuszowi Łuczykowi, skarbnikowi zarządu okręgowego w Słupsku Jackowi Zabiegłemu za wielkie zaangażowanie i pomoc, byłym pracownikom, pani poseł Agnieszce Błachnio i Jackowi Żukowskiemu za piękną prezentację multimedialną. Podziękowania składam pani prezydent Słupska Krystynie Danileckiej-Wojewódzkiej za wszelką okazaną pomoc organizacyjną i wielkie wsparcie. Chciałbym podziękować pani dyrektor oraz współpracownikom Telewizji Polskiej w Gdańsku, Joannie Jereczek i Rafałowi Ostrowskiemu - autorom dokumentu oraz całemu zespołowi pracowników, dzięki których pracy powstał reportaż „Ja się nie upominam o siebie” Wieczorem do Słupska przyjechała pani marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbieta Witek i złożyła kwiaty na grobie oraz przy tablicy.

Jolu, pamiętamy i będziemy pamiętać o tobie. Pani poseł Joanna Fabisiak, klub Koalicja Obywatelska.

Wysoka Izbo! To dobrze, że podjęto próbę uporządkowania sprawy recept dla wygody pacjentów. Ale czy na pewno dla wygody? Otóż ten proces przechodzenia z recepty papierowej na e-receptę w Wielkiej Brytanii trwał kilka lat, w Polsce będzie trwał kilka miesięcy. Jakie zagrożenia widzą i lekarze, i pacjenci?

Jaki to procent? To dotyczy, powiedzmy, 30%. Pozostałe osoby muszą się do tego przygotować. Ten czas jest za krótki. W tej sprawie już 2 grudnia była interpelacja, której autor skoncentrował się przede wszystkim na tym, że lekarze, a mamy ponad 60% lekarzy starszych, mogą sobie nie poradzić, mogą odchodzić z pracy. Ja się z tym nie zgadzam. Lekarze sobie poradzą. Natomiast czy poradzą sobie pacjenci? Pacjenci, którzy będą dostawali kod, przyzwyczajeni są do recepty. Można nie wiedzieć, można nie mieć. Ale są poważniejsze problemy. Pierwszy to zawodność systemów komputerowych.

Nie dalej jak dzisiaj jeden z lekarzy włączył komputer. I co zobaczył zamiast możliwości wystawienia recepty? A więc nie jest to do końca przygotowane. Moje oświadczenie po tej interpelacji, która na razie nie wywołała żadnego skutku, jest w tym celu, aby ministerstwo jeszcze zmieniło tylko jedną rzecz - bo przecież mamy posiedzenie - wydłużyło vacatio legis przynajmniej o pół roku.

A więc może od razu. Nie warto wprowadzać niepokoju. Dla pacjenta, bo to on nie dostanie recepty. A jeśli w małej miejscowości nie działa czy nie będzie w danym momencie działał Internet, to czym to będzie skutkowało dla pacjenta? Tym, że będzie musiał ponownie przyjść do lekarza i czekać na receptę ileś czasu - a dojechać czasami kilkadziesiąt kilometrów. Tych problemów jest znacznie, znacznie więcej, np. służby ratownicze nie zawsze dysponują laptopem, nie zawsze są do tego przygotowane. Czasami, jak mówili mi lekarze - miejscowości są bardzo małe - ciężko jest dojechać, nie mówiąc o wystawieniu recepty. Jest jeszcze czas, dobry czas, aby z samego założenia bardzo dobrą inicjatywę dobrze przeprowadzić, bez niepokoju pacjentów, bo w nich głównie uderzą wszystkie nieprawidłowości i brak należytego przygotowania.

Nie chodzi o średnią krajową. Chodzi o każdego pacjenta, szczególnie tego starszego, szczególnie tego niepełnosprawnego.

Pani poseł Małgorzata Chmiel, klub Koalicji Obywatelskiej. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Od 1 stycznia 2020 r. obowiązywać będzie nowa ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. W związku z tym władze kolejnych gmin zmuszone są do podnoszenia opłat za wywóz śmieci. Kalkulują to od kilku tygodni.

To kolejna ustawa wprowadzona przez ten rząd, której skutkami obciążane są samorządy, czyli my, mieszkańcy. Gminy chciałyby zmniejszyć te podwyżki, ale bez dotacji z budżetu państwa, choć częściowej, nie będzie to możliwe. Tak drastyczny wzrost cen powodują m.in. te zapisy ustawy.

Po drugie, nałożenie na firmy zajmujące się odpadami dodatkowych wymagań - tj. monitoring, kaucje, rejestry - powoduje wzrost kosztów ich działalności nawet o 1 mln rocznie. Kolejnym powodem zwiększenia ceny wywozu odpadów jest wzrost opłaty za tzw. korzystanie ze środowiska.

Mimo że rząd PiS obiecywał, że nie będzie tych wzrostów, to one będą, i to bardzo drastyczne.

W związku z powyższym chciałabym zapytać pana ministra o to, w jaki sposób rząd zamierza rekompensować gminom wprowadzenie ustawy o odpadach, która w tak drastyczny sposób odbija się na mieszkańcach. Dziękuję bardzo. Pani poseł Krystyna Skowrońska, klub Koalicji Obywatelskiej. Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Różne dzisiaj oświadczenia były wygłaszane z tej mównicy. Powiem, że dla Polaków jedno z najważniejszych oświadczeń to oświadczenie pana posła Rafała Grupińskiego mówiące czy gratulujące naszej rodaczce Oldze Tokarczuk Literackiej Nagrody Nobla. Przyłączamy się jako klub Koalicji Obywatelskiej.

Działań nie ma. Moja koleżanka powiedziała o gospodarce odpadami, ważnej dla samorządów. Chciałabym się skupić na ważnej sprawie dla samorządów, ale również dla nas, tj. na finansowaniu oświaty i na brakującej subwencji dla samorządów. Z raportu, który przygotował Związek Miast Polskich, wynika, że łączna luka finansowania w oświacie liczona jako różnica między wydatkami a subwencją oświatową wynosi 27 mld zł. Luka ta szczególnie mocno zwiększyła się w latach 2017 i 2018, czyli w okresie przeprowadzania reformy w systemie edukacji. Jak wskazują samorządy, obecnie nie pokrywa się nawet kosztów wynagrodzeń, nie mówiąc o kosztach utrzymania szkół czy niezbędnych inwestycjach, których też przybywa ze względu na konieczność dostosowania klas do nowych warunków.

Otrzymałam pismo od jednego z samorządów.

Tych 10 mld zł budżet państwa w subwencji nie dał samorządowi. 30 października Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego omawiała kwestie związane z gwałtownym wzrostem wydatków samorządowych na oświatę będącym wynikiem reformy edukacji, a także podwyżek dla nauczycieli. W związku z tym tą drogą, bo nie ma projektu budżetu na rok 2020, a samorządy muszą podejmować decyzje o swoich budżetach, pytam pana premiera: Jak wyglądają dane dotyczące przydziału subwencji ogólnej na rok 2020 dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, ale i w województwie podkarpackim? Jakie działania zamierza podjąć rząd, jeżeli przewidziane kwoty środków finansowych przekazywane samorządom w subwencji oświatowej w 2020 r. okażą się tak znacząco niewystarczające? O tyle jest mniej inwestycji albo są wyższe podatki lub opłaty. Nie sprawdziła się gospodarka odpadami, a finansowanie samorządów.

Pan poseł Bartłomiej Dorywalski, klub Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! „Bezpieczne Świętokrzyskie” Bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności i jest gwarantem jego zachowania oraz szansą na doskonalenie. Bezpieczeństwo to jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Odznacza się brakiem ryzyka utraty czegoś dla człowieka szczególnie cennego: życia, zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr materialnych i dóbr niematerialnych. Człowiek, aby w pełni móc rozwijać swój potencjał i produktywnie funkcjonować w społeczeństwie, potrzebuje czuć się bezpiecznie. Spełnienie tego warunku pozwala mu na stabilizację i działalność dla dobra swojej rodziny i kraju. Województwo świętokrzyskie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom swoich mieszkańców, zainicjowało program „Bezpieczne Świętokrzyskie” Początkowo zakładano, że program będzie funkcjonował przez 5 lat. Sukces, jaki odniósł, a także entuzjazm, z jakim się spotkał, spowodowały, że trwa on do dnia dzisiejszego, a następstwem zdrowej, kreatywnej rywalizacji między powiatami województwa świętokrzyskiego jest nagroda „Koziołka” Idea wyróżniania powiatów, które szczególnie zaangażowały się w realizację celu mającego zapewnić mieszkańcom województwa świętokrzyskiego maksymalny poziom bezpieczeństwa, zrodziła się wśród kieleckich policjantów. Mając na uwadze to, że wizerunek Koziołka Matołka z Pacanowa budzi powszechną sympatię, postanowiono na bohatera statuetki wybrać postać owego koziołka.

Od tego czasu, to znaczy od 2000 r., jest on doroczną nagrodą za wkład w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców. Zamiarem ufundowania nagrody Koziołka było przede wszystkim wsparcie aktywności oraz promocja samorządów, w rejonie których poprzez działania osób fizycznych i prawnych doszło do zauważalnej poprawy stanu bezpieczeństwa obywatelskiego oraz zabezpieczenia majątku państwowego, komunalnego i prywatnego. Utrwalane postawy społeczne mają umacniać ład, porządek, obywatelską postawę i prawidłową reakcję na wydarzenia, które zaistnieją w najbliższym otoczeniu mieszkańca ziemi świętokrzyskiej. W ten sposób ukazane są dobre przykłady, osiągnięcia, a także możliwości działania na rzecz walki z przestępczością i patologią. Udział w programie „Bezpieczne świętokrzyskie”, a co za tym idzie rywalizacja między powiatami oswaja społeczeństwo z działaniami służb i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa obywateli i ochrony ich praw oraz majątków. Dla najlepszych, którzy swoją postawą i działaniami udowodnią, że zasługują na wyróżnienie prestiżową statuetką koziołka, zagwarantowane jest wsparcie finansowe na realizowane projekty związane z programem „Bezpieczne świętokrzyskie” Aby znaleźć się w gronie kandydatów do nagrody, powiaty województwa świętokrzyskiego muszą podjąć czynności daleko wykraczające poza ich zwykłe obowiązki na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Przy eliminacjach do nagrody dokonywana jest analiza działań takich, jak: wzrost poziomu bezpieczeństwa, zabezpieczenie majątku państwowego bądź prywatnego, przyczynienie się do upowszechnienia podstaw społecznej aktywności w zakresie bezpieczeństwa innych ludzi oraz ładu i spokoju publicznego. Początkowej oceny powiatów dokonuje zespół roboczy oddelegowany przez kapitułę nagrody Koziołka, składający się z przedstawicieli wojewody świętokrzyskiego, marszałka województwa świętokrzyskiego oraz świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Policji w Kielcach. Zespół ten co roku odwiedza poszczególne powiaty, które zgłosiły chęć uczestnictwa w konkursie, i na miejscu przygląda się realizowanym działaniom podnoszącym bezpieczeństwo w regionie. Zespół roboczy przy kapitule nagrody Koziołek po podsumowaniu sprawozdań z realizacji programu „Bezpieczne świętokrzyskie” kwalifikuje poszczególne powiaty do grona kandydatów na laureata corocznej edycji nagrody Koziołka. Ostateczną decyzję na posiedzeniu niejawnym podejmuje jednak kapituła Koziołka, w której skład wchodzą: wojewoda świętokrzyski, marszałek województwa świętokrzyskiego, świętokrzyski komendant wojewódzki Policji, prezes stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego. Zwycięzca oraz powiaty, które zajęły drugie i trzecie miejsce, otrzymują nagrodę rzeczową Koziołka oraz nagrody pieniężne, które należy przeznaczyć na realizację programu „Bezpieczne świętokrzyskie” Z osobistych względów pragnę nadmienić, że w tym roku nagroda Koziołka powędrowała do powiatu włoszczowskiego. Jest to szczególne wyróżnienie, biorąc pod uwagę, że odbyło się podczas jubileuszu 20. edycji nagrody, także było uhonorowaniem działań na rzecz bezpieczeństwa mających miejsce w 100-lecie odzyskania niepodległości. Powiat włoszczowski nie mógł lepiej uczcić rocznicy tak ważnej dla milionów Polaków, niż angażując się w 2018 r. podniesienie ich komfortu i bezpieczeństwa. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie osób i instytucji, które z wielkim poświęceniem realizowały program. Należy tutaj wymienić Komendę Powiatową Policji na czele z komendantem Mariuszem Przyborowskim, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej na czele z komendantem Krzysztofem Cioskiem, fundację Dzwonek „Jesteśmy blisko”, a także szereg indywidualnych osób, w tym wyróżnionego Marcina Sztukę. Nagroda Koziołka to wspaniała inicjatywa ze strony świętokrzyskiej policji. Refleksja nad programem „Bezpieczne świętokrzyskie”, a co za tym idzie nagrodą Koziołka, nie może być inna niż to, że praca zespołowa jest najważniejsza. Indywidualizm ceniony jest przez chwilę, nic nie przynosi najlepszych efektów niż praca razem.

Wysoka Izbo! W 2011 r. rządząca Warszawą Platforma sprzedała Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Ta miejska spółka była monopolistą na rynku warszawskim, jeżeli chodzi o dostarczanie ciepła do mieszkań. Spółka ta była właścicielem miejskiej sieci ciepłowniczej i posiadała ogromną liczbę patentów, ale także przynosiła miastu ogromne dochody.

Jak to się stało, że państwowej firmie z Francji opłacało się kupić Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, a miastu stołecznemu Warszawa nie opłacało się posiadać spółki, która była monopolistą na rynku warszawskim? Od tego czasu nastąpiło pogorszenie jakości świadczonych usług. Nowy właściciel zlikwidował dzielnicowe Zakłady Energetyki Cieplnej odpowiedzialne za usuwanie awarii i konserwację urządzeń. O braku odpowiedniej konserwacji może świadczyć ostatnia awaria magistrali, która odcięła kilka dzielnic Warszawy od dostaw ciepła. W przeciągu kilku lat nastąpiły znaczne podwyżki opłat za ciepło w Warszawie, chociaż Platforma Obywatelska w 2011 r. obiecywała, że się tak nie stanie. SPEC, czyli kura znosząca złote jaja, została sprzedana, a nowy właściciel sieci ciepłowniczej może bezkarnie łupić mieszkańców Warszawy. Miasto stołeczne Warszawa pozbawiło się dywidendy z posiadania SPEC-u.

Obecne roczne przychody tej spółki sięgają ponad 100 mln zł. Platforma w Warszawie, sprzedając Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej za relatywnie niską cenę, doprowadziła do tego, że miejski monopolista trafił w ręce zagranicznej państwowej spółki, która podwyższyła ceny dostarczania ciepła, a jednocześnie obniżyła standard usług. Czy to jest działanie dla dobra mieszkańców? Dziękuję bardzo. Na tym zakończyliśmy oświadczenia poselskie.